Trybunału Sprawiedliwości. Wniosek do dzisiaj nie został wycofany. Komisja Europejska przyłącza się do skargi po stronie czeskiej, a polski rząd dalej nic nie robi. Ja rozumiem, że macie kłopot, bo zajmujecie się sprawdzaniem, co mieliście na skrzynkach prywatnych, jakie niejawne informacje przesyłaliście sobie na prywatne skrzynki, ale Polska jest dzisiaj w niebezpieczeństwie. Możemy płacić 5 mln euro kary dziennie za waszą nieodpowiedzialność. Wysoka Izba jako organ kontrolny rządu powinna wysłuchać informacji na ten temat.

Dlatego nie będziemy o tym dyskutować przedwcześnie. Ale ponieważ złożył pan wniosek o przerwę, ten wniosek przegłosujemy. W związku z tym, że został zgłoszony wniosek formalny o przerwę, poddam ten wniosek pod głosowanie. Kto z pań i panów posłów jest za zarządzeniem przerwy w obradach, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Wniosek nie przeszedł. Proszę bardzo, pan poseł Robert Obaz, Lewica - wniosek formalny. Wysoka Izbo! 30 tys. ludzi, którzy są związani z Bogatynią, z kopalnią, czekało dzisiaj na informację rządu. Centrale związkowe, pani Stasia, pani Zosia, pan Michał, wszyscy czekali, żeby dowiedzieć się, co tak naprawdę zrobił polski rząd. A zrobił kompletnie nic. Nic się nie wydarzyło. Do dzisiaj pracownicy Kopalni Węgla Brunatnego Turów w Bogatyni oraz pracownicy elektrowni, która także znajduje się obok tego kompleksu, nie wiedzą, co dalej. Wszystkie firmy współpracujące zarówno z kopalnią, jak i z elektrownią są zupełnie rozstrojone, ponieważ nie wiedzą, czy za miesiąc, dwa, rok czy półtora roku będą miały pracę.

Proszę bardzo.

Panie i Panowie Posłowie! Mieszkańcy Turowa mają prawo wiedzieć, jaka przyszłość ich czeka. Orzeczenie nie jest dobre dla nikogo. Naraża nas na wysokie kary, pracowników Turowa i ich rodziny naraża na utratę pracy, pieniędzy i godności. Może podważyć bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju. Wykluczyliście górników węgla brunatnego z systemu i z jakichkolwiek umów. Nie tworzycie żadnych programów kompensacyjnych, żadnych programów transformacyjnych. Straszyliście dziką transformacją, a tak naprawę dziś sami ją inicjujecie.

Poddam ten wniosek pod głosowanie. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za odroczeniem posiedzenia, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Proszę bardzo, pan poseł Jacek Protasiewicz, Koalicja Polska. Wysoki Sejmie! Pani marszałek Gosiewska zainspirowała mnie, żeby poprosić o powstanie i uczczenie minutą ciszy pamięci Witolda Jerzego Kieżuna, bohaterskiego powstańca warszawskiego odznaczonego za swoje czyny w trakcie tej nierównej walki Orderem Virtuti Militari przez gen. Okulickiego, skazanego na łagry sowieckie, wybitnego profesora ekonomii, prawnika, człowieka niezwykłego.

Teraz przejdę do wniosku formalnego. W imieniu Koalicji Polskiej chciałbym zaprotestować przeciwko zdjęciu na posiedzeniu Konwentu Seniorów z porządku obrad informacji o Turowie. To, co rząd wyprawia w sprawie Turowa, to jest dosłownie czeski film. Być może nie wszyscy pamiętają, co to znaczy, a zwłaszcza młodsze pokolenie. To było określenie na czeskie firmy awangardowe z lat. W tej sprawie też nikt nie wie, o co chodzi. Tam był doktor Strosmajer, który mówił: Gdyby głupota umiała latać, to unosiłaby się pani jak gołębica. Otóż gdyby głupota umiała latać, to w tej sprawie rząd powinien się wzbijać całymi stadami, tabunami i latać pod niebiosa. To co wyczyniacie z tymi negocjacjami, jak informujecie, a w zasadzie dezinformujecie, Polaków, górników, hutników, elektryków, to jest naprawdę przejaw bezdennej głupoty. Dziękuję, panie pośle. Na drugi raz nie warto kłamać ani mnie oszukiwać, panie pośle, trzeba było powiedzieć, o co panu chodzi, naprawdę.

Po pierwsze, to są kłamstwa, że rząd nic nie robi. W tej sprawie odbyły się dwa posiedzenia Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych. Ci, którzy w nich uczestniczyli, usłyszeli, jaka jest sytuacja.

To są fakty niezbite. Gdybyście państwo się tym zainteresowali, tobyście wiedzieli. że Czesi trochę naciągają sytuację. Ale skandalem jest to, że taka mentalność zdrajców, która dominuje na opozycji. powoduje, że stajecie. po stronie innego państwa w sporze z Polską.

Szanowni Państwo! Nie potrzebują tych polityków Platformy i Lewicy, którzy mówią, żeby zamykać polskie górnictwo, którzy cieszą się z tego, że Komisja Europejska, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nas atakują. Szanowni państwo, to, co powiedział pan Marek Suski, to jest prawda. Wy nie wiecie, co to jest lojalność wobec Polski. Nie wiecie. Wy się cieszycie z tego, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nas atakuje. Chcecie pomóc górnikom? Chcecie pomóc Turowowi? Dziękuję bardzo, panie pośle. Proszę nie. Panie przewodniczący, proszę bardzo, ma pan minutę. Pani Marszałek! Proszę o stanowczą reakcję w takiej sytuacji, kiedy ze strony pana posła Marka Suskiego w kierunku opozycji padają słowa o mentalności zdrajców. To jest absolutny skandal, że takie słowa padają. Wnoszę oficjalnie o to. żeby pan poseł Suski był wykluczony z obrad. I proszę o stanowczą reakcję pani marszałek wtedy, kiedy takie słowa padają w tej Izbie. Jeżeli my sobie pozwolimy w polskim Sejmie, żeby słowa o zdradzie padały w taki prosty sposób, to przypomnę, że pan premier Morawiecki powiedział, że sprawa Turowa jest załatwiona. publicznie kłamał w tej sprawie, w sprawie negocjacji z Czechami. To jest wasza odpowiedzialność, wasza wina. Dzisiaj próbujecie od tego uciec. A pan nie powinien na tej sali dzisiaj zabierać głosu. Bo prawda jest taka, że to jest. Zamieniliście w propagandę prawdziwe działanie i prawdziwą dyplomację. Po prostu weźcie się do roboty.

Proszę państwa, była mowa o mentalności. Ja słyszałam naprawdę znacznie gorsze określenia z państwa strony na tej sali.

Wysoka Izbo! Liczę na to, że to będzie oznaczało, że wyłączony zostanie system głosowania tabletowego, mam nadzieję. Szacunek, pani marszałek, dziękuję bardzo za te decyzje. Ze względu na temperaturę sporu, która tutaj się pojawiła, wnioski formalne odrzucane w sprawie Turowa i jeszcze kwestię rzecznika praw obywatelskich oraz nagle zwołane posiedzenie dotyczące cyberbezpieczeństwa, szanowni państwo, pani marszałek, Wysoka Izbo, zgłaszam wniosek o zamknięcie obrad. I wtedy pani marszałek zwołuje nowe posiedzenie, ale nowe posiedzenie - zgodnie z tym, co było powiedziane na posiedzeniu Konwentu Seniorów - już w pełnym składzie. Dla niektórych będzie to bolesny powrót po roku nieobecności na tej sali, ale mam nadzieję, że jakoś to przeżyją, w końcu od tego tutaj są. No i życzę państwu wszystkim zdjęcia maseczek i powrotu do normalności. Tak że wniosek o zamknięcie obrad.

Pomijam to. Pan sobie zdaje sprawę z tego, że w tej chwili nie ma możliwości, żeby wszyscy, którzy są poza salą, nagle przyjechali. Doskonale pan o tym wie. Proszę państwa, były problemy z dojazdem na jutro na godz. 9 rano, więc myślę, że. Proszę państwa, padł wniosek o zamknięcie obrad. Poddam ten wniosek pod głosowanie. Kto z pań i panów posłów jest za zamknięciem obrad, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 1. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (druki nr 1243 i 1254) Proszę panią poseł Annę Paluch o przedstawienie sprawozdania komisji. Dziękuję bardzo. Wysoka Izbo! W imieniu Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa przedstawiam sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Projekt zawarty w druku nr 1243 został w dniu 4 czerwca skierowany do komisji. Projekt jest krótki, obejmuje zaledwie trzy artykuły.

Usuwane obecną nowelizacją przepisy zostały wprowadzone ustawą z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw i miały na celu zachowanie ciągłości prowadzenia wydobycia węgla kamiennego, węgla brunatnego i siarki rodzimej wydobywanej metodą otworową bez konieczności uprzedniego uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Przepisy wówczas ustanowione dozwalały, aby w przypadku wydłużania terminu obowiązywania koncesji na wydobycie węgla kamiennego ze złoża w ramach prowadzenia działalności w granicach obszaru górniczego wyznaczonego obowiązującą koncesją nie był stosowany wymóg uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Podobnie dla węgla kamiennego było możliwe wydłużenie koncesji do 6 lat, podobnie dla trzeciej wymienionej kopaliny. Wydłużenie było jednorazowe. Wprowadzenie tych zmian było w oczywisty sposób uzasadnione racjonalną gospodarką złożami kopalin, wykorzystaniem całości dostępnych zasobów oraz zachowaniem ciągłości wydobycia. Wysoka Izbo! Obecnie brak jest uzasadnienia dla dalszego obowiązywania tych przepisów.

Art. 2 projektu zawiera przepis przejściowy stanowiący, że do wszczętych i niezakończonych postępowań administracyjnych w sprawie wydłużenia terminu obowiązywania koncesji, tych, o których mowa w art. 72 ust. 2 pkt 2 lit. j-l ustawy, stosuje się przepisy nowe, tzn. do wszystkich wniosków o wydłużenie koncesji na wydobycie przedmiotowych kopalin będzie konieczne uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Art. 3 z kolei stanowi, że ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania. Wysoka Izbo! Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa przeprowadziła pierwsze czytanie tego projektu w dniu 11 czerwca, po czym przeprowadziła nad nim szczegółowe prace.

W imieniu Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa proszę o uchwalenie projektu ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko bez poprawek, tzn. w wersji z przedłożenia rządowego. Dziękuję bardzo, pani poseł. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół. Jako pierwszy głos zabierze pan poseł Jan Duda, Prawo i Sprawiedliwość.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie i Panowie Posłowie! Po wystąpieniu posła sprawozdawcy niewiele zostało do powiedzenia, ale postaram się przedstawić stanowisko klubu parlamentarnego w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zawartego w druku nr 1243.

Uchylone przepisy dotyczą zwolnienia z obowiązku uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczących jednorazowego przedłużenia koncesji na wydobywanie węgla kamiennego, węgla brunatnego i siarki. Art. 2 to przepisy przejściowe, a art. 3 - czas wejścia w życie ustawy.

Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość w pełni podziela argumentację rządu i będzie głosował za przyjęciem przedstawionego w druku nr 1243 projektu ustawy. Bardzo proszę, pani poseł Urszula Zielińska, Koalicja Obywatelska. Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Zieloni odnośnie do projektu ustawy zawartego w druku nr 1243. Debatujemy nad krótką nowelizacją tzw. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz - uwaga - o ocenach oddziaływania na środowisko, a konkretniej w tym przypadku o braku tych ocen.

Te niezgodne z prawem przepisy pozwalały na jednokrotne przedłużenie koncesji wydobywczej na węgiel kamienny, brunatny, siarkę, węglowodory bez konieczności przeprowadzenia procedury środowiskowej lub procedury zastępczej przewidzianej dyrektywą. W tym miejscu należy zapytać: Ale w jaki sposób niezgodny z prawem europejskim zapis znalazł się w polskiej ustawie i kto za to odpowiada? Otóż przepisy te wprowadzili w życie w czerwcu 2018 r. główny geolog kraju pan Mariusz Orion Jędrysek pod nadzorem ministra środowiska pana Henryka Kowalczyka w rządzie premiera Mateusza Morawieckiego. Na podstawie tych niezgodnych z prawem przepisów inwestor mógł bez problemu przedłużyć sobie możliwość wydobycia np. węgla kamiennego nawet o 40 lat, bez konieczności przedstawienia wpływu tego wydobycia na zdrowie pracowników i mieszkańców, na bezpieczeństwo ludzi, na zanieczyszczenie wody, gleby, powietrza, na degradację przyrody. Po wprowadzeniu tych niezgodnych z prawem przepisów minister zdrowia w rekordowym tempie przedłużył 20 koncesji wydobywczych, niektóre nawet o 40 lat. Wszystkie bez procedury i pozwolenia środowiskowego. To pokazuje gigantyczną skalę naruszeń względem ludzi i środowiska, która odbywa się w naszym kraju. To oznacza, że mieszkańcy wielu terenów wydobywczych, m.in. rejonów kopalni: Silesia, Budryk, Sośnica, Ruda, Knurów-Szczygłowice i wielu innych, mają znikome, jeżeli jakiekolwiek, informacje o prawdziwym wpływie wydobycia węgla, siarki, węglowodorów na ich zdrowie, na jakość wody, na ryzyko zapadania się terenu, na którym mieszkają i budują domy, na poziom hałasu, na jakość powietrza i wiele innych czynników. Mają też bardzo ograniczone możliwości zaskarżenia do sądu tego, co dzieje się często dosłownie pod powierzchnią ich domów.

Okazały się mniej ważne niż interesy rządu i wielkich spółek. Te procedury są dla inwestorów zbyt skomplikowane - argumentował minister Orion Jędrysek, uzasadniając ustawę w 2018 r. Dziś ten sam rząd w pośpiechu naprawia wyłom w prawie, który sam utworzył. Dlaczego? Bo jak sam przyznaje, nie ma już potrzeby. Rząd wydał już wszystkie koncesje, które chciał wydać, choćby z naruszeniem prawa. Rząd wie też, że naruszył dyrektywę, i słusznie boi się, że Komisja Europejska złoży przeciwko Polsce kolejny już pozew do Trybunału Sprawiedliwości. Jako Klub Koalicji Obywatelskiej będziemy oczywiście głosować za tą ustawą. Poprawimy też niedopatrzenie, zapis, który pozostawia w ustawie możliwość przedłużenia koncesji na złoża węglowodorów, znów bez pozwolenia środowiskowego. Niestety szkody już uczynione tą ustawą nie zostaną naprawione choćby najlepszą poprawką. Żeby je naprawić, potrzebujemy planu sprawiedliwej transformacji, inwestycji tworzących czyste, nowoczesne źródła energii i realne miejsca pracy w regionach górniczych, stabilnego miksu czystej energii produkowanej tutaj, w Polsce, nieimportowanej z Rosji, nieimportowanej ze Stanów Zjednoczonych, z krajów nordyckich - produkowanej tutaj, w Polsce.

Dziękuję bardzo, pani poseł. Bardzo proszę, pani poseł Anita Sowińska, Lewica. Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko klubu parlamentarnego Lewicy odnośnie do projektu ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 2 miesiące temu prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację tej właśnie ustawy. Powodem nowelizacji była możliwość wszczęcia przez Komisję Europejską procedury naruszenia prawa unijnego. Wtedy rząd przekonywał nas, że ta ustawa spełnia wymogi dyrektywy EIA, pomimo że strona społeczna i opozycja wskazywały, że tak nie jest. W lutym i marcu zgłosiliśmy do tej ustawy kilkanaście merytorycznych poprawek, które zostały odrzucone. Piszecie na kolanie, zmieniacie jeden artykuł, który pozwalał na przedłużenie koncesji na wydobycie węgla bez decyzji środowiskowej. Polki i Polacy są bezbronni w starciu z państwem i grupami interesu. Tą ustawą pozbawiliście ich prawa do odwołania się od złych decyzji środowiskowych, inwestycyjnych. Ludzie byli pozbawiani wody, czystego powietrza. Rolnicy ponosili straty z tytułu niższych plonów i nie dostawali za to rekompensaty.

Na posiedzeniu komisji ochrony środowiska, podczas pierwszego czytania ustawy zapytałam pana ministra, jakie jest ryzyko, że Polki i Polacy zaczną dochodzić swoich praw w sądach, tak samo jak dochodzą prawa Czesi. Nie uzyskałam odpowiedzi, dlatego zadaję to pytanie drugi raz. Na posiedzeniu komisji pytałam również o cel tej ustawy i także nie uzyskałam jasnej odpowiedzi. Naprawa tego przepisu nic nie zmienia w stanie faktycznym, ponieważ nowe kopalnie już się otworzyły, a nowych już nie będzie, zgodnie z polityką energetyczną.

To, co robicie, to są tylko pozorowane działania. Nie wystarczy zmienić jednego artykułu, bo do zmiany jest cała ustawa. Ta ustawa nadal odbiera obywatelkom i obywatelom prawo do współdecydowania i odwoływania się od złych decyzji inwestycyjnych. Ludzie nadal mają bardzo ograniczone prawo do informacji. Tę ustawę trzeba zmienić, szczególnie że w planach są potężne inwestycje wynikające z Krajowego Planu Odbudowy. Powinniśmy inwestować, ale trzeba to robić z głową. Przykładowo: aby wybudować zakład, fabrykę samochodów elektrycznych nie trzeba wycinać kilkudziesięciu hektarów lasu, można je wybudować na terenie zdegradowanym, poddawszy go rekultywacji, z korzyścią dla całego społeczeństwa i dla środowiska.

Zamiast bezmyślnie wycinać i niszczyć można naprawiać, pielęgnować i budować z rozumem. Taka jest rola polityków i polityczek: służenie społeczeństwu i przyrodzie. Wiem, że to się wam nie mieści w głowie, ale my nie pozwolimy, abyście zniszczyli nasz dom. Ta ustawa jest bublem prawnym, dlatego składamy dwie merytoryczne poprawki. Dziękuję, pani poseł. Bardzo proszę, pan poseł Andrzej Grzyb, Koalicja Polska. Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Jest to niewielka, jak się wydaje, zmiana, bo dotyczy skreślenia tylko kilku liter, od j do l w art. 72 ust. 2 pkt 2, ale to jest właśnie ten incydentalny przepis, który został wprowadzony w 2018 r.

Warto przypomnieć przy okazji tej dyskusji, że art. 74 ust. 3 konstytucji mówi, że każdy - jeszcze raz to podkreślam: każdy - posiada prawo do informacji o stanie ochrony środowiska. Ten sam przepis jest również w ustawie zmienianej dzisiaj poprzez skreślenie akurat niektórych zapisów w art. 72 ust. 2 pkt 2.

Myślę, że to jest pewna nauka.

To jest również zobowiązanie poprzednich rządów. Ja tego w żaden sposób nie próbuję kamuflować. Stąd też ta nowela, dopiero co podpisana przez prezydenta, która wprowadza zasady udziału społeczeństwa obywatelskiego, w tym organizacji pozarządowych, w sprawach dotyczących ochrony środowiska, ale również możliwości postępowania przed sądami. To również ta zmiana, która jest na wniosek rządu. Wydaje mi się, że ona ma też pewien kontekst odnoszący się do tego, co było przedmiotem dzisiejszej porannej dyskusji, dotyczącej również Turoszowa.

Zresztą eksperci, chociażby z tego portalu, tak się wypowiadają. Konkludując: popieramy tę zmianę (Dzwonek) jako klub Koalicji Polskiej. Uważamy, że ona jest potrzebna i zasadna.

Panie Przewodniczący Komitetu do spraw Bezpieczeństwa Kaczyński! Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Na podstawie złego prawa przez 3 lata wydaliście 20 koncesji na przedłużenie funkcjonowania kopalń bez potrzeby wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Dwa razy dla Turowa, a poza tym dla: KWK Silesia, Budryk, Sośnica, Ruda, Knurów, Szczygłowice, Makoszowy, Wujek, Staszic, Mysłowice-Wesoła, Piast-Ziemowit, Bolesław Śmiały. Oznacza to, że kopalnie, które powstawały w 70., 80. latach, nigdy nie przechodziły procedury oceny oddziaływania na środowisko. Nie wiemy, ile osób przez te kopalnie choruje na raka, choroby płuc, a może ma problemy z wodą i jej jakością. I jak te kopalnie wpływają na zanieczyszczenie środowiska, na faunę, florę, jaki generują poziom hałasu. Jakie będą kary za kolejne koncesje? Nawet jeżeli akurat w pobliżu jakiejś kopalni nie mieszkają Czesi, to przecież pozywać Polskę mogą też Polki i Polacy. 5 mln euro dziennie za Turów niczego was nie nauczyło? Panie ministrze, pytam wprost: Do jakich kar doprowadzą koncesje z pominięciem decyzji środowiskowych? Czy ktoś to w rządzie policzył? Czy są przeznaczone na to środki w budżecie, a jeżeli tak, to jakie? Dziękuję bardzo, pani poseł. Pani poseł Beata Maciejewska, Lewica. Wysoka Izbo! Polityka PiS-u wobec środowiska jest jedna: ciąć, rżnąć i truć.

Domaga się wstrzymania tej decyzji.

Tak dzisiaj działa minister, który powinien bronić środowiska.

Lewica mówi jasno: nie zgadzamy się na to. Bardzo proszę, pan poseł Michał Urbaniak, Konfederacja. Nie ma pana posła.

Wysoka Izbo!

Nie robicie nic.

Chciałbym się dowiedzieć, na jakim etapie jest ten plan. To jest jedno pytanie. Czy wybraliście technologię? To jest drugie pytanie.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! PiS usunął z dzisiejszego porządku obrad informację rządu na temat Turowa. Boicie się.

Nie macie nic innego poza tym, że Komisja Europejska dołączyła do skargi Czechów przeciwko Polsce.

Kiedy spojrzycie prawdzie w oczy? Kiedy przedstawicie ambitny plan odejścia od węgla i sprawiedliwej transformacji do 2030 r. nie tylko dla rejonu Turoszowa, lecz także dla całej Polski? Dziękuję bardzo. Pan poseł Grzegorz Rusiecki, Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo!

Mamy zobowiązania wobec kolejnych pokoleń. Tymczasem ochrona środowiska w wydaniu realizowanym przez PiS to traktowanie środowiska w sposób przedmiotowy. Przyjęto ustawę, wycięto w całym kraju bez żadnego trybu. Dzisiaj, proszę państwa, robicie dokładnie to samo. Przyjęliście ustawę w 2018 r. Bardzo proszę, pani poseł Joanna Fabisiak, Koalicja Obywatelska.

Wysoka Izbo! W 2011 r. Unia Europejska przegłosowała dyrektywę chroniącą środowisko. W 2018 r. rząd przepchnął ustawę pozwalającą na przedłużenie koncesji wydobywczych nawet o 40 lat dla 20 kopalni. Dzisiaj poprawia tę ustawę, ale poprawia tylko do przodu. Co stanie się z tymi kopalniami?

Boryka się z problemami finansowymi - brak pieniędzy dla pacjentów jest przecież rzeczą normalną - a jednocześnie wyraża zgodę, chyba cyniczną zgodę, na to (Dzwonek), żeby Bo koncesje wydane na 40 lat to naprawdę trucie ludzi przez najbliższe dziesiątki lat, przez najbliższe dekady. Bardzo proszę, pan poseł Tomasz Piotr Nowak, Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo! Rząd ma wyraźny problem z tym chodzeniem na skróty. Chodzicie na skróty w dyplomacji europejskiej, chodzicie na skróty w gospodarce, staracie się stworzyć politykę faktów dokonanych i to jest taki przykład tworzenia polityki faktów dokonanych, ale przy okazji wywracają się takie projekty jak właśnie Turów. Czy w Turowie nie mieliśmy do czynienia z działaniem dotyczącym przyspieszenia wydania koncesji, która spowodowała ten kryzys, który mamy obecnie? Czy konsultacje transgraniczne w ocenie oddziaływania na środowisko nie powinny być przeprowadzane dłużej i skuteczniej, tak żeby nie było wątpliwości przy wydaniu tej koncesji i żeby nie skutkowała ona kolejnym kryzysem? Obawiamy się, że tych kryzysów może być o wiele więcej. Wskazanie na elektrownię atomową też nie jest przypadkowe (Dzwonek), ale także na offshore, na wiatraki na morzu, bo tutaj również oddziaływanie na środowisko może być przemożne, a nie mamy raportu, czy będzie postępowanie transgraniczne i czy ono jest wymagane. Dziękuję bardzo, panie pośle. Pan poseł Mirosław Suchoń, Polska 2050.

Bardzo dziękuję. Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Wydaje się, że oczywisty jest fakt, że takie uregulowanie, które miało miejsce, które dzisiaj państwo zmieniają, spowodowało, że po pierwsze, nie trzeba było podnosić kosztów tych wszystkich ocen oddziaływania na środowisko na społeczeństwo, które funkcjonuje w obrębie inwestycji, a po drugie, nie zbadano także dokładnego wpływu i kosztów, które są z tym związane. W związku z tym mamy dwa efekty. I pytanie: Ile zaoszczędzono z powodu takiego uregulowania przepisów, które dzisiaj zmieniamy?

Natomiast pytanie, panie ministrze: O ile odsunęli państwo w sposób oczywiście szkodliwy tę transformację energetyczną? Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani poseł Agnieszka Hanajczyk, Koalicja Obywatelska. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Procedowana ustawa jest kolejną zmianą, która miała miejsce niedawno. Tło jest dzisiaj bardziej wyraźne, bo po pierwsze, w tle jest Turów, są kopalnie węgla, którym wcześniej rząd bardzo szybko przyznał koncesje bez odpowiedniego zbadania, jaki to będzie miało wpływ na życie mieszkańców, i sama bardzo istotna ocena środowiska. Ustawa, która - jak się wydaje - jest potrzebna, jest niewątpliwie odpowiedzią na konflikt z Czechami i w sposób dla mnie oczywisty maskowaniem nieodpowiedzialnych wcześniejszych działań rządu. Natomiast moje pytanie dotyczy dwóch spraw. Mianowicie: Ile koncesji na wydobycie węglowodorów jest obecnie w procedurze przyznawania?

Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani poseł Małgorzata Niemczyk, Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo!

Chodzi o to, żeby kochać Polskę, kochać środowisko, kochać ludzi, którzy mieszkają, i wiedzieć, jak co oddziałuje. Nie ponosicie kosztów w związku z przebadaniem tego oddziaływania, więc nawet nie wiecie, jakie koszty będziecie musieli później ponosić, aby usunąć skutki waszych decyzji. Czy planujecie w ogóle naprawić te swoje błędy kiedykolwiek? Jeżeli są teraz te koncesje powydawane na 40 lat czy w ciągu tych 40 (Dzwonek) lat, to najlepiej jeszcze w tej kadencji zbadajcie, jakie są tego skutki. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan poseł Janusz Kowalski, Prawo i Sprawiedliwość. Droga Opozycjo! Jednej rzeczy kompletnie nie rozumiecie. Kwestia dotycząca koncesji to jest kwestia dotycząca suwerenności, suwerenności energetycznej i suwerenności dotyczącej bezpieczeństwa energetycznego Polski. Zdolność polskiego państwa do tego, aby wydawać koncesje i bronić przed zewnętrznymi atakami czy to czeskimi, niemieckimi czy brukselskimi, to jest zdolność do zachowania władztwa nad polskimi zasobami energetycznymi. Bez polskiego węgla nie ma mowy o tym, żebyśmy produkowali energię elektryczną. Dlatego bronię suwerenności energetycznej, bronię polskiego węgla i mam nadzieję, że również koncesja na złoże Złoczew zostanie wydana po to, żeby zabezpieczyć elektrownię Bełchatów. Nie ma co uzależniać się od importu energii elektrycznej z Niemiec, ze Skandynawii, z Czech. Nie ma co stawiać na niestabilne źródła energii. Polsce bezpieczeństwo energetyczne. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani poseł Magdalena Łośko, Koalicja Obywatelska. Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Jeziora Pojezierza Gnieźnieńskiego znajdujące się na terenie Wielkopolski i Kujaw wskutek funkcjonowania odkrywek węgla od lat ulegają stopniowej degradacji. Przede wszystkim należy przywrócić równowagę hydrologiczną, która została naruszona wskutek funkcjonowania tych odkrywek. Miejscowości dotychczas turystyczne zamierają, a kwestia rekultywacji jest o wiele szerszym problemem, aniżeli przedstawiciele ministerstwa zobrazowali to na posiedzeniu komisji. Pani poseł Krystyna Skowrońska, Koalicja Obywatelska. Szanowna Pani Marszałek! Panie i Panowie Posłowie!

Chcę powiedzieć: nie mówicie nic o bezpieczeństwie energetycznym i nie mówicie nic o bezpieczeństwie zdrowotnym. 100 tys. zgonów nadmiarowych z tytułu COVID. Chciałam zapytać pana ministra: Ile było zgonów Polaków w związku z zanieczyszczeniem środowiska?

Powiedzcie młodemu pokoleniu i powiedzcie nam, że będziemy żyć i że nie będziecie tworzyć iluzorycznych ustaw, które będą wpływały na pogorszenie stanu środowiska. Dziękuję. Dziękuję bardzo, pani poseł. Na pytania odpowie podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska pan Piotr Dziadzio. Bardzo proszę.

Pani Marszałek! Szanowni Państwo! Wysoka Izbo!

Szanowni Państwo!

Szanowni państwo, z tego wynika, że bardzo dobrze rozumieliście i rozumiecie potrzeby Rzeczypospolitej i w związku z tym takie były rezultaty państwa głosowania. Niemniej jednak większość zarzutów, które tutaj padły, dotyczy Turowa.

Szanowni państwo, nie uprawiajmy nieprawdy. Mówmy tak, jak wygląda rzeczywistość. Większość pytań dotyczyła odpowiedzialności za energetykę, odpowiedzialności za czyste powietrze, za klimat. Szanowni państwo, w polityce energetycznej państwa do 2040 r. większość zagadnień, o których mówimy czy o których państwo mówiliście, jest uregulowana, jest wskazana. To, jaka jest linia bezpieczeństwa energetycznego i całej transformacji energetycznej, jest bardzo dobrze przedstawione i wykazane. Dbamy tam przede wszystkim o odnawialne źródła energii. Żebyśmy jednak mogli mieć odnawialne źródła energii, o czym państwo dyskutujecie na co dzień z sobą, musimy mieć kontynuację naszej działalności i bezpieczeństwa energetycznego, które są oparte w tej chwili na węglu kamiennym, węglu brunatnym. Żeby sprawiedliwie przeprowadzić tę transformację, musimy stopniowo odchodzić od jednych źródeł i zastępować je innymi źródłami, tak żebyśmy mogli uzyskać neutralność klimatyczną. Do tego dążymy.

Szanowni Państwo!

Szanowni państwo, działamy w interesie Rzeczypospolitej. Nie mamy żadnych ukrytych interesów, które tutaj państwo próbujecie nam zasugerować (Dzwonek) czy przedstawić. To jest chyba wyjaśnienie, na które państwo oczekiwaliście. Proszę kończyć, panie ministrze.

Dziękuję bardzo, panie ministrze. Dziękuję bardzo. Wysoka Izbo! Słyszeliśmy w wystąpieniach klubowych kategoryczne stwierdzenia o niezgodności z prawem europejskim. Przypominam, że Komisja Europejska pisze o potencjalnej niezgodności, o zagrożeniu potencjalną niezgodnością, więc oszczędźcie sobie tych kategorycznych sformułowań. Słyszeliśmy o prawie mieszkańców do życia w czystym środowisku. Ale czasami to prawo pozostaje w kolizji z prawem do pracy, prawem do możliwości uzyskania środków do życia, prawem do tego, żeby jeśli się 40 lat pracowało w jakimś zakładzie pracy, jeszcze te 10 lat dopracować, a nie martwić się, co się stanie po zamknięciu zakładu.

Tą grupą interesów są Polacy korzystający ze źródeł energii, z tego, że mamy stabilny system energetyczny, który w części jest oparty na węglu.

To są inne sprawy niż te w projekcie, który w tej chwili omawiamy. I jeszcze raz to podkreślę, chociaż już to w swoim wstępnym wystąpieniu powiedziałam: chodzi o racjonalną gospodarkę złożem i działanie w ramach obowiązujących koncesji. Powiedziałam to wyraźnie: to nie są jakieś nowe sytuacje. Jeżeli się kilkadziesiąt lat eksploatowało złoże, to zdrowy rozsądek wymaga, żeby je wyeksploatować do końca, a potem zamknąć wydobycie.

A więc myślę, że dobrze by było jednakowo obdarzyć uwagą wszystkie te przedsięwzięcia, o których mówimy.

Usłyszałam deklaracje, przynajmniej z niektórych klubów, poparcia przedmiotowego projektu ustawy, za które dziękuję.

Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych w sprawie trzech poselskich projektów uchwał, których tytuły wymieniła pani marszałek. Jest to bardzo nietypowa sytuacja.

Wzywamy też Stany Zjednoczone Ameryki jako naszego sojusznika w NATO do utrzymania oraz rozszerzenia sankcji wymierzonych w podmioty uczestniczące w budowie gazociągu. Unia Europejska i NATO od 30 lat podejmowały wielorakie wysiłki zmierzające do ułożenia stosunków z Rosją. Wszystkie one zostały potraktowane przez Rosję jako przygotowanie gruntu dla imperialnej ekspansji, a przyświecające im zasady prawa międzynarodowego zostały przez nią brutalnie podeptane w aktach zbrojnej agresji na Gruzję w 2008 r. i na Ukrainę w okresie od 2014 r., których skutki w postaci nielegalnych okupacji części ich terytoriów, podobnie jak nielegalnej secesji Naddniestrza oderwanego od Mołdawii, nadal trwają. Eksport węglowodorów jest źródłem finansowania rosyjskich zbrojeń i jako taki jest istotnym instrumentem agresywnej polityki Rosji względem nie tylko państw ościennych, ale również innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Nord Stream 2 ma na celu wyłącznie zmianę tras dostaw, a nie ich dywersyfikację. Wyrażamy przekonanie, że akceptacja kontynuacji projektu dotyczącego Nord Stream 2 w opisanych okolicznościach jest przyzwoleniem na prowadzenie przez Federację Rosyjską polityki opartej na gwałceniu międzynarodowych standardów praw człowieka, naruszaniu integralności państw ościennych i wywieraniu presji na państwa Unii Europejskiej i NATO. W Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej w Komisji Spraw Zagranicznych nie było najmniejszych wątpliwości, że ostry język, jaki zawiera ten projekt uchwały, jest właściwą odpowiedzią na działania rządów Republiki Federalnej Niemiec i Federacji Rosyjskiej. Dziękuję bardzo, panie pośle. Jako pierwszy głos zabierze pan poseł Janusz Kowalski, Prawo i Sprawiedliwość.

Rzeczywiście jest tak, że w sprawie uchwały dotyczącej Nord Stream 2, a więc projektu, który dzieli Unię Europejską, dzieli Europę, dzieli Europę Środkowo-Wschodnią, wszyscy mówimy jednym głosem. Jest to bardzo ważne, że w Komisji Spraw Zagranicznych ten projekt został przyjęty przez aklamację, a więc adresaci naszej uchwały, uchwały polskiego Sejmu, wiedzą, że sprawa ta jednoczy wszystkich Polaków ponad podziałami politycznymi.

Kwestia przemocy ze strony państwa rosyjskiego i łamania praw międzynarodowych pokazuje, że musi być jasno powiedziane: stop.

Uderzy też w bezpieczeństwo Polski, uderzy w bezpieczeństwo państw bałtyckich, będzie zachętą dla Rosji Władimira Putina do dalszej agresji na Ukrainę. Dzisiejsza uchwała, dzisiejszy projekt uchwały anty-Nord-Stream w istocie jest wezwaniem do pokoju w Europie, jest próbą przewidzenia tego scenariusza, który może się wydarzyć - oby się nie wydarzył. Ale ten ważny, ponadpolityczny głos, głos ponad bieżącymi kwestiami politycznymi wszystkich ugrupowań polskiego Sejmu jest jasny dla całej opinii międzynarodowej, za co bardzo serdecznie wszystkim chcę podziękować, ponieważ my jako Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości w sposób absolutnie naturalny nawiązujemy do dziedzictwa śp. prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, który przecież w roku 2006 zapoczątkował cały projekt dywersyfikacji dostaw nośników energii do Polski, czyli projekt budowy gazoportu i projekt budowy Baltic Pipe, i który w 2008 r. wystąpił w obronie integralności i suwerenności Gruzji. W związku z tym, szanowni państwo, przyjmijmy ten projekt ponad podziałami politycznymi, za co bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę, pan poseł Paweł Kowal, Koalicja Obywatelska. Wielce Szanowna Pani Marszałek! Szanowny Panie Ministrze! Panie i Panowie Posłowie! Debatujemy o sprawie kluczowej z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski w kluczowym momencie i zbieramy fakty. Fakty są takie: ten projekt, projekt gazociągu północnego, jest już praktycznie skończony, ale jeszcze go można zatrzymać. Na ten projekt można ogłosić moratorium, jeszcze jest bardzo dużo możliwości działania.

To jest nasz głos i nasze wsparcie dla rządu, dla jego działania.

My nie chcemy ministra, który się skarży, że mu nie wyszło z Amerykanami czy z Niemcami. Chcemy - i proszę to, panie ministrze, bo znam pana osobiste zaangażowanie, przekazać panu ministrowi, szefowi MSZ-u - ministra aktywnego do ostatniego momentu. Wiemy, że dzisiaj trzeba zademonstrować wspólną determinację, że synergia działań wszystkich partii i stronnictw w tej Izbie może zatrzymać tej projekt, który jest groźny dla bezpieczeństwa Polski, [[Oklaski]] bo tutaj rzecz idzie o bezpieczeństwo Polski. Dzisiaj chcemy mieć pewność, że w departamencie stanu są polscy dyplomaci i przekonują urzędników departamentu stanu i waszyngtońskie think tanki, że nie wolno dopuścić do uruchomienia Nord Streamu. Chcemy mieć pewność, że dyplomaci, którzy pracują u pana ministra, są dzisiaj u Zielonych w Niemczech, są dzisiaj u chadeków i zabiegają o to, żeby rozwiązać tę sytuację do ostatniego momentu. Nie chcemy polityki zagranicznej, która polega na tym, że Polska ogłasza, że nam nie idzie. Nie chcemy polityki zagranicznej, która polega na tym, że publikuje się zdjęcia ze spotkania z prezydentem Stanów Zjednoczonych w korytarzyku.

Proszę popatrzeć, panie ministrze, i popatrzcie na to, koledzy - tylko, jak widzę, dwie osoby z większości rządowej - nas na to stać. Rozumiemy, co to znaczy zgromadzić się wokół racji stanu. Potrafimy działać wspólnie, ale chcemy waszej aktywności, a nie waszego płaczu. Chcemy waszej wizji polityki zagranicznej, a jeśli wam nie idzie, to dajcie sobie pomóc. I dlatego przyjmijcie dzisiaj nasze wsparcie dla tej uchwały, która pochodzi za późno. Nie jako brawa, nie jako ckliwość - przyjmijcie je jako wezwanie do roboty, żeby nie było za późno.

I bardzo proszę, pan poseł Maciej Konieczny, Lewica. Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Faktycznie rzadko zdarza się w polskim Sejmie taka zgodność, jaka wystąpiła w przypadku Nord Stream 2. Komisja Spraw Zagranicznych przez aklamację przyjęła uchwałę wzywającą naszych sojuszników z Unii Europejskiej, ale także Stany Zjednoczone do zablokowania szkodliwego, niebezpiecznego projektu, jakim jest Nord Stream 2. Zgadzamy się co do tego, że gazociąg stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa Europy i jest przejawem rosyjskiego imperializmu - tego samego imperializmu, który doprowadził do agresji na Ukrainie i zajęcia części ukraińskich ziem, tego samego, który doprowadził do wojny w Gruzji, tego samego, który doprowadza do brutalnej polityki wobec białoruskiej i rosyjskiej opozycji. To także przewaga Rosji wobec naszych bliskich wschodnich sąsiadów. Nieprzypadkowo Władimir Putin powiedział, że po tej inwestycji nasi wschodni sąsiedzi, w tym Ukraina, będą musieli być bardziej grzeczni. Rzadko zdarza się taka zgodność, rzadko zdarza się, aby rząd miał taki silny jednoznaczny mandat Sejmu, całego polskiego Sejmu. Trudno jednak być optymistą, słuchając gorzkich żali ministra Raua, który skarży się, że Amerykanie z nim nie rozmawiają, patrząc na wątpliwą renomę, jakiej Polska dorobiła się na arenie europejskiej, wsłuchując się w głosy padające także ze strony kręgów rządzących w takim tonie, jakby sprawa była już przegrana, jakby został nam do rozegrania już tylko mecz o honor, jakby sprawa była przesądzona i jedyne, co nam pozostało, to obwinienie Niemców za zaistniałą sytuację. Oczywiście Niemcy mają swoje na sumieniu, ale rozdzieranie szat i obwinianie kogokolwiek nie wystarczy, żeby zapewnić Polsce i naszej części Europy bezpieczeństwo. Może gdybyśmy nie tracili regularnie okazji do wykazania solidarności z naszymi najbliższymi partnerami, ostatnio przy okazji podatku od korporacji, to chętniej by z nami rozmawiali. Może gdybyśmy nie uchodzili w Europie za państwo łamiące prawo, to łatwiej byłoby nam nakłonić Niemców do przestrzegania europejskiego prawa.

Niestety budowane przez polski rząd relacje zagraniczne są zupełnie oderwane od materialnych interesów naszego kraju. Polski rząd ściska się z Wiktorem Orbánem, najbardziej prorosyjskim prezydentem Europy. Powstać ma nawet specjalna frakcja z Parlamencie Europejskim składająca się z Kaczyńskiego, Orbána, włoskich faszystów i francuskiej radykalnej prawicy. Tuż przed wizytą w Europie Joe Bidena Polska postanowiła stanąć okoniem w sprawie globalnego podatku od korporacji. To jest w ogóle świetny pomysł, ale poza tym bardzo ważny dla nowej administracji amerykańskiej. Trudno się dziwić, że taka polityka zagraniczna, bazująca na sympatiach, antypatiach i obsesjach rządzącej prawicy, dramatycznie zawodzi w najtrudniejszych momentach, takich jak ten, kiedy decyduje się przyszłość Nord Stream 2. Jeszcze jedna rzecz tu powinna paść. W kwestii Nord Stream 2 chodzi także o klimat. Ta ogromna inwestycja w gaz ziemny, a więc jakby nie było paliwo kopalne, to niezwykle niebezpieczny sygnał ze strony naszych zachodnich sąsiadów. Niemcy lubią się przedstawiać jako awangarda zielonej rewolucji energetycznej. Jednocześnie dezaktywują swoje elektrownie atomowe i sięgają po gaz, który nie jest ani zielony, ani bezpieczny. Odchodzą więc od zielonego źródła energii, energii z atomu, aby stać się europejskim centrum spalania i dystrybucji rosyjskiego gazu. Sprawa Nord Stream 2, ta rosyjsko-niemiecka umowa ponad naszymi głowami, powinna być więc dla Polski jeszcze jednym ważnym sygnałem. Sygnałem, że odejście od paliw kopalnych w stronę zielonych źródeł energii, a więc odnawialnych źródeł energii i energetyki jądrowej, to nie jest tylko kwestia klimatu, ale niezależności i bezpieczeństwa energetycznego Polski. Naprawdę dużo rzeczy w tej kwestii można było zrobić lepiej. Nie ma co udawać, sytuacja Polski w tym momencie jest ciężka. Równolegle została wstrzymana budowa Baltic Pipe. Nie jesteśmy w kwestii Nord Stream 2 w o wiele lepszej sytuacji niż nasza reprezentacja na Euro po meczu ze Słowacją, ale oczekujemy od polskiego rządu jednego: grania do końca, a nie bezradnego machania rękami i narzekania na sędziego. Polska Lewica jednoznacznie sprzeciwia się budowie i funkcjonowaniu gazociągu Nord Stream 2. To ważne, aby w tej konkretnej kwestii cały polski Sejm mówił jednym głosem. Dlatego też oczywiście głosujemy za tą ważną, potrzebną i dobrą uchwałą. Bardzo proszę, pan poseł Władysław Teofil Bartoszewski, Koalicja Polska. Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Jest to tak naprawdę skandaliczny projekt polityczny, który jest efektem, nazwijmy to po imieniu, korupcji politycznej. Pan Gerhard Schröder, kanclerz Republiki Federalnej Niemiec, podpisuje porozumienie z Federacją Rosyjską na budowę Nord Stream, po czym przegrywa wybory parlamentarne 2 tygodnie później i przyjmuje bardzo wysoko płatną pracę de facto dla Gazpromu. Przyjmuje tę pracę i utrzymuje się tam do tej pory. Jak to nie jest korupcja polityczna, to nie wiem, co nią jest. Jest to projekt, który godzi w interesy bezpieczeństwa energetycznego Polski, godzi w interesy polityczne Polski, Ukrainy, państw bałtyckich, ale również państw nordyckich, chociaż jeden z parlamentarzystów fińskich również dał się przekupić Rosjanom i prowadził lobbing. Problem został podniesiony przez moich kolegów posłów. Polega on na tym, że gdyby nasza służba zagraniczna i nasze służby, trzeba powiedzieć, funkcjonowały sprawnie, to nawiązalibyśmy alianse i porozumienia z wieloma państwami Unii Europejskiej, w tym nordyckimi, takimi jak Szwecja przede wszystkim, żeby przeciwko temu projektowi walczyć. Nasze zdolności dyplomatyczne, jeśli chodzi o Niemcy, są w tej chwili żadne. W Berlinie nikt z naszym ambasadorem nie rozmawia z powodów wszystkim wiadomych. Akurat mam niezłe stosunki w Niemczech.

Jest to oczywiste zaniedbanie z tego powodu, że ten projekt narusza również prawo europejskie, dlatego że niemal na całej długości, jak pan minister wie, gazociąg ten jest również niezgodny z zasadami rozdziału działalności przesyłowej od działalności wydobywczej i obrotu gazem ziemnym, przez co surowiec importowany tą trasą będzie w uprzywilejowanej pozycji, konkurencyjnej względem gazu sprowadzanego trasami, na których przestrzegane jest prawo Unii Europejskiej, w szczególności zasady dotyczące kalkulacji taryfy przesyłowej i dostępu stron trzecich, wynikające z tzw. trzeciego pakietu energetycznego. Mieliśmy tam pewne sukcesy w związku z ograniczeniem przepustowości OPAL-u, i to było bardzo dobre. Tak jak Czesi podnoszą argumenty przeciwko Turowowi, tak my powinniśmy podnosić argumenty przeciwko Nord Stream 2. To jest wyjątkowo szkodliwa inicjatywa, która rozbija solidarność energetyczną Unii Europejskiej.

Tak jak moi koledzy, poprzedni mówcy wzywam MSZ i polski rząd do intensywnej pracy w wielu państwach, żeby zatrzymać np. proces certyfikacji tego gazociągu.

Znaleźliśmy się w niezwykle ważnym dla europejskiej solidarności momencie dziejowym. Dziś od naszych partnerów w Unii Europejskiej, w NATO, w stolicach demokratycznego świata oczekujemy głębokiego namysłu i zrozumienia, zrozumienia sytuacji, w której podejmowane decyzje nie tylko będą ważyć na powszechnym bezpieczeństwie energetycznym kontynentu, ale i mogą doprowadzić do powstania nowego muru, takiego muru, który wspólnie burzyliśmy ponad 30 lat temu. Tylko ten nowy mur, choć budowany przez naszych przyjaciół z Niemiec, powstanie w zupełnie innym miejscu. Ten mur podzieli Europejczyków, ten mur przedzieli europejską solidarność, oddzieli Europejczyków i narody demokratycznego świata od wartości, które połączyły nas w Unii Europejskiej, w NATO. Za tym murem zostaną kobiety, mężczyźni, dzieci, zostaną ludzie, którzy też chcą żyć w pokoju. W istocie jest to narzędzie geopolityczne. Ma on bowiem umożliwić wykorzystywanie surowców energetycznych, tak jak wykorzystuje się każdą inną broń, do wywierania presji na rządy państw demokratycznego świata, by odwracały wzrok od tego, co będzie się działo za tym nowym murem. A to, co może się dziać, widzimy dziś na wschodniej Ukrainie bądź też w cyberprzestrzeni. Dlatego od naszych partnerów w Unii Europejskiej i w NATO, w stolicach demokratycznego świata oczekujemy głębokiego namysłu, zrozumienia tej sytuacji i wycofania jakiegokolwiek poparcia dla budowy tego gazociągu oraz przerwania budowy Nord Stream 2. Wysoka Izbo! Nord Stream to nie tylko narzędzie geopolityczne. Planowane podwojenie przepustowości tego gazociągu neguje cele naszej polityki klimatycznej i opóźni transformację energetyczną. Warto więc przy tej okazji przypomnieć wszystkim, że naszym celem, celem Europy, jest redukcja emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. i neutralność klimatyczna do 2050 r. Gaz powinien więc być traktowany tylko jako paliwo przejściowe, inaczej zniszczymy naszą planetę. Trzeba więc dziś także zapytać o przyszłość dzieci, przyszłość kolejnych pokoleń Europejczyków, o świat, w którym przyjdzie im żyć, ponieważ włączenie tak ogromnej przepustowości nie tylko wzmacnia lobby dążące do niszczenia klimatu, ale również wzmacnia te ośrodki, które patrzą z niechęcią na zieloną transformację. Tymczasem Polska, Niemcy, ale i cała Europa potrzebują raczej wzmocnienia działań chroniących naszą planetę przed zniszczeniem. Ten gazociąg zagraża bezpieczeństwu dostaw i konkurencji na naszych rynkach gazowych.

Ten apel skierowany był do Rządu Federalnego Niemiec i niemieckich partii demokratycznych. Wzywamy rząd do podjęcia wszystkich działań, które doprowadzą, po pierwsze, do wstrzymania poparcia dla tego szkodliwego dla Polski, dla naszego regionu i dla całej Europy projektu, po drugie, do zatrzymania budowy tego gazociągu. I dziś od naszych partnerów w Unii Europejskiej, w NATO i we wszystkich demokratycznych stolicach na całym świecie oczekujemy głębokiego namysłu, oczekujemy refleksji, oczekujemy zrozumienia sytuacji, w jakiej znaleźliśmy się my i cała Europa, i wycofania poparcia dla budowy tego gazociągu oraz przerwania budowy Nord Stream 2. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan poseł Robert Winnicki, Konfederacja. Wysoka Izbo! Takie są fakty. I ten energetyczny odpowiednik paktu Ribbentrop-Mołotow jest realizowany przez Republikę Federalną Niemiec zarządzaną od kilkunastu lat przez kanclerz Angelę Merkel. Jest realizowany bez sprzeciwu Unii Europejskiej, mimo że Donald Tusk był szefem Rady Europejskiej. Jest realizowany brutalnie przez Niemcy, tak, demokratyczne, liberalne Niemcy, którymi tak lubicie się podpierać w debacie publicznej, w ich własnym, narodowym, dobrze pojętym interesie i przeciwko interesowi Polski, ale i całego regionu, we współpracy z autorytarną Rosją. Dokładnie tak jest. I zdajcie sobie wszyscy z tego sprawę, wy, którzy tak często w walce z polskimi interesami powołujecie się na dobro Europy, na jedność, na solidarność europejską - solidarność europejska leży na dnie Bałtyku. Taka jest prawda. I tak wygląda europejska polityka klimatyczna - na dnie Bałtyku, w rurze. Ona nie istnieje, jest twarda gra interesów narodowych - wszystkich, którzy w tym uczestniczą. Ten energetyczny pakt Ribbentrop-Mołotow jest również realizowany dlatego, że bezrozumne rządy ostatnich lat postawiły wszystko nie tylko na Stany Zjednoczone, ale na jedną ekipę w Stanach Zjednoczonych, na ekipę Trumpa. I z całym szacunkiem, panie pośle Kowalski, ale kiedy pan wymienia jako autorytet Żurawskiego vel Grajewskiego, tego samego, który w zeszłym roku napisał wprost, że trzeba postawić na ekipę Trumpa i zignorować wszystkie inne opcje, to jest to właśnie poziom wyobraźni, szerokość horyzontów zaplecza PiS-owskiego w tym zakresie.

To jest właśnie efekt jednowektorowej polityki proamerykańskiej i jednowektorowej polityki proniemieckiej. Żaden efekt. Polskie elity z Platformy i z PiS, nadwiślańskie elity, się skompromitowały - skompromitowały się brakiem wyobraźni. W 2016 r. tutaj, na sali kolumnowej, ogłaszaliśmy program „Suwerenny naród” - suwerenność polityczna, suwerenność na arenie międzynarodowej. Pisaliśmy jasno, że determinantą najważniejszą naszej pozycji na arenie międzynarodowej będą w najbliższych latach dwa czynniki: rywalizacja amerykańsko-chińska i wzrost znaczenia Niemiec i Rosji. To opisaliśmy 5 lat temu, ogłaszaliśmy i staraliśmy się, by hasło: polityka wielowektorowa, czyli polityka, gdzie widzimy i Waszyngton, i Pekin, a nie tak jak pan minister Rau - po 5 latach w panice jedzie do Pekinu, bo się nagle odmieniła karta w Waszyngtonie. No, każdy, kto miał głowę na karku, mógł się spodziewać, szanowni państwo. Myśmy już 5 lat temu o tym pisali: Nie zamykać drogi do wektora chińskiego. Pamiętać, że Niemcy i Rosja pozostają najważniejszymi graczami na arenie europejskiej. Nie stawiać wszystkiego na jedną kartę, unijną czy amerykańską. Prowadzić szeroką politykę wielowektorową między tymi stolicami, między tymi mocarstwami, między Pekinem a Waszyngtonem, między Berlinem a Moskwą, bo to jest realny wektor. Gdzie jest dzisiaj Międzymorze? Nie ma ich. Jest w Turowie. Czas skończyć z tymi romantycznymi mitami i zobaczyć, jak wygląda realna polityka międzynarodowa. A realna polityka międzynarodowa to ciągle egoizm narodowy, interes narodowy poszczególnych państw, to twarda, brutalna gra każdego z każdym, niezależnie czy jest demokratyczny, autorytarny, postkomunistyczny, liberalny czy jakikolwiek inny. I zacznijmy wreszcie rozmawiać w tym parlamencie o polityce zagranicznej za pomocą tych kategorii, i zacznijmy wreszcie otwierać oczy, zamiast żyć złudzeniami. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie pośle. Czy ktoś z pań i panów posłów chce jeszcze zgłosić się do zadania pytania? Zamykam listę.

Wysoka Izbo! Nord Stream 2 i jego dokończenie to jest dowód na słabość polityki zagranicznej rządu PiS, szczególnie wobec Unii Europejskiej. Chciałbym zadać panu ministrowi pytanie: Jakie koalicje budowaliście przez te lata, ażeby zatrzymać Nord Stream 2?

Bowiem tak naprawdę Nord Stream 2 powoduje, że bezpieczeństwo energetyczne całej Europy może być zagrożone.

Tak że pytanie o tę wielką samotność czy też o sprawność negocjacyjną. Pan poseł Marek Krząkała, Koalicja Obywatelska. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Nikt na tej sali nie ma wątpliwości, że projekt budowy drugiej nitki Gazociągu Północnego jest szkodliwy i zagraża bezpieczeństwu energetycznemu nie tylko Ukrainy, ale i całej Unii Europejskiej. Nie zmienia to faktu, że działania rządu są mocno spóźnione. Dzisiaj nie przerwiemy jego budowy, ale możemy się domagać, by gazociąg nie został uruchomiony, a jeżeli tak się nie stanie, by korzystanie z niego było oparte na przestrzeganiu dyrektyw gazowych i unijnego prawa. Ale chciałem zapytać pana ministra o inną kwestię. Za 2 dni będziemy obchodzić 30. rocznicę podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Źle by się stało, gdyby te 30 lat było postrzegane jedynie przez pryzmat Nord Stream 2. Dlatego proszę pana ministra o odpowiedź na piśmie na następujące pytania. Jaka jest ocena Ministerstwa Spraw Zagranicznych realizacji postanowień traktatu na przestrzeni 30 lat? Które wspólne (Dzwonek) projekty gospodarcze, społeczne i polityczne udało się zrealizować? Jaka jest ocena i skuteczność prac, zwłaszcza w ostatnich latach okrągłego stołu powołanego do tego, by rozwiązywać problemy między naszymi krajami? I wreszcie jakie są strategiczne kierunki przyszłej współpracy polsko-niemieckiej? Bo w tej materii widać deficyt informacji. Pan poseł Michał Szczerba, Koalicja Obywatelska. Pani Poseł Beata Maciejewska, Lewica. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Rzeczywiście muszę się zgodzić z moimi przedmówcami, że jeśli chodzi o naszą dyplomację, to ona ciągle szwankuje i budowa tej nitki gazociągu jest ze szkodą dla Polski, ale sami sobie także szkodzimy, i to jeśli chodzi zarówno o nasze stosunki w Unii Europejskiej, w ogóle teraz także już na świecie, jak i o politykę energetyczną. Chcę powiedzieć, przypomnieć przy okazji tej dyskusji o tym, że bezpieczeństwo energetyczne możemy zapewnić sobie wtedy, kiedy będziemy dostarczać Polkom i Polakom energię z tego źródła energetycznego, które już mamy: ze słońca i z wiatru, kiedy będziemy stosować się do tych przepisów i tych wskazań Unii Europejskiej, które są dzisiaj dla nas kluczowe. Zamiast angażować się w spory, które są już dzisiaj bardzo spóźnione, zamiast marzyć (Dzwonek) o wielkich inwestycjach, które będą zastępować bloki węglowe, zajmijmy się tymi źródłami energii, które dzisiaj są najbardziej skuteczne dla naszych kieszeni i dla ochrony klimatu. Dziękuję. Pan poseł Artur Łącki, Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo!

Turkish Stream, turecki potok, gazociąg biegnący z Rosji do Turcji dnem Morza Czarnego, omijający Ukrainę.

Pytanie jest takie. Co nasza dyplomacja zrobi, jeśli ten wystartuje? Wystartuje i pan dobrze o tym wie. Nie macie. Pan poseł Andrzej Szejna, Lewica. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Przecież, panie ministrze, pan zna się na sprawach niemieckich, pisał pan doktorat, przecież Neue Ostpolitik, polityka energetyczna Niemiec jest znana od lat 70., tylko wy wszystko robiliście przez te lata, aby - jak się okazuje - niszczyć politykę energetyczną Polski albo aby w ogóle jej nie było. Dzisiaj polityka energetyczna to jest core polityki zagranicznej każdego kraju.

I na koniec powiem panu taką ciekawą rzecz. Dzisiaj spotyka się Biden z Putinem. Otóż tak się składa, że dzięki dobrej policy to polityka zagraniczna Rosji okazuje się być chomikiem, a polityka zagraniczna PiS robi z nas szczura politycznego na arenie międzynarodowej. Dziękuję. Bardzo proszę, pan poseł Tomasz Olichwer, Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo! Oczywiście zgadzam się z meritum tej uchwały oraz cieszę się, że wszyscy wnioskodawcy ponad podziałami wypracowali wspólne stanowisko, lecz czytając wcześniej uzasadnienie pierwszego projektu, podpisanego przez posłów głównie Solidarnej Polski, przecierałem oczy ze zdumienia. Piszecie w nim, zresztą całkiem słusznie, że projekt Nord Stream 2 w swoich założeniach podważa zasadę europejskiej solidarności energetycznej oraz przeczy regułom konsultacji i współpracy w ramach Unii Europejskiej. Przypominacie również wyrok TSUE w sprawie gazociągu OPAL. Na koniec, również słusznie, sugerujecie państwo, że Niemcy w imię europejskich zasad winny natychmiast porzucić partykularne interesy i zacząć kierować się przede wszystkim interesem Unii Europejskiej jako wspólnoty państw członkowskich. Wszystko pięknie, tylko nasuwa się pytanie: Skąd u was taka zmiana narracji i szacunek do wartości europejskich? Ale to dobrze wróży na przyszłość. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan poseł Jan Warzecha, Prawo i Sprawiedliwość. Panie Ministrze! Wysoki Sejmie! Miło słyszeć, że w wielu kwestiach jesteśmy zgodni. Miło było słuchać pana posła Władysława Teofila Bartoszewskiego.

Przykro było słuchać wypowiedzi niektórych z państwa krytykujących rząd, że rzekomo mało robi, nic w tej kwestii nie robi, że rzekomo mamy ambasadora, który przez Niemców nie jest podziwiany. Drodzy państwo, jeśli ktoś broni swoich interesów, nigdy nie będzie lubiany, podziwiany przez drugą stronę i tak jest z panem ambasadorem Niemiec.

Dziękuję bardzo. Pan poseł Michał Gramatyka, Koalicja Obywatelska. Nie ma pana posła. Pan poseł Dariusz Rosati, Koalicja Obywatelska.

Szanowna Pani Marszałek! Panie Ministrze! Oczywiście wszyscy poprzemy tę uchwałę, bo jakie mamy wyjście w tej sytuacji, ale nie sposób nie zadać sobie pytania, jak mogło do tego dojść. Jak mogło dojść do sytuacji, w której polski minister spraw zagranicznych skarży się, że o wycofaniu sankcji amerykańskich dotyczących Nord Stream 2 dowiedział się z mediów? Panie ministrze, co robiła polska dyplomacja? Co robią te dziesiątki ludzi zatrudnionych przez was w placówce w Waszyngtonie?

Może wreszcie zadacie sobie pytanie, jak mogło dojść do tej sytuacji.

Może wreszcie dowiemy się, dlaczego wszystkie drzwi w Waszyngtonie są dla was i dla waszych urzędników zamknięte, w Berlinie również i w Brukseli także. Dziękuję bardzo, panie pośle. Pani poseł Małgorzata Niemczyk, Koalicja Obywatelska.

Panie Premierze! Chciałabym, aby pan odpowiedział na pytanie: Czy poznał pan już przyczyny, czy już pan wie, dlaczego nie jesteście skuteczni w prowadzeniu polityki zagranicznej, dlaczego ciągle ponosicie porażki? Co zrobiliście skutecznego w sprawie niewybudowania Nord Stream? Brakuje partnerów Polski do zablokowania tego projektu. Oponowaliście, protestowaliście? Uważaliście, że wam się to uda samym? W 1997 r. młody doktorant Władimir Putin napisał, że zapotrzebowanie na energię w Europie stwarza okazję do zbudowania trwałej zależności energetycznej, a od kiedy rządzicie, Polska traci sojuszników. Poza wyjechaniem na San Escobar, bo mam uczucie, że tam większość polityki zagranicznej jest uprawiana. Panie Ministrze! Wysoka Izbo!

Chcę zapytać, jak to jest możliwe, że dzisiaj rozmawiamy na ten temat. PiS po 5 latach przypomniał sobie, że mamy do czynienia z ogromnie poważną sprawą, sprawą budowy Nord Stream 2. I jest kolejny symbol, a w zasadzie już nawet tego symbolu nie ma, to polityka zagraniczna. To, o czym dzisiaj rozmawiamy, jest emanacją braku polityki zagranicznej. Nie słabej polityki, ale jej braku.

Pozycja Polski w sposób oczywisty słabnie również w Unii Europejskiej i w regionie. Szybkie pytanie, bo my oczywiście będziemy głosować, ale jaka jest alternatywa dla jamalskiego gazociągu? Co rząd planuje zrobić, jeśli zostanie wyłączony jamalski gazociąg?

Bardzo proszę, pan poseł Grzegorz Rusiecki, Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo! Bezpieczeństwo to kwestia polskiej racji stanu. Ale czy wasze działania oparte są na partnerstwie? Wątpliwe sukcesy dyplomacji PiS-owskiej budzą już nie tylko nasz sprzeciw, ale powodują także realne niebezpieczeństwo dla państwa. Podstawową zasadą współpracy, relacji ogólnoludzkich jest szacunek. Jeżeli domagamy się go od innych, to sami najpierw musimy go okazać naszym partnerom. Jeżeli ten szacunek państwo okazujecie w ten sposób, w jaki dzisiaj uwidaczniacie - zwracam się do rządu - szacunek dla tej Izby, a w zasadzie jego brak, bo nie ma na sali ani premiera, ani ministra spraw zagranicznych, a wszyscy zgadzamy się, że temat, o którym dyskutujemy, jest niezwykle istotny, to strach pytać, jak wyglądają (Dzwonek) szacunek i relacje, jeśli chodzi o naszych partnerów międzynarodowych. Ale w związku z tym chciałbym zapytać, z kim dziś współpracujemy, kogo pozyskaliśmy dla naszych racji, kto razem z nami będzie dbał o interes Polski. Bardzo proszę, pani poseł Małgorzata Tracz, Koalicja Obywatelska. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Nord Stream 2 stanowi wielkie zagrożenie dla Polski i dla jedności Unii Europejskiej, stanowi wielkie zagrożenie dla ochrony klimatu. Projekt Nord Stream 2 uderza w bezpieczeństwo Polski i Europy, służy Kremlowi jako klin do rozbicia europejskiej solidarności, do skonfliktowania krajów Unii Europejskiej, bo słaba i skłócona Unia Europejska jest w interesie Moskwy. Nord Stream 2 jest bardzo złym projektem dla klimatu. Będzie na kolejne lata utrwalał dominację paliw kopalnych w miksie energetycznym, a przecież cała Europa zgodnie z polityką klimatyczną ma odchodzić od paliw kopalnych w stronę energii ze źródeł odnawialnych, w stronę ograniczenia emisji o 55% do 2030 r. i neutralności klimatycznej do 2050 r. W Niemczech we wrześniu będą wybory.

Bardzo proszę, pani poseł Krystyna Skowrońska, Koalicja Obywatelska.

Powiem dzisiaj: Wielce Szanowna Pani Marszałek! Panie Ministrze! To prawda, państwo powinni się wytłumaczyć.

Państwo powinniście się wytłumaczyć z tego, dlaczego na tamtym etapie tego nie zablokowaliście, nie podjęliście skutecznych działań, aby te 1222 km rurociągu nie powstały.

Państwo zmarnowali ostatnie 6 lat.

Dziękuję bardzo. Ostatnie pytanie, pan poseł Jan Szopiński, Lewica. Wysoka Izbo! Debata nad apelem o zaprzestanie budowy gazociągu Nord Stream 2 w chwili, gdy poinformowano o zakończeniu budowy pierwszej nitki i rozpoczęciu napełniania jej surowcem, jest chyba jednak kompromitująca. Równie kompromitujące są argumenty, że istnienie gazociągu doprowadzi do zerwania z zasadą dywersyfikacji dostaw paliw do Europy, gdyż istnienie gazociągu oraz potencjalnego dostawcy gazu niczego nie zmienia. Czy nie jest tak - chciałbym otwarcie zapytać - że głównym powodem protestu rządu jest utrata opłat transferowych oraz pominięcie Polski w chwili podejmowania decyzji o budowie gazociągu, a nie wymieniana w dokumentach agresja Rosji na Ukrainę? Trzeba postawić jasno pytanie, dlaczego inwestorzy zdecydowali się na wielokrotnie droższą trasę morską omijającą nasz kraj. Dziękuję bardzo.

Pani Marszałek! Może zacznę od pewnej korekty kalendaryjnej, bo mam wrażenie, że pani poseł Skowrońska się pomyliła. To są lata poprzednich rządów Prawa i Sprawiedliwości. Wtedy rząd Prawa i Sprawiedliwości w sposób bardzo zdecydowany i jasny to krytykował i podejmował działania sprzeciwiające się powstaniu Nord Stream 1, bardzo wyraźnie zaznaczam: pierwszej nitki gazociągu. Miałem zaszczyt współpracować z europosłem Marcinem Libickim. Byłem współautorem, pracowałem nad projektem rezolucji Parlamentu Europejskiego sprzeciwiającej się budowie Nord Stream 1, przyjętej zdecydowaną większością głosów europosłów w Parlamencie Europejskim. Ale później, po roku 2007 polska polityka zagraniczna się zmieniła, pani poseł. Władzę objęła Platforma Obywatelska. Bo było też pytanie o zaangażowanie Donalda Tuska ze strony pana posła Jana Warzechy. W 2008 r. zaangażowanie Donalda Tuska było takie, że mówił, że Władimir Putin to jest nasz człowiek w Moskwie. To za państwa rządów ta pierwsza nitka Nord Stream 1 - ten pierwszy krok burzący solidarność energetyczną Unii Europejskiej - została oddana. A więc przepraszam bardzo, po pierwsze, jeśli chodzi o kalendarium, wyjaśniam, że to za czasów rządu Platformy Obywatelskiej zbudowano pierwszą nitkę gazociągu i oddano do użytku pierwszą nitkę gazociągu Nord Stream, więc akurat państwo macie najmniejszy tytuł, żeby w tej sprawie zadawać pytania i podnosić wątpliwości co do skuteczności i efektywności działań obecnego rządu. To rzecz pierwsza. Kalendarium powstawania nitki Nord Stream 2. Być może pani poseł tutaj też nie ma precyzyjnej wiedzy. 18 czerwca 2015 r. - to, zdaje się, też jeszcze państwa rządy, jeśli dobrze pamiętam - podpisane memorandum między Gazpromem a niemiecką firmą E.ON, brytyjską firmą Shell, austriacką firmą OMV na budowę drugiej nitki gazociągu Nord Stream 2. 4 września 2015 r. - państwa rządy. Co wówczas robi rząd Platformy Obywatelskiej? Ja pani odpowiem, co robi. Wówczas rząd Platformy Obywatelskiej zajmuje się migrantami i łamaniem solidarności w Grupie Wyszehradzkiej. To jest wówczas temat dla rządu Platformy Obywatelskiej, a nie umowy i rozpoczynające się działania zmierzające do powstania Nord Stream 2.

Padło pytanie, czy zbudowaliśmy koalicję, pan poseł Piotr Nowak o to pytał. Kiedy przejmowaliśmy rządy, byliśmy osamotnieni, bo Platforma nie potrafiła zbudować żadnej koalicji w tej sprawie. Tymczasem Prawo i Sprawiedliwość ten problem zinternacjonalizowało. Okazało się, że można pozyskać aktywny głos krajów bałtyckich; że można nawet w ostatnim czasie pozyskać aktywny głos Francji, głos jednego z francuskich ministrów; że można nawet wywołać w Niemczech debatę i pozyskać sojuszników, np. w gronie niemieckich Zielonych bardzo jasno wypowiadających się w tej sprawie; że można pozyskać życzliwość administracji amerykańskiej. To, że dzisiaj administracja amerykańska popełnia, w naszej opinii, błąd, i to, że pan minister Rau publicznie na ten błąd wskazuje, to nie jest żadne żalenie się, panie pośle, to nie jest żadne płakanie po gazetach. To jest jasny sygnał, że nie będziemy zamykać oczu na błędy naszego ważnego strategicznego sojusznika. Bo nie jest tak, że jeżeli ktoś jest naszym strategicznym sojusznikiem, to my milczymy, gdy chodzi o jego błędy, i udajemy, że nic się nie dzieje. O tym też trzeba publicznie mówić, jeżeli ten sojusznik popełnia błędy. Chciałem jednak skoncentrować się na tej uchwale, bo dyskusja. Rozumiem, że jest potrzeba wyrażenia różnych głosów, skrytykowania rządu, zadania różnych pytań. Chętnie bym państwu jeszcze szczegółowo poopowiadał, ale widzę, że ograniczenie czasowe jest bezlitosne. Moją satysfakcją jest jedno, że ze strony tej sali - i za to pragnę panu posłowi Kowalskiemu, panu posłowi Kowalowi, państwu posłom, wszystkim, koalicji i opozycji, bardzo serdecznie podziękować, że z tej sali płynie silny, jednoznaczny, jednolity i ponadpartyjny głos krytykujący tę inwestycję, głos solidarności, bo jest to głos nie tylko w imieniu Polski, ale solidarności z Ukrainą, z państwami bałtyckimi. Polska jest krajem solidarności. Polska jest krajem solidarności i (Dzwonek) nie może godzić się na projekt łamiący solidarność, odtwarzający podziały w Europie, projekt egoistyczny, realizujący partykularne interesy. Jest to projekt zgłoszony we właściwym momencie, kiedy niestety pojawiają się sygnały o planowanych błędnych decyzjach ze strony naszego strategicznego sojusznika, w momencie rozczarowującego sygnału ze strony Stanów Zjednoczonych, w momencie, w którym w Niemczech jest otwarta debata i zbliżają się wybory. To nie jest głos spóźniony. Gdyby działania dyplomacji polskiej były spóźnione, gazociąg Nord Stream byłby już oddany do użytku. Nie jest oddany do użytku i mamy nadzieję, że nie będzie nigdy uruchomiony właśnie ze względu na skuteczne i aktywne działania polskiej dyplomacji.

Także w zeszłym tygodniu miałem okazję spotykać się z przedstawicielami fundacji, zarówno fundacji Adenauera, ważnej fundacji związanej z niemieckim CDU, jak i fundacji Bölla związanej z niemieckimi Zielonymi. I jesteśmy w stałym kontakcie z wieloma niemieckimi partnerami. W tym tygodniu wizyta niemieckiego prezydenta, w zeszłym tygodniu odbyło się kolegium w Pałacu Prezydenckim przygotowujące do tej wizyty. Temat Nord Stream 2 na pewno będzie jednym z kluczowych tematów tej wizyty, ale będzie też wizyta ministra spraw zagranicznych Niemiec na początku lipca w Warszawie. Zapewniam państwa: rząd Polski jest aktywny, ma kontakt ze wszystkimi ważnymi partnerami tak na niemieckiej scenie politycznej, jak i na scenach politycznych wielu krajów w Europie i ten temat podnosi wysoko i aktywnie w agendzie. Ale ta uchwała Sejmu, za którą jeszcze raz państwu serdecznie dziękuję, wzmacnia nasz mandat do rozmowy, zostanie wykorzystana przez placówki zaraz po przyjęciu, aby przekazać ją naszym partnerom i powiedzieć o jednolitym, ponadpartyjnym głosie polskiego Sejmu. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan poseł Bartoszewski. Panie Ministrze! Oczywiście, że wszyscy na tej sali, cała opozycja, dajemy rządowi do ręki mocną i zdecydowaną uchwałę, jasno wyrażającą stanowisko naszego parlamentu w sprawie budowy Nord Stream 2, ale, jak mówił pan poseł Kowal, wy tego nie zmarnujcie, dlatego że nie chodzi o to, żeby jeździć wyłącznie do Niemiec i rozmawiać z partnerami niemieckimi, jakkolwiek by to było ważne.

Po pierwsze, nie było rozmów z Niemcami, bo wtedy prowadziliśmy politykę zdecydowanie antyniemiecką, a po drugie, nie wykorzystaliśmy możliwości z innymi potencjalnymi sojusznikami, np., że wymienię jedno państwo, Szwecja, która była gotowa przeciwko temu występować, ale po cichu, a nie publicznie. Oczywiście gdyby budowa tego gazociągu była spóźniona i do rządu weszła partia Zielonych, co jest całkiem prawdopodobne, byłaby lepsza sytuacja, no ale jest, jak jest. Francja, o której pan wspomniał. Ale Białoruś nie ma tutaj głosu. Najpierw poparli nas, a potem poparli Niemców. Zwracam się z apelem, tak jak pan poseł Kowal: nie zmarnujcie tej szansy. A do pana ministra Kamińskiego z apelem: wykorzystujcie służby, które są w stanie was ostrzec przed tym, co się dzieje, cośkolwiek wcześniej. Dziękuję. W trybie sprostowania pani poseł Krystyna Skowrońska. Szanowna Pani Marszałek!

Decyzje, które były podejmowane od 2005 r., w 2006 r., pierwsza nitka, druga nitka - to państwa nieudane negocjacje, to państwa nieudane działanie. Wy przyznajcie się do własnych. Cała sala, cały Sejm poprze tę uchwałę, ale państwo musicie się wziąć do roboty, o czym mówili pan poseł Bartoszewski, pan poseł Kowal i pan poseł Rosati.

Bo pan wstaje i oczywiście zaczyna mówić o tym, że to jest wina Tuska i w ogóle wszystkich po kolei, tylko nie wasza. Ja zadałem konkretne pytanie.

Tylko powiem to: Rozbijanie solidarności europejskiej jest wtedy, kiedy Niemcy korzystają z Nord Stream 2, a nie ma rozbijania solidarności europejskiej wtedy, kiedy Węgrzy korzystają z Turkish Stream. Albo walczymy w ogóle z Rosją i z przesyłem jej gazu, i ratujemy Ukrainę, albo jesteśmy hipokrytami i przyznajmy to. Ale to nie było sprostowanie. Zamykam dyskusję. Do głosowania nad projektem uchwały przystąpimy w bloku głosowań. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 3. porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo bankowe (druk nr 1236) Proszę podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów pana Jana Sarnowskiego o przedstawienie uzasadnienia projektu ustawy. Mam przyjemność przedstawić Wysokiej Izbie rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo bankowe. To jest drugi pakiet Slim VAT, czyli ustawa wdrażająca kilkanaście postulowanych przez firmy uproszczeń w rozliczaniu VAT-u. Pierwszy pakiet uproszczeń wszedł w życie w styczniu tego roku. To jest jego druga odsłona. Źródłem tych rozwiązań są propozycje zgłaszane do ministerstwa przez rzecznika małych i średnich przedsiębiorców, organizacje zrzeszające przedsiębiorców, w szczególności Konfederację Lewiatan i Polską Organizację Handlu i Dystrybucji. Kluczowe zmiany to wygodniejsze korygowanie rozliczeń, ułatwienia w obrocie nieruchomościami i elastyczniejsze korzystanie z ulgi na złe długi i z mechanizmu podzielonej płatności w VAT. Np. łatwiej będzie firmie skorygować rozliczenie, jeśli zapomniała zgłosić nam fakturę, wpisano na nią złą cenę albo np. pojawił się rabat post factum. Dzięki zmianom firmy będą mogły łatwo grupować korekty, dzięki czemu ich rozliczanie będzie znacznie wygodniejsze. Tylko w zeszłym roku takie błędy, takie korekty zgłosiło aż 55 tys. podatników, którzy rozliczyli za późno 1,5 mln faktur. Teraz łatwiej będzie dokonywać takich korekt. Wydłużymy czas na skorzystanie z ulgi na złe długi w VAT z 2 do 3 lat. Nie będzie już potrzebne specjalne oświadczenie wysyłane do urzędu skarbowego - strony transakcji będą mogły po prostu złożyć oświadczenie o objęciu VAT-em transakcji przez adnotację na samym akcie notarialnym. Dzięki zmianom w mechanizmie podzielonej płatności otworzymy podatnikom możliwość płacenia z konta VAT-owskiego należności wobec KRUS-u oraz przekazywania środków między rachunkami VAT w różnych bankach. Teraz w ramach mechanizmu podzielonej płatności z konta VAT-owskiego można płacić nie tylko VAT na konta kontrahentów, ale również regulować należności z tytułu VAT-u, z tytułu podatków dochodowych, akcyzy, cła oraz ZUS-u. Dzięki naszej propozycji będzie można również regulować składki KRUS - to będzie realne ułatwienie dla 84 tys. podatników, którzy są czynnymi podatnikami VAT i prowadzą działalność rolniczą. Przedstawiając powyższe, uprzejmie proszę Wysoką Izbę o przyjęcie projektu ustawy w wersji zaproponowanej przez rząd. Dziękuję. Dziękuję, panie ministrze. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół. Jako pierwszy pan poseł Sylwester Tułajew, Prawo i Sprawiedliwość. Szanowna Pani Marszałek! Mam ogromny zaszczyt i honor przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość wobec rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo bankowe. Art. 1 wprowadza 12 zmian w ustawie o podatku od towarów i usług.

Ten projekt już właściwie został dosyć szczegółowo przedstawiony przez pana ministra. Chciałbym zaznaczyć, że celem proponowanych rozwiązań jest dalsze uproszczenie rozliczania przez podatników podatku od towarów i usług, chodzi o tzw. pakiet Slim VAT 2, o którym wspominał również pan minister.

Chciałbym zaznaczyć, że wprowadzenie w ostatnich latach narzędzi uszczelniających system VAT oraz związane z tym efekty w zakresie walki z nadużyciami w systemie VAT pozwoliły na weryfikację rozwiązań dotyczących rozliczania VAT, w niektórych przypadkach obowiązujących od roku 2004. Celem przeprowadzonego audytu tych rozwiązań było wyeliminowanie obciążeń administracyjnych w zakresie rozliczania podatku VAT po stronie podatników. Pakiet Slim VAT 2, o którym dyskutujemy, wpisuje się również w odpowiedź na postulaty przedsiębiorców, które są kierowane do prezesa Rady Ministrów, do ministra finansów z prośbą o ich uwzględnienie, ale również mówimy tutaj o zapisach, które przeciwdziałają negatywnym skutkom społeczno-gospodarczym pandemii COVID-19.

Dopuszczenie możliwości regulowania z rachunku VAT również składek ZUS zrównuje sytuacje podatników opłacających składki na ubezpieczenie społeczne, gdyż obecnie funkcjonujące przepisy umożliwiały w takim przypadku regulowanie wyłącznie składek ZUS. Ta zmiana ma istotne znaczenie w konsekwentnym zmniejszaniu ewentualnego ryzyka dotyczącego pogarszania się płynności finansowej podatników wynikającego z ograniczonej dyspozycyjności środków zgromadzonych na rachunku VAT. W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość proszę Wysoką Izbę o przyjęcie tego bardzo dobrego projektu ustawy. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan poseł Wojciech Saługa, Koalicja Obywatelska. Dziękuję bardzo, pani marszałek. Wysoka Izbo!

Po przemówieniu pana ministra Sarnowskiego chciałoby się bić brawo i powiedzieć: świetnie.

Ustawa o VAT ma razem z rozporządzeniami 1 tys. stron i przedsiębiorcy kompletnie jej nie rozumieją, a jest to główna przeszkoda w prowadzeniu działalności, bo ludzie mówią: nie stawki. Szczególnie dotyczy to ustawy o VAT, zniechęca to ludzi do prowadzenia działalności gospodarczej.

Kto to ma zrozumieć? Bo korporacje z prawnikami na etatach, z doradcami podatkowymi, z kancelariami prawnymi, urzędnicy zrozumieją to, ale, tak jak mówię, piekarz, hurtownik czy restaurator będą mieć bardzo duże kłopoty ze zrozumieniem tej ustawy i w ogóle przepisów, które obowiązują w Polsce.

Potem trzeba to jeszcze zrozumieć, zapamiętać.

Dlaczego? Pytamy przedsiębiorców, dlaczego nie chcą korzystać z tak świetnych rozwiązań, o których mówił pan minister Sarnowski i zapewniał, że będzie świetnie. To jest główna bolączka przepisów podatkowych w Polsce. Oczywiście, te rozwiązania, o których dzisiaj mówimy, wydają się bardzo korzystne.

Jeżeli człowiek nie rozumie prawa, nie może go stosować, nie chce go stosować i odrzuca je.

Wysoka Izbo!

Dziękuję bardzo.

Brawo, brawo dla pana posła. Panie Ministrze! Wysoka Izbo!

Celem proponowanych rozwiązań jest dalsze upraszczanie rozliczenia przez podatników podatku od towarów i usług, tzw. pakietu SLIM VAT 2.

Niewątpliwie takie projekty i takie zmiany przybliżają nas do tego celu, dlatego już w tym momencie zadeklaruję wsparcie i poparcie tego projektu.

Niemniej jednak będzie to porządkować niektóre sprawy, dlatego też należy zmodyfikować definicję państwa członkowskiego. Liczę na to, że tego typu projektów ustaw, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, będzie więcej, nawet jeśli to drobne kroki.

Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan poseł Czesław Siekierski, Koalicja Polska. Szanowna Pani Marszałek! Szanowni Państwo! Z początkiem tego roku zaczął obowiązywać nowy pakiet zmian w podatku VAT. Miał on na celu uszczelnienie tego podatku oraz wprowadzenie uproszczeń dla podatników.

Te zmiany zostały zaproponowane właśnie w omawianym projekcie. Ja chciałbym wskazać tylko trzy. Po pierwsze, umożliwienie podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonywania korekty deklaracji w sytuacji, gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowy sposób wysokości podatku. Po drugie, ulgi za złe długi. Tutaj chodzi o to, że wierzyciel będzie mógł skorzystać z tej ulgi na złe długi, jeżeli wierzytelność zostanie potwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu. Po trzecie, wprowadzono możliwość wydania zgody na uwolnienie środków z rachunku VAT, jeżeli posiadane przez podatnika zaległości podatkowe zostały odroczone lub rozłożone na raty. Stworzono także możliwość uproszczenia rozliczeń, jeśli chodzi o nową sytuację związaną z brexitem. Jednak chciałbym skorzystać z możliwości odniesienia się do pewnych informacji, pewnych poglądów, które są związane ze sprawami VAT-owskimi. Rząd PiS-u często podkreśla swoje zasługi w zakresie ściągalności podatków czy też skutecznej walki z mafiami VAT-owskimi. Jednocześnie deprecjonuje dokonania rządu PO-PSL w tym zakresie. Od listopada 2015 r., kiedy został utworzony rząd PiS, w swoich działaniach, pracach wykorzystał - i dobrze, że wykorzystał - i wprowadził większość działań, które wcześniej zostały przygotowane przez rząd PO-PSL w zakresie przestrzegania przepisów podatkowych i organizacji administracji podatkowej. Zostały one przygotowane w resorcie finansów, kiedy ministrem był Mateusz Szczurek. W kwietniu 2014 r. został przyjęty dokument pt. „Działania zwiększające stopień przestrzegania przepisów podatkowych i poprawiające efektywność administracji podatkowej na lata 2014-2017” Dokument ten określał listę koniecznych działań na lata 2014–2017, definiując dla każdego projektu cel, planowane narzędzia, adresatów oraz szacowane pozytywne skutki dla sektora finansów publicznych. Istotną grupę w tym dokumencie stanowiły projekty, których celem był pozytywny wpływ na poprawę ściągalności podatku. Dotyczyły one zarówno usprawnienia samego procesu egzekucji należności podatkowych, jak i zwiększenia stopnia dobrowolnego regulowania należności podatkowych. Zaproponowane w dokumencie działania dotyczyły także wykorzystania systemów informatycznych i baz danych w celu identyfikacji i analizy zagrożeń, co miało poprawić skuteczność i efektywność działań legislacji podatkowej.

Prowadzone wtedy przez ministra Szczurka działania miały korzystny wpływ na poprawę realizacji strategicznych celów, jakimi były poprawa ściągalności podatków oraz zwiększenie efektywności administracji podatkowej.

Tylko trzeba mówić o tym, kto je przygotował. W tym czasie w ekipie ministra Szczurka był pan minister i myślę, że trzeba o tym mówić, [[Dzwonek]] bo przyszliście na gotowe, [[Oklaski]] dobre rozwiązania i efekty przyszły dopiero w waszym okresie. Bardzo proszę, pan poseł Mirosław Suchoń, Polska 2050. Szanowny panie pośle, zostawił pan okularki, tak mi się wydaje. Okulary pan zostawił, tak. Bardzo proszę.

Szanowna Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić w imieniu Koła Parlamentarnego Polska 2050 stanowisko wobec rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo bankowe ujętego w druku nr 1236. Wysoka Izbo! W przedstawionym do projektu uzasadnieniu rząd wskazał, iż celem proponowanych rozwiązań jest uproszczenie rozliczenia przez podatników podatku od towarów i usług. Przedstawione Wysokiej Izbie rozwiązania nazwano pakietem slim VAT 2. I choć wielkie deklaracje wydają się na wyrost, ponieważ sam projekt nie jest zbyt duży, a na dodatek zawiera także inne przepisy, to jednak każde rozsądne rozwiązania, w tym ułatwienia dla przedsiębiorstw, uważamy za dobre. Polska 2050 proponuje systemowe podejście do kompleksowego odbiurokratyzowania, ponieważ system podatkowy jest zbyt skomplikowany, a obsługa stanowi zbyt istotny element obciążający podmioty gospodarcze, co oczywiście ma dla tej gospodarki negatywne skutki. Na szczegółowe rozpatrywanie projektu przyjdzie czas podczas posiedzenia komisji, natomiast chciałbym powiedzieć o kilku zmianach ujętych w tym projekcie. Po pierwsze, wprowadzenie regulacji, która w przypadku eksportu towarów lub wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów określałaby wyraźnie, której dostawie należy przypisać wysyłkę lub transport. Takie rozwiązanie nie wpłynie na obecnie stosowaną praktykę, jednak zwiększy pewność prawną podmiotów biorących udział w transakcjach łańcuchowych, co oczywiście jest dobrym rozwiązaniem. Zmianą na plus jest także umożliwienie podatnikowi rozliczającemu podatek VAT z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonania korekty tej deklaracji w sytuacji, gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku. Brak dzisiaj jednoznacznych regulacji w tym zakresie powoduje wątpliwości prawne podatników i jest przedmiotem wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych, co jest zasadniczo wielkim problemem naszego systemu podatkowego. Ważną zmianą jest również wydłużenie terminu złożenia informacji o poniesieniu pierwszego wydatku na pojazd samochodowy wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika w powiązaniu z momentem złożenia JPK za zakończony okres. Obecnie podatnik dokonujący nabycia czasami nie ma możliwości terminowego złożenia naczelnikowi urzędu skarbowego informacji, która umożliwia odliczenie podatku. Projektowana zmiana poprawia sytuację podatników w tym zakresie, choć sam system skomplikowanego rozliczenia użytkowania pojazdów to jest zasługa ni mniej, ni więcej, tylko siedzącego tutaj, obecnego rządu. Projekt zawiera również przepisy dopuszczające możliwość składania oświadczenia o wyborze opodatkowania nieruchomości w akcie notarialnym. W efekcie podatnicy dokonujący wyboru złożenia tego zgodnego oświadczenia w akcie notarialnym nie będą mieli odrębnego obowiązku składania oświadczenia. To oczywiście jest również krok w dobrą stronę. W projekcie ujęto ponadto inne zmiany dotyczące terminów odliczeń, uwalniania środków czy korekt deklaracji, o czym szerzej będziemy rozmawiać w trakcie posiedzenia komisji. Po pierwsze, w projekcie ujęto szereg przepisów, które kilka lat temu zostały przepchnięte przez Sejm przez obecny rząd, choć były sprzeczne z prawem europejskim i bardzo niekorzystne dla przedsiębiorców, takich jak regulacje dotyczące złych długów, o czym wtedy mówiliśmy, panie ministrze. Dziś rząd wycofuje się z tego rakiem, oczywiście po orzeczeniu Trybunału. Można było wtedy posłuchać naszych merytorycznych argumentów i w ogóle to odrzucić. Po drugie - mówiłem o tym na początku - jest to dosyć skromna nowelizacja, a jednocześnie kolejna zmiana przepisów ustaw podatkowych w tym roku.

Pojawia się pytanie systemowe: Czy nie należy wprowadzić pewnych zasad, które uspokoją ten legislacyjny pęd? Wreszcie po trzecie, ważne jest to, czego w tej ustawie nie ma. Zabrakło zdecydowanie szerszych zmian upraszczających życie naszym przedsiębiorstwom i, co najważniejsze, przyspieszenia zwrotów podatkowych. Panie ministrze, biorąc pod uwagę kosmiczny poziom informatyzacji, którym rząd chwali się na lewo i prawo, oraz - co za tym idzie - łatwy dostęp do danych (Dzwonek), nie powinna już stanowić problemu trwającego kilkadziesiąt długich dni ocena, czy zwrot się należy, czy nie. Te zwroty podatkowe powinny więc być zdecydowanie szybsze. Dlatego w imieniu Koła Parlamentarnego Polska 2050 wnoszę o przekazanie projektu do komisji w celu dalszych prac. Dziękuję bardzo, panie pośle. Na początku trochę niemerytorycznie, ale nie mogę się powstrzymać, żeby się trochę nie popastwić nad tą nieszczęsną nazwą. Chciałbym wiedzieć, co, do jasnej Anielki, w polskim języku urzędowym, w języku urzędowym Rzeczypospolitej znaczy nazwa: slim VAT.

To nie jest slang młodzieżowy, to nie jest kolejna reklama telewizyjna nowego designu kołpaków, tylko jednak to jest źródło prawa.

Myślę jednak, że to nie jest przypadek, bo może jest to dobra ilustracja tego, jak bezsensowny, zawiły, niekonsekwentny i pełen złych pomysłów z importu jest nasz system podatkowy. Rzeczywiście skrótowce: VAT, PIT, CIT też niczego nie oznaczają w polskim języku urzędowym. Obawiam się, że tego rodzaju całkowicie zbędne zapożyczenia są niestety odzwierciedleniem naszego kompleksu niższości wobec Zachodu. Chyba uważamy tak, że nasz język nie jest wystarczająco fajny, fachowy, żeby nazywać nowe zjawiska po swojemu. Wydaje nam się, że jak jakąś głupotę powiemy po angielsku, to ona zaraz przestaje być taka głupia. Od razu tak powiało Europą. Ale dobrze, dość już lingwistycznych zmartwień. Sama ustawa to właściwie jest krok w dobrym kierunku, ale chyba jednak lepiej powiedzieć: kroczek. Mamy do pokonania daleką drogę do normalności. Jesteśmy w środku ciemnej, gęstej dżungli, przez którą podatnik musi się przedzierać z maczetą w ręce. Całe wielkie odchudzanie VAT-u to tylko spiłowanie kilku najbardziej dokuczliwych gałązek. I to jest prawdziwa skala tej plagi, jaką jest nasz system podatkowy. Gdybyśmy chcieli zrobić odważny krok do przodu, powinniśmy zająć się czymś tak fundamentalnym jak np. data powstania obowiązku podatkowego. Jest to całkowicie niedorzeczny pomysł, żeby obowiązek zapłacenia podatku powstawał w momencie wykonania usługi czy dostarczenia towaru, a nie w momencie otrzymania zapłaty. Ludzie muszą w wielu sytuacjach płacić podatek od pieniędzy, których nigdy nie zobaczyli.

Sama stabilizacja prawa, sama pewność prawa jest ważną wartością dla przedsiębiorców. Trzeba radykalnie uprościć ten podatek, zlikwidować cały bizantyjski system stawek, zwolnień, wyjątków, wyjątków od wyjątków, wyłączeń od wyjątków od tamtych wyjątków. Przedsiębiorca ma się zajmować produkcją i usługami, a nie studiowaniem kolejnych leksykonów. Wtedy może ten podatek zasłuży sobie wreszcie na jakąś ładną polską nazwę, ładny polski skrótowiec, bo na razie mimo tych zmian nadal jest to podatek antypolski. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie pośle. Kto z pań i panów posłów zgłosił się do zadania pytania? Czy są jeszcze chętni? Zamykam listę. Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W uzasadnieniu powołujecie się państwo, mówicie o uszczelnieniu systemu podatkowego, o gigantycznym postępie technologicznym w tym zakresie, że w gruncie rzeczy ten postęp umożliwia troszkę ułatwień, jeśli chodzi o rozliczenia podatkowe. Mam taką refleksję. Gdzie dzisiaj bylibyśmy, jak daleko mogłyby iść te ułatwienia, gdybyście państwo zrealizowali swoje własne plany, a także kontynuowali to, co w swoich założeniach wam swego czasu przygotowaliśmy? Mówię tu o rejestrze faktur on-line, rejestrze, który polegałby na uwierzytelnianiu faktur w rzeczywistym czasie na serwerze ministra finansów.

W ubiegłym roku usłyszałem, że prace trwają.

Pani poseł Krystyna Skowrońska, Koalicja Obywatelska. Szanowna Pani Marszałek! Pan poseł Cichoń panu ministrowi powiedział, jak po 3 mld zł miesięcznie wypływa z naszego budżetu i jak państwo lekką ręką zrobili takie koryto dla 200 mld zł, które wypłynęły z VAT-u.

Państwo umożliwiacie zapłatę niektórych zobowiązań. Namawiam pana ministra, aby uzgodnił również z Komisją Nadzoru Finansowego, aby klientowi można było przy wyliczaniu zdolności kredytowej wyliczać te środki, które ma na oddzielnym rachunku, bo to jest również przeszkoda, która utrudnia działanie przedsiębiorcom. Pani poseł Małgorzata Niemczyk, Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo! Jeśli mowa o VAT, należy poruszyć problem ulgi za złe długi. Problem każdej firmy, każdego przedsiębiorcy to problem braku płatności. Przedsiębiorcy narzekają. Ktoś nie płaci, uchyla się. To jest bardzo ważny problem. Kiedy skutecznie rząd PiS ten problem rozwiąże? Zatory płatnicze powodują efekt domina. Ulga za złe długi. Fiskus zdał sobie sprawę z tego problemu.

Proszę o pisemną informację, jak jest oceniane dzisiaj wprowadzenie tej ulgi i jaka jest efektywność tego przepisu? Ile wynosi w tej chwili umorzenie podatku z tego tytułu? Pan poseł Wojciech Saługa, Koalicja Obywatelska. Pani Marszałek!

Na 200 tys. spółek, które mogłyby z tego skorzystać, do końca maja zapisało się 360. Co się stało, panie ministrze? Czy to jest błąd tej ustawy? Bo my mówiliśmy, że jest zbyt skomplikowana. Czy przyznajemy się do tego, że jest to zbyt skomplikowane? Będziemy robić jakąś nowelę? Co dalej, panie ministrze, z tym estońskim CIT-em? Przepraszam, że przy ustawie o VAT, ale to bardzo ważny temat, bo to miało po prostu ułatwić pracę polskim przedsiębiorcom i otworzyć przedsiębiorcom szeroko wrota na świat. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan poseł Dariusz Olszewski, Prawo i Sprawiedliwość. Szanowna Pani Marszałek! Szanowny Panie Ministrze! Wysoki Sejmie! Dziękując za zmiany wprowadzane w ustawie, chciałbym zauważyć, że w dobie cyfryzacji i wprowadzania nowoczesności w wielu aspektach życia społecznego i gospodarczego zgodnie z wymogami i oczekiwaniami społeczeństwa XXI w. należy unowocześnić przepisy dotyczące odliczania podatku VAT od środków transportu, zwłaszcza od zakupu samochodów osobowych na cele działalności gospodarczej, i rozliczania kosztów ich użytkowania. Każda osoba prowadząca działalność gospodarczą powinna mieć swobodę w wyborze środka transportu, jaki uzna za najlepszy do wybranego przez siebie zakresu działalności, a jeśli jednocześnie jest płatnikiem podatku VAT, winna mieć prawo do pełnego rozliczania tego podatku z tytułu zakupu pojazdu i jego użytkowania. Krótkie pytanie: Czy i kiedy rząd przewiduje zmiany w sprawie przeze mnie poruszanej? Pan poseł Jan Szopiński, Lewica. Wysoka Izbo! Rząd zgodnie z projektem przewiduje przykładowo karanie polskiego podatnika za błędy powstałe po stronie dostawców, czyli wystawców faktur.

I przeciwnie: Czy w przypadku nadpłaty podatku VAT powstałego w wyniku błędnie wystawionej, a następnie skorygowanej faktury podatnik otrzyma rekompensatę ze strony Skarbu Państwa? Przedsiębiorcy z Kujaw i Pomorza pytają, jak mają się poruszać w gąszczu tak niezrozumiałych i nielogicznych dla zwykłego obywatela przepisów. I chciałbym też zapytać: Jak mikroprzedsiębiorstwa mogą zastosować się do proponowanych przepisów bez ponoszenia ogromnych (Dzwonek) kosztów na doradztwo podatkowe? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan poseł Dariusz Rosati, Koalicja Obywatelska.

Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Szczyci się pan, że projekt ustawy wychodzi naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, że upraszcza im życie. Chciałem w związku z tym zapytać: Czy zechciałby pan jeszcze pójść pół kroku dalej i np. skrócić termin zwrotu VAT z rachunków w ramach split payment z 30 dni do np. 15 dni? Słyszę o postępach, jeśli chodzi o cyfryzację resortu i aparatu skarbowego, a zatem być może to by się udało zrobić. Poddaję to pod rozwagę. I mam drugie pytanie związane z wielokrotnym informowaniem opinii publicznej przez premiera Morawieckiego o tym, że rząd PiS odebrał pieniądze mafiom VAT-owskim i przekazał na zbożne cele, np. na polskie dzieci. Chciałem pana zapytać: Ile tych pieniędzy odebrano mafiom VAT-owskim do dziś? Dziękuję bardzo, panie pośle. Pan poseł Krzysztof Grabczuk, Koalicja Obywatelska. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Wszelkie ułatwienia, które decydują o tym, że łatwiej będzie się prowadziło działalność gospodarczą, oczywiście będą przez nas popierane, zwłaszcza że okres pandemii w sposób szczególny temu sprzyja. Ale to jest wciąż za mało, panie ministrze, jeśli chodzi o łatwość prowadzenia działalności gospodarczej w naszym kraju w porównaniu z innymi krajami na świecie. W ostatnim okresie zamiast iść do góry, wciąż spadamy. Zachęcam państwa, abyście państwo poszli zdecydowanie dalej w tym zakresie. Cieszę się, że państwo wycofujecie się ze złych pomysłów, które wprowadziliście tutaj, w tej Izbie, ale znowu powtarza się ten sam mechanizm. Państwo nie chcecie słuchać opozycji, nie chcecie słuchać dobrych propozycji, które na tej sali się pojawiają. Gdybyście państwo słuchali, nigdy do takich sytuacji by nie dochodziło. Przyłączam się do tego apelu, bo państwo ciągle mówicie o mafiach VAT-owskich. Jedyna, którą państwo złapaliście, to ta, którą sami utworzyliście w Ministerstwie Finansów. Bardzo proszę, pokażcie państwo, jakie fundusze z tego tytułu trafiły do naszego budżetu. Również proszę o odpowiedź na piśmie. Teraz pan poseł Mirosław Suchoń, Polska 2050. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chciałem zapytać o terminy zwrotu podatku VAT w odniesieniu do poszczególnych kategorii, jeżeli chodzi o wielkość podatników. Bardzo bym prosił o to, aby pan minister poinformował Wysoką Izbę, jaki jest dzisiaj czas oczekiwania na taki zwrot - właśnie nie średni dla wszystkich podatników, ale w odniesieniu do poszczególnych grup podatników. Również bardzo proszę o przekazanie takiej analizy w formie pisemnej. Dziękuję bardzo. Teraz głos zabierze podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów pan Jan Sarnowski.

W pierwszych słowach chciałbym gorąco podziękować państwu posłom za poparcie dla tego projektu. Rzeczywiście jest to projekt przygotowany dla przedsiębiorców, na ich prośbę i po konsultacji z nimi. Rzeczywiście wraz z elektronizacją wiele obowiązków i terminów może zostać albo ograniczonych, albo przedłużonych.

Pojawiło się wiele pytań na temat przyspieszenia zwrotów, na temat tego, czy ta nasza elektronizacja nie mogłaby również do tego doprowadzić. Tydzień temu zakomunikowaliśmy wprowadzenie od stycznia przyszłego roku nowej kategorii podatnika, mianowicie podatnika bezgotówkowego.

Przechodząc do państwa pytań. Co do kwestii metody kasowej, czyli momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT dopiero w chwili otrzymania zapłaty, już teraz niektórzy przedsiębiorcy mogą korzystać z tej możliwości i nie jest to rozwiązanie, z którego chętnie korzystają. Pan poseł Cichoń pytał o dalszy los projektu „e-faktury” Tutaj spieszę z wyjaśnieniami. Prace nad tym projektem rozpoczęte zostały w końcu roku 2019, to już były prace legislacyjne mające na celu przelanie tej idei na język przepisów. Sam projekt uzyskał wpis do wykazu w grudniu zeszłego roku.

Co do kwestii poruszonej przez panią poseł Skowrońską, kwestii zdolności kredytowej w związku z środkami, które są na rachunkach VAT-owskich - ten temat również przeanalizujemy w Ministerstwie Finansów i damy odpowiedź na piśmie. W zakresie estońskiego CIT-u chciałbym gorąco przypomnieć, że możliwość skorzystania z tej opcji opodatkowania otwarta jest dla przedsiębiorców przez cały rok. Pierwszym jest ryczałt od dochodów spółek kapitałowych, a drugim rezerwa inwestycyjna wzorowana na rozwiązaniu niemieckim. Niemiecka rezerwa inwestycyjna to jest rozwiązanie, zgodnie z którym podatnicy deklarują skorzystanie z niego dopiero po zakończeniu roku podatkowego.

Już na etapie komunikowania estońskiego CIT-u mocno podkreślaliśmy, że naszym celem jest to, żeby rozwiązania proinwestycyjne były otwarte dla jak największej liczby przedsiębiorców, dlatego już od 1 stycznia przyszłego roku estoński CIT będzie zdecydowanie szerzej otwarty, nie tylko na spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i na spółki akcyjne, ale również na spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne oraz na spółdzielnie, przynajmniej w zakresie rezerwy inwestycyjnej. Co więcej, nie będzie już limitu przychodowego, czyli będzie on również otwarty dla większych firm średniego i dużego biznesu. Nie będzie również warunku inwestycyjnego. Realna stawka opodatkowania u małego podatnika spadnie i nie będzie podatku na wejściu, a to również mogło stanowić pewnego rodzaju element zniechęcający podmioty do tego rodzaju rozliczenia.

W zakresie dalszych pytań odnośnie do wykorzystania tego rodzaju środka częściowo do działalności biznesowej, a częściowo do działalności gospodarczej, również odpowiemy na piśmie, też co do dalszych kroków podejmowanych przez Ministerstwo Finansów. Tak samo, tak jak państwo posłowie prosili, odnośnie do terminu zwrotu VAT-u w zakresie kategorii poszczególnych przedsiębiorców w zależności od ich wielkości. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Marszałek Sejmu, po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu, proponuje, aby Sejm skierował rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo bankowe, zawarty w druku nr 1236, do Komisji Finansów Publicznych w celu rozpatrzenia. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycję przyjął. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 4. porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych (druk nr 1264) Proszę sekretarza stanu w Ministerstwie Cyfryzacji pana Adama Andruszkiewicza.

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Celem projektu ustawy o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych jest przesunięcie terminu wdrożenia systemu e-doręczeń oraz terminu, od którego organy administracji rządowej i centralnej oraz ZUS, KRUS i NFZ będą miały obowiązek korzystania z publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego, z publicznej usługi hybrydowej. Pierwszym i najważniejszym założeniem ustawy o doręczeniach elektronicznych jest to, że obywatel powinien mieć prawo do komunikacji elektronicznej z organami państwa i należy mu takie prawo zapewnić. Realizacją powyższego założenia jest zasada, zgodnie z którą, jeśli obywatel złoży deklarację, że chce otrzymywać korespondencję kierowaną do niego od państwa w sposób elektroniczny, to organy państwa będą w stanie mu to zapewnić. Ze względu na ten kluczowy cel wprowadzenia systemu e-doręczeń w Polsce istotne jest, by organy państwa, które będą go realizować, były dobrze przygotowane. Elementem niezbędnym do osiągnięcia stanu gotowości jest przeprowadzenie odpowiednich testów systemu i szkoleń urzędników. Trwający od ponad roku okres pandemii COVID-19 z jednej strony charakteryzuje się dynamicznym postępem cyfryzacji państwa prowadzonej przez administrację naszego rządu, z drugiej jednak powoduje konieczność szybkiego wdrażania nowych projektów niezbędnych do działań w zakresie minimalizacji skutków pandemii oraz wywołuje trudności z wdrażaniem systemów teleinformatycznych, w tym systemu e-doręczeń. Okres pracy zdalnej utrudnia dostosowanie stacji roboczych urzędników, m.in. rekonfigurację i doposażenie, wykonywanie szerokich testów nowego rozwiązania, jak również przeprowadzenie szerokich i efektywnych szkoleń przyszłych użytkowników systemu. Zarówno testy, jak i szkolenia użytkowników są natomiast elementem koniecznym do sprawnego wdrożenia systemu. Naszym obowiązkiem jest przy tym nie pośpiech, lecz przekazanie obywatelom sprawnej, sprawdzonej usługi doręczenia elektronicznego.

Zaproponowane zmiany mają na celu zapewnienie prawidłowego przygotowania administracji do realizowania tak ważnej dla obywateli usługi, jaką są e-doręczenia, oraz jednolite czasowe jej wprowadzenie przez jak największą grupę podmiotów publicznych. Przesunięcie terminu wejścia w życie ustawy o 3 miesiące oznacza wdrożenie bazy adresów elektronicznych oraz usług świadczonych przez operatora wyznaczonego po okresie wakacyjnym. Natomiast wydłużenie terminu obowiązku stosowania e-doręczeń przez pierwsze grupy podmiotów publicznych, które mają wejść w system, ma na celu ujednolicenie terminów dla administracji rządowej i pozostałej administracji centralnej. Ważne jest bowiem, by w pierwszym terminie do systemu weszła jak największa grupa podmiotów publicznych. Wydłużenie zaś okresu pomiędzy wejściem w życie ustawy a obowiązkiem jej stosowania pozwoli na przeprowadzenie szerokich testów i szkoleń dla użytkowników systemu, utrudnionych w okresie pandemii. W efekcie pozwoli to natomiast na bardziej sprawną obsługę obywateli. Mając na uwadze powyższe, wnoszę o przyjęcie rządowego projektu ustawy. Bardzo dziękuję, panie marszałku. Bardzo dziękuję. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół.

Pan poseł Witold Czarnecki, Prawo i Sprawiedliwość, w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość przedstawić stanowisko mojego klubu w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych, druk sejmowy nr 1264. Celem projektu ustawy o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych jest przesunięcie terminu wdrożenia systemu e-doręczeń oraz terminu, od którego organy administracji rządowej i centralnej oraz ZUS, KRUS i NFZ będą miały obowiązek stosowania e-doręczenia. Kluczowe jest, by organy państwowe, które będą realizować e-doręczenia, były dobrze przygotowane. Jak wskazano w uzasadnieniu projektu, bardzo ważnym elementem osiągnięcia stanu gotowości jest przeprowadzenie odpowiednich testów systemu i szkoleń urzędników. Pandemia COVID-19, która trwa już ponad rok, powoduje duże trudności we wdrażaniu wielu systemów teleinformatycznych, w tym również systemu e-doręczeń. Okres pracy zdalnej utrudnia również techniczne dostosowanie sprzętu, systemów informatycznych, a także przeprowadzanie testów nowego rozwiązania, jak również przeprowadzenie szkoleń dla użytkowników systemu e-doręczeń. Zaproponowane przesunięcie terminu wejścia w życie ustawy o 3 miesiące, a także zmiana terminu, od kiedy trzeba będzie stosować e-doręczenia, dla administracji rządowej o 9 miesięcy, a dla administracji centralnej oraz ZUS, KRUS i NFZ - o 6 miesięcy oraz, jak się wydaje, skuteczne wychodzenie z pandemii COVID-19 umożliwią odpowiednie przygotowanie administracji do zrealizowania tak ważnych dla obywateli usług, jakimi są e-doręczenia. Zyskany czas pozwoli również na przeprowadzenie testów i szkoleń, których organizacja była utrudniona w okresie pandemii. Mając powyższe na uwadze, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość pozytywnie ocenia i popiera przedstawiony projekt rządowy. Równocześnie składam na ręce pana marszałka wniosek o przejście do drugiego czytania. Dziękuję. Pan poseł Michał Gramatyka, Koalicja Obywatelska.

Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W zasadzie od początku prac legislacyjnych było wiadomo, że polski rząd nie jest gotowy na wdrożenie tego gigantycznego systemu, nowego systemu, systemu przełomowego, co warto przyznać, systemu doręczeń elektronicznych. Tym bardziej że narzucono jako dostawcę usługi Pocztę Polską. Nie zdążycie z rejestrem podmiotów niepublicznych, przesuwacie to o kolejne miesiące. Nie zdążycie z gotowością na przyjmowanie elektronicznych pism przez organy rządowe - to też ulega przesunięciu o kolejne miesiące. Ustawa umarza postępowania administracyjne, które już się toczą przed Urzędem Komunikacji Elektronicznej. Na szczęście dotykacie również art. 9, który zobowiązuje do zakładania skrzynek w systemie przedstawicieli wolnych zawodów prawniczych, ale nie tylko prawniczych.

Specjaliści liczą, że to ok. 0,5 mld w skali roku - ukryty podatek, który obciąży samorządy, polskich przedsiębiorców, bo ich jako pierwszych dotknie wasz pomysł na powszechną cyfryzację. I to właśnie dlatego apelowaliśmy podczas prac legislacyjnych, że warto wyłonić operatora elektronicznych doręczeń na konkurencyjnym rynku. Dziś sytuacja wygląda tak, że prywatne firmy za elektroniczne listy polecone życzą sobie ok. złotówki. Ale taki jest efekt promowania na siłę państwowego molocha, który zresztą zgodnie z ostatnim raportem Najwyższej Izby Kontroli ma bardzo poważny problem z przetwarzaniem danych osobowych Polek i Polaków bez podstawy prawnej. Taki jest prawdziwy obraz cyfrowej Polski według PiS. Minister przechowuje na prywatnej skrzynce rządowe dokumenty, a potem się dziwi, że ktoś mu się włamuje na tę skrzynkę. Szefem resortu cyfryzacji zostaje polityk, który jest zamieszany w niejasne finansowo dostawy maseczek i respiratorów, również w czasie COVID-u, tego samego, który zatrzymał wdrożenie ustawy o doręczeniach elektronicznych. A poseł, który składa oświadczenie majątkowe poprzez rządową platformę gov.pl, dowiaduje się w polskim Sejmie, że polski Sejm nie przyjmie mu takiego oświadczenia majątkowego, bo polski Sejm gov.pl nie widzi, mimo że jest w Polsce i że jest polskim Sejmem. Co chwilę kolejni znani politycy padają ofiarą hakerskich ataków, najczęściej na prywatne skrzynki pocztowe, bo i państwo, i ja wiemy, że te rządowe czy sejmowe są świetnie zabezpieczone, a CERT-ABW robi bardzo dobrą robotę. Ale opinia publiczna nie dowie się o karkołomnej wręcz niefrasobliwości polityków, bo Sejm zdecydował o utajnieniu posiedzenia poświęconemu temu tematowi. Jedno wychodzi wam świetnie, to jest gromadzenie danych o Polkach i Polakach bez ich wiedzy, bez ich zgody, bez wpływu, pod każdym możliwym pozorem: pandemia, opłaty za drogi, spis rolny, spis powszechny, podatek VAT itp. Kompletnie bez umiaru. W swoim ostatnim niemal gierkowskim planie 5-letnim nazywacie to Cyber Poland, zupełnie nie wiadomo dlaczego po angielsku. Polska nazwa: Cyfrowy Chaos, byłaby chyba dużo bardziej stosowna. Pan poseł Robert Kwiatkowski, klub Lewicy, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Otrzymaliśmy do rozpatrzenia druk nr 1264 o nowelizacji ustawy o doręczeniach elektronicznych. Pierwsza refleksja, jaką mam panie marszałku, to taka, że chyba doszło do jakiejś literówki. Myśmy dostali ten druk do przeczytania wczoraj o godz. 18.28, nie minęło 20 godzin, a już Wysoka Izba rozpatruje to przedłożenie rządowe.

Wydaje się, że nie wpływa to - mówiąc szczerze - na zwiększenie autorytetu Wysokiej Izby, nie wpływa też na polepszenie jakości prac, na co pewnie przede wszystkim powinniśmy zwrócić uwagę. I to jest, panie marszałku, pierwszy powód, dla którego klub Lewicy będzie głosował za odrzuceniem tego rządowego przedłożenia już w pierwszym czytaniu. W uzasadnieniu tego przedłożenia czytamy o przesunięciu wprowadzenia w życie tej usługi - usługi doręczeń elektronicznych - która, przypomnę, ma ostatecznie zostać wdrożona do końca 2029 r. Potrzebne są poszczególne przesunięcia, ponieważ - uwaga - rząd nie spodziewając się, a może nie doceniając znaczenia i skutków pandemii, musi przesunąć szkolenia i testy. Naprawdę? Przesunąć szkolenia i testy dotyczące tej usługi w sytuacji, w której borykając się ze skutkami pandemii, uporali się z tym hotelarze, gastronomia, szkoły, kościoły? Wszyscy, tylko nie rząd. Przesunięcie tego o 4 do 8 miesięcy - panie ministrze, chyba mówimy o takich liczbach - pan minister był uprzejmy skomentować, czy uzasadnić, w taki oto sposób, że obywatel ma prawo do tej usługi.

To jest drugi powód. Trzeci jest związany z tym, co czeka nas jutro. Jutro będziemy na tajnym posiedzeniu dyskutować, a może tylko wysłuchiwać informacji o cyberzagrożeniach. Mówimy w tej chwili o doręczeniach elektronicznych, które mają być pod kontrolą państwa, bezpieczne, godne zaufania, nadzorowane przez właściwe organy państwa. Czy nie widzicie państwo związku między jednym a drugim?

Przecież absurd tego przedłożenia rządowego w połączeniu z jutrzejszym tematem nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu aż bije w oczy. Czwarty powód jest związany z operatorem wyznaczonym do świadczenia tej usługi, czyli mówiąc po polsku i po ludzku, z Pocztą Polską. Poczta Polska nie wyrobiła się z testami, nie wyrobiła się ze szkoleniami.

Za to Poczta Polska ma czas na organizację wyborów kopertowych, na spory zbiorowe z pracownikami, których w skali masowej się zwalnia, na prowadzenie sklepików z dewocjonaliami i artykułami spożywczymi, i czym tam jeszcze. Na wszystko Poczta Polska, reprezentowana przez zarząd, ma czas, tylko nie ma czasu na zajęcie się usługą, która decydować będzie o być albo nie być tej instytucji, tej firmy, która niedługo będzie obchodziła 500-lecie. Tak, tak - 500-lecie. Ale jeśli ona jest w takich rękach, w jakich znajduje się obecnie, to czarno widzę nie tylko świętowanie tej rocznicy, ale w ogóle przyszłość tej zasłużonej instytucji, jakże potrzebnej w codziennym życiu (Dzwonek) Polek i Polaków. Reasumując, wnosimy o odrzucenie tego przedłożenia już w pierwszym czytaniu.

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe, Unia Europejskich Demokratów, Konserwatyści mam zaszczyt przedstawić nasze stanowisko w sprawie zmiany ustawy o doręczeniach elektronicznych. Głównym celem proponowanej zmiany jest przesunięcie terminów wdrożenia publicznej usługi rejestrowego doręczenia elektronicznego oraz publicznej usługi hybrydowej w celu zapewnienia jak najwyższej jakości dla użytkowników końcowych.

Zasłanianie się COVID-19 może jest zasadne, lecz właśnie okres pandemii pokazał, jak ważna jest cyfryzacja naszego kraju i jak ważne jest to, aby obywatele mogli doręczać pisma i korzystać z dobrodziejstw cyfryzacji. Natomiast my nie potrafimy wprowadzić tej ustawy.

Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan poseł Janusz Korwin-Mikke, koło Konfederacja. Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Proszę państwa, pamiętam czasy, kiedy pan Aleksander Kwaśniewski, późniejszy prezydent Polski, był jako młody komunista w komisji, która przygotowywała warunki komunizacji Polski.

W odróżnieniu od mojego przedmówcy, posła Koalicji Polskiej, czyli PSL, jak rozumiem, ja się nie boję, że nam zajrzy Huawei, bo Huawei nie ma do nas pretensji granicznych ani też nie prowadzi imperialnej polityki w Europie.

To jest dziwne, bo Lewica zawsze popiera zdzieranie pieniędzy przez państwo od prywaciarzy a tutaj, proszę, dopuściła takie rzeczy.

Nie bardzo rozumiemy, dlaczego nie można tego zrobić szybko.

Nie mogą zrozumieć, bo prywatne koncerny mają lepszych informatyków i tam postęp galopuje, a rządy z najwyższym trudem za nim nadążają albo w ogóle nie nadążają. Jeżeli będą to robili nasi eksperci, to z przykrością oznajmiam.

Dziękuję za uwagę. Pani poseł Hanna Gill-Piątek, koło Polska 2050. Wysoka Izbo! Polska 2050 poparła ustawę o doręczeniach elektronicznych, nad którą pracowaliśmy w zeszłym roku. Dziś rząd przedkłada nam projekt, w którym znacznie opóźnia się wprowadzenie tych rozwiązań w życie. Przypomnę, że ustawa ta miała nas przenieść z ery papieru do nowoczesnego świata, w którym bez naklejania znaczków i kolejek na poczcie możemy z instytucjami wymieniać korespondencję tanio, ekologicznie, pewnie i szybko za pomocą narzędzi współczesnej komunikacji. Dla tych, którzy z różnych powodów nie mogli korzystać z dobrodziejstw cyfryzacji, wymyślono przesyłkę hybrydową, drukowaną na poczcie i wkładaną do skrzynki, bez kosztownego transportu, bez zbytecznego czekania. Dziś mówicie ludziom, że nie dacie rady wdrożyć tego, co od lat w Polsce powinno być standardem, że potrzebujecie jeszcze kilka długich miesięcy i że to według oceny skutków regulacji będzie kosztowało obywateli 24 mln zł. Rozumiemy, że to przez epidemię, ale to już niestety reguła, że w wygodnych i potrzebnych wam politycznie sprawach działacie błyskawicznie, a w usprawnianiu państwa zawsze macie czas na zwłokę. A takiego państwa dziś oczekują od nas obywatele, co jako Polska 2050 doskonale wiemy, rozmawiając z nimi w całej Polsce - państwa sprawnego, państwa nowoczesnego, o wysokim poziomie usług publicznych. Po ostatnich wydarzeniach nasuwa się jeszcze jedno pytanie: Czy pomimo wydłużenia czasu jesteście w stanie zapewnić temu systemowi bezpieczeństwo? To przecież ważne sprawy urzędowe Polek i Polaków, które nie powinny dostać się w niepowołane ręce.

Poczcie, która współpracuje z ok. 1 tys. prywatnych podmiotów prowadzących agencje pocztowe, do których trafi nasza korespondencja w przypadku przesyłek hybrydowych, ale tym razem już nie w zamkniętych kopertach. Mam nadzieję, że lepiej niż korespondencja rządowa. Nie można jednak zapomnieć, że operator doręczeń elektronicznych, Poczta Polska, wciąż nie wyjaśnił, co stało się z bazą danych PESEL przekazanych jej przez Ministerstwo Cyfryzacji w marcu poprzedniego roku, przy nieudanych wyborach kopertowych, dodajmy, przekazanych bezprawnie. Podsumowując, Polska 2050 na pewno nie poprze waszych opóźnień, za które zwykli obywatele zapłacą 24 mln zł. Pozostaje otwarte pytanie, czy będzie to system bezpieczny i czy w ogóle rząd jest w stanie sprostać temu zadaniu, czyli zabezpieczyć naszą korespondencję, skoro nie potrafi zabezpieczyć własnej.

Pan poseł Michał Gramatyka, Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo! Art. 9 ustawy o doręczeniach elektronicznych zobowiązuje pewną bardzo szeroką grupę wolnych zawodów do zakładania skrzynek do doręczeń już od października tego roku, w obecnie obowiązującym stanie prawnym. Oczywiście to jest dzisiaj niemożliwe, dlatego że Poczta Polska nie udostępnia, nie daje takiej możliwości, i pewnie nie udostępni do końca roku. Każdy z tych podmiotów dzisiaj może za darmo dostarczać korespondencję do wszystkich organów administracji rządowej z wykorzystaniem platformy gov.pl. Kto zrekompensuje koszty poniesione przez te wolne zawody w momencie, kiedy wasza ustawa wejdzie w życie?

Pan poseł Jan Szopiński, klub Lewicy. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W ramach nowej usługi każdy obywatel ma dostać darmową skrzynkę mailową. Niestety doręczenie darmowe już nie będzie, wszystkie instytucje wysyłające listy płacą 4,30 zł.

Nie wiem, czy ze strony rządu jest to rekompensata wydatków poniesionych na wybory kopertowe, ale pierwszy raz słyszę, aby dostarczenie maila było droższe od wysłania tradycyjnego listu. Przypomnę jedynie, że takie firmy jak Google czy Microsoft świadczą usługi szerzej, szerzej są one zakrojone i są zupełnie bezpłatne. Mam takie pytanie: Czy Poczta Polska po tym, jak weszła w buty Państwowej Komisji Wyborczej i zajęła się organizacją wyborów, tym razem dostała zadanie zorganizowania systemu e-doręczeń?

Panie Ministrze! Cyfryzacja jest koniecznością. Okres pandemii pokazał, jak wiele mamy do zrobienia w tym zakresie. Ale nie w ten sposób. Nie może być takiej sytuacji, że projekt ustawy pojawia się w ostatniej chwili. Jest tam bardzo dużo zapisów, nie można nad tym w ostatniej chwili procedować. Drugi element. Państwo cały czas zbieracie dane od różnych instytucji, od różnych osób. Co się z tym w przyszłości stanie?

Będą fruwały do różnych niepożądanych osób. Ostatnia rzecz.

Polska 2050. Szanowni Państwo! Wysoka Izbo!

Bardzo proszę o poinformowanie, ilu pracowników miało zostać przeszkolonych, ilu do dnia dzisiejszego przeszkolono, ilu zostało do przeszkolenia, kto był odpowiedzialny i jakie konsekwencje zostały wyciągnięte w stosunku do osób, które dopuściły (Dzwonek) do takiego rażącego zaniedbania w tej ważnej dziedzinie.

Panie Ministrze! Dlaczego fundujecie Polakom najdroższy model dostarczania wiadomości elektronicznie?

Czego zatem państwo próbujecie, jeżeli nakładacie obowiązki na przedsiębiorców? Jeżeli nakładacie na określone grupy dodatkowe obowiązki, to państwo nie martwicie się o ich koszty. Jeżeli ustalacie dla Poczty Polskiej wysokość tej opłaty, to kalkulacja, chcemy wam powiedzieć, jest zła. Nie pamiętam, ile mają Węgry. Ale proszę nie mówić, że... Fundujecie nam najdroższe (Dzwonek) elektroniczne doręczenie. Głos zabierze sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji pan Adam Andruszkiewicz.

Szanowny Panie Marszałku!

To jest w ogóle niepoprawne nazywanie tej usługi, która jest bardzo wysoko zaawansowaną usługą korespondencji pomiędzy obywatelem a instytucjami państwa.

Tak że tutaj w żaden sposób nie narażamy obywateli na wypłynięcie żadnych danych.

Szanowni Państwo! Bardzo dziękuję. Zamykam dyskusję. W dyskusji zgłoszono wnioski: o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu oraz o przystąpienie niezwłocznie do drugiego czytania. Do głosowania nad tymi wnioskami przystąpimy w bloku głosowań. Ogłaszam przerwę do godz. 14.45.

Wznawiam obrady. Obecnie, proszę państwa, przystąpimy do stwierdzenia kworum. Bardzo proszę o naciśnięcie dowolnego przycisku w celu potwierdzenia obecności na posiedzeniu.

posiedzeniu bierze udział 453 posłów. Stwierdzam kworum. Właściwe komisje przedłożyły sprawozdanie o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw, druk nr 1260. W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, podjęłam decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący rozpatrzenie tego sprawozdania. Proponuję, aby w tym przypadku Sejm wyraził zgodę na skrócenie terminu, o którym mowa w art. 54 ust. 5 regulaminu Sejmu. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Prezydium Sejmu, po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów, przedłożyło wniosek w sprawie zmian w składach osobowych komisji sejmowych, druk nr 1265. W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, podjęłam decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący rozpatrzenie tego wniosku.

Powracamy do rozpatrzenia punktu 4. porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych. W dyskusji zgłoszono wnioski: o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu oraz o przystąpienie niezwłocznie do drugiego czytania. W pierwszej kolejności poddam pod głosowanie wniosek o odrzucenie projektu ustawy. Jego odrzucenie oznaczać będzie, że Sejm wyraził zgodę na przystąpienie niezwłocznie do drugiego czytania, bez odsyłania projektu ustawy do komisji. Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych, zawartego w druku nr 1264, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm wniosek odrzucił, a tym samym wyraził zgodę na przystąpienie niezwłocznie do drugiego czytania projektu ustawy. Przystępujemy do drugiego czytania projektu ustawy. Czy ktoś z pań i panów posłów pragnie zabrać głos w drugim czytaniu tego projektu ustawy? Proponuję, aby Sejm wysłuchał 2-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół, jeżeli takie będą. Proszę bardzo, panie pośle. Słabo słyszę, pani marszałek, przepraszam. Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość składam wniosek o przystąpienie do trzeciego czytania rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych bez odsyłania do komisji poprawek i wniosków zgłoszonych do tego projektu ustawy i po doręczeniu ich posłom.

Wysoka Izbo!

Nie jesteście w stanie zrealizować zobowiązań, które sami na siebie nakładacie. Przecież to są wasze terminy, wasze propozycje i okazuje się, że obywatele nie mogą skorzystać z ustawy, która zresztą - uwaga - wejdzie w całości w życie dopiero pod koniec 2029 r. Ale po drodze trzeba, drodzy państwo, wykonać normalną, codzienną urzędniczą pracę. Musi pracować ministerstwo cyfryzacji, zresztą przez was zlikwidowane.

Ano dlatego, że była pandemia. W całej Polsce pandemia przeszkodziła, ale nie przeszkodziła w wykonywaniu pracy, nie przeszkodziła w otwieraniu hoteli, gastronomii, ba, kościołów, tylko wam przeszkodziła w tym, żeby wykonać normalne urzędnicze obowiązki, żeby - jak to napisano, pani marszałek, Wysoki Sejmie, w uzasadnieniu - doprowadzić do tego, żeby były przeprowadzone testy, żeby przeszkolono ludzi, którzy mają się zajmować tymi doręczeniami. Wszystkiego tego zabrakło. Moi Drodzy! Czym wy się zajmujecie? My za chwilę, już jutro będziemy in pleno rozmawiać o zagrożeniach cyberatakami, o cyberbezpieczeństwie. Przecież doręczenia elektroniczne to jest forma nowoczesnego zabezpieczenia obrotu dokumentów. Nie widzicie związku między jednym a drugim? Poczta Polska prowadzi rozliczne działania, zastępując Państwową Komisję Wyborczą.

Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Głosowaliśmy zresztą za tą ustawą w momencie, kiedy ona była poprzednim razem procedowana. Ale teraz, kiedy okazało się, że po raz kolejny nie daliście rady, w dodatku obdarzacie Polki i Polaków doręczeniami elektronicznymi, w przypadku których mail będzie kosztował ok. 3,75 zł. I nie wiadomo, kto te koszty poniesie, bo tak naprawdę pojawia się kolejny parapodatek, który dotknie nas wszystkich, którzy będą chcieli komunikować się z organami administracji rządowej w sposób elektroniczny, co dzisiaj, co warto podkreślić, jest darmowe. Może to jest czas, żeby przy okazji uświadomić ministrów waszego rządu, że nie należy trzymać służbowej korespondencji w prywatnych, otwartych i darmowych skrzynkach pocztowych, bo potem pojawiają się z tego powodu różne niespodzianki, o których nie wolno podobno dyskutować w sposób jawny, tylko trzeba taką dyskusję utajnić, zupełnie nie wiadomo dlaczego. Nigdy nie jest za późno na dobrą dyskusję o bezpiecznej i odpowiedzialnej cyfryzacji. Porozmawiajmy na temat rozwiązań tej ustawy na łonie odpowiedniej komisji. Proszę bardzo, pani poseł Hanna Gill-Piątek, Polska 2050. Wysoka Izbo! Tak jak już podkreślałam w poprzednim wystąpieniu, ten druk jest przepychany przez Sejm kolanem. O ile jako Polska 2050 byliśmy jak najbardziej za rozwiązaniami dotyczącymi doręczeń elektronicznych, bo to powinno być dawno w Polsce standardem. To jest standard sprawnego i nowoczesnego państwa, którego jeszcze w Polsce cały czas nie mamy i poczekamy na nie kolejne 9 miesięcy, ponieważ chcecie to odłożyć. Przerzucacie te koszty na obywateli, którzy będą czekać na tanie, nowoczesne i sprawne państwo jeszcze dłużej. To jest po prostu coś niesamowitego. Na pewno będziemy się sprzeciwiać temu, żeby przejść od razu do trzeciego czytania. To jest po prostu coś, czego nie możemy tutaj zaakceptować. I bardzo proszę, żeby tego typu praktyki były w tym Sejmie jak najrzadsze, żeby ich w ogóle nie było. Co to jest, żeby pchać taki druk kolanem przez Sejm w ciągu jednej doby? Proszę. Wysoka Izbo! Najlepsze, co wynosimy z tej całej tragedii COVID-owej, tragedii gospodarczej, tragedii zdrowotnej, jest to, że cyfryzacja państwa, gospodarki przyspieszyła. Okazało się nagle, że masa urzędów może załatwiać elektronicznie, może załatwiać na telefon, może załatwiać bez konieczności stania i przynoszenia dziesiątków papierków rzeczy, których wcześniej nie można było załatwić, które wcześniej były nie do załatwienia inaczej niż tylko poprzez osobiste wielokrotne stawiennictwo.

To jest sedno sprawy. To, co państwo proponują, niestety tego nie rozwiązuje.

To jest sklonowanie po raz kolejny czegoś, co nie działa, po prostu nie działa. Co więcej, państwo tę sprawę przynosicie za pięć dwunasta. Przepychacie w wariackim trybie w Sejmie sprawę, którą spokojnie można było zrealizować już dawno. Co to w ogóle jest? Przestańcie, skończcie z tym dziadostwem legislacyjnym i skończcie z tym dziadostwem, jeśli chodzi o zarządzanie państwem polskim. Naprawdę. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Przystępujemy do trzeciego czytania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku.

Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 1264, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał?

Przypominam, że był wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu. Powiedziałam, że w pierwszej kolejności poddam pod głosowanie ten wniosek, a jego odrzucenie oznaczać będzie, że Sejm wyraził zgodę na przystąpienie niezwłocznie do drugiego czytania bez odsyłania projektu ustawy do komisji.

Powracamy do rozpatrzenia punktu 1. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Dodatkowe sprawozdanie komisji to druk nr 1254-A. Proszę panią poseł Annę Paluch o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji. Dziękuję bardzo. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W drugim czytaniu rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko złożono do tego projektu cztery poprawki.

Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 1243. Komisja przedstawia również w dodatkowym sprawozdaniu poprawki, nad którymi głosować będziemy w pierwszej kolejności. Poprawki 1. i 2. zgłoszone zostały do art. 1 ustawy nowelizującej zawierającego zmiany do ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki.

Sejm poprawkę odrzucił. Z poprawką tą łączy się poprawka 3. Nad nimi głosować będziemy łącznie.

Sejm poprawki odrzucił. W 4. poprawce do art. 2 projektu ustawy nowelizującej wnioskodawcy proponują, aby przepis ten dotyczył postępowań wszczętych i niezakończonych prawomocną decyzją. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawki 4., zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Sejm poprawkę odrzucił. Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 1243, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Proszę. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska chciałam zgłosić wniosek formalny o przerwę po to, by posłanki i posłowie mogli wsłuchać się w głos protestujących pielęgniarek i położnych. protestujących ratowników medycznych, protestujących z wszystkich środowisk medycznych, [[Oklaski]] którzy od wielu dni mówią: mamy dość, którzy od wielu dni mówią: mamy dość przeciążenia pracą, niskich pensji, braku dialogu z ministrem zdrowia i ignorancji rządu. Posłowie PiS-u, Solidarnej Polski i Porozumienia Gowina! Przed głosowaniem, proszę, zwróćcie uwagę na protestujących medyków, którzy od ponad roku walczą na pierwszej linii frontu z pandemią ponad swoje siły, narażając swoje zdrowie i życie. Dziś w upale walczą o słuszne podwyżki, o godziwą płacę. Walczą o lepsze warunki pracy. Dziś pielęgniarki i ratownicy medyczni pracują za pięć osób, na kilku etatach, w stresie, w przeciążeniu, z narażeniem swojego zdrowia i życia. Wysoka Izbo!

Pani poseł... ...wniosek formalny o przerwę, głosujemy nad nim.

Kto się wstrzymał?

Wniosek nie został przyjęty. Wysoka Izbo! Składam wniosek formalny o odroczenie obrad, tak aby przedstawiciele rządu, w tym przede wszystkim Ministerstwa Zdrowia, mogli odbyć spotkanie z przedstawicielkami pielęgniarek i położnych, które protestują przed Sejmem. One domagają się jednego: żeby poprzeć wszystkie poprawki Senatu. Chodzi przede wszystkim o to, żeby docenić ich ciężką pracę, ale również wykształcenie i doświadczenie zawodowe, żeby mogły otrzymać godną płacę za swoją pracę.

Sejm wniosek odrzucił. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 5. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Zdrowia o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1257 i 1260) Proszę pana posła Bolesława Piechę o przedstawienie sprawozdania komisji.

Sprawozdanie dotyczy uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw.

Co to znaczy? To znaczy. Niech pan nie krzyczy. Jest pan młodszy, uszanuj pan też trochę wiek. Chciałem powiedzieć jedno.

Skutki tego: 8, 16, 20 mld zł. W programie, w ogólnopolskiej debacie politycznej senator opozycji wskazał źródło finansowania: wystarczy wstrzymać, zawiesić, opóźnić realizację programu 500+. Jest moja głęboka niezgoda jako lekarza, jako posła i jako zwykłego obywatela, żeby za uchwały Senatu płaciły polskie dzieci. Przypominam, że Sejm odrzuca poprawki Senatu bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Jeżeli Sejm nie odrzuci poprawki Senatu, uważa się ją za przyjętą. Głosować będziemy nad wnioskami o odrzucenie poprawek Senatu. W 1. poprawce Senat proponuje dodać art. 3b do ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Głosujemy.

Sejm odrzucił poprawkę bezwzględną większością głosów. Komisje wnoszą o jej odrzucenie. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 2. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Sejm odrzucił poprawkę bezwzględną większością głosów.

Szanowni Państwo! Mam nadzieję, że one też wyjaśnią pewną perspektywę, którą zaproponowaliśmy w tej ustawie. Otóż w momencie gdy dochodziliśmy do apogeum trzeciej fali i zdawaliśmy sobie sprawę, że następuje przesilenie, liczba zakażeń powoli zaczyna spadać, pierwszym krokiem, pierwszym ruchem, który chcieliśmy wykonać względem środowiska sektora medycznego, było przygotowanie projektu ustawy o najniższych wynagrodzeniach. To był pierwszy ruch pandemiczny związany z wynagrodzeniami. Te głosy, które tutaj się pojawiają, że nie rozmawiamy, nie prowadzimy dialogu, są głosami po prostu nieprawdziwymi.

rozmawialiśmy o tym, jak kształtować wynagrodzenia. Oczywiście to nie były proste rozmowy, to nie były rozmowy, które kończyły się wspólnymi wnioskami, ale zdecydowaliśmy się na podzielenie tych ruchów płacowych na dwa kroki. Pierwszy krok, który ma polegać na tym, że przyspieszamy i zwiększamy poziom minimalnego wynagrodzenia w roku 2021, bo do tej pory rozwiązanie ustawowe oznaczało, że podwyżki najniższego wynagrodzenia miały być w grudniu. My to przesunęliśmy od 1 lipca, a po drugie, podwyższyliśmy wskaźniki. Koszt tej operacji i kwoty, które realnie skierujemy na wynagrodzenia, m.in. pielęgniarek, to jest 4 mld zł. Ale to absolutnie nie kończy rozmów. W międzyczasie zaprezentowana została koncepcja Nowego Polskiego Ładu, w którym padła deklaracja 7% PKB z przeznaczeniem na system opieki zdrowotnej. I to jest realna deklaracja, która oznacza poprawę względem dotychczasowej ścieżki, w ramach której mieliśmy realizować ten cel w postaci 6% PKB. Sytuacja wygląda tak, że drugim etapem rozmów po przyjęciu tej ustawy w pierwotnym kształcie ma być kontynuacja rozmów dotyczących najniższych wynagrodzeń, które mają zagwarantować wszystkim przedstawicielom zawodów w środowisku medycznym partycypację, czyli udział w tych zwiększających się nakładach. I chcemy zdefiniować, zbudować ścieżkę wzrostu najniższych wynagrodzeń do roku 2027, do którego mamy zrealizować ten cel w postaci wzrostu nakładów do 7% PKB. Szanowni Państwo! To głosowanie będzie pokazywało, czy zachowujemy się odpowiedzialnie z jednej strony, czy rzucamy puste obietnice. Ta odpowiedzialność to jest gwarancja wzrostu o 4 mld w ciągu pół roku. nakładów na wynagrodzenia w systemie opieki zdrowotnej, czyli 8 mld zł skutku rocznego. To, co znalazło się w poprawkach Senatu, które dosyć arbitralnie podwyższyły o 30% wskaźniki. to jest obietnica bez pokrycia. Roczny koszt to jest 12 mld zł. Szanowni państwo, jednorazowo 12 mld zł rocznie. To jest obietnica bez pokrycia. To jest szalenie ważne głosowanie i namawiam wszystkich państwa do odpowiedzialnego wyboru, a nie składania obietnic bez pokrycia. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 3. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Dawno się państwo nie widzieliście, widzę, i tu taka konwersacja się toczy z jednej strony, ale proponuję przenieść to po głosowaniach potem w kuluary.

Sejm odrzucił poprawkę bezwzględną większością głosów. Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 6. porządku dziennego: Powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich (druki nr 1223, 1224 i 1235) Zgodnie z art. 209 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 3 ust. 1 ustawy o Rzeczniku Praw Sejm powołuje rzecznika praw obywatelskich za zgodą Senatu. Grupy posłów zgłosiły następujące kandydatury na stanowisko rzecznika praw obywatelskich: panią Lidię Staroń oraz pana Marcina Wiącka. W imieniu grupy posłów z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość kandydaturę pani Lidii Staroń przedstawi pani poseł Barbara Bartuś. Bardzo proszę. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Pani Lidia Staroń jest inżynierem budownictwa, przedsiębiorcą, m.in. pełniła funkcję prezesa firmy handlowo-usługowej, a od 2005 r. zarządzała nieruchomościami. W 2005 r. pani Lidia Staroń uzyskała mandat poselski w okręgu olsztyńskim. W wyborach parlamentarnych w 2007 r. skutecznie ubiegała się o reelekcję, a w wyborach 2011 r. po raz trzeci z rzędu została wybrana na posła z wynikiem ponad 16 tys. głosów. W październiku 2015 r. pani Lidia Staroń uzyskała mandat senatorski, uzyskując go z własnego komitetu wyborczego Lidia Staroń - Zawsze po stronie ludzi.

Jest jedynym parlamentarzystą w Polsce, który zasiada w parlamencie wyłącznie z mandatu wyborców, bez żadnego poparcia formacji politycznych. W Senacie jest wiceprzewodniczącą Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz wiceprzewodniczącą Komisji Ustawodawczej. Jest członkiem Rady do spraw Pokrzywdzonych Przestępstwem, a także ekspertem zespołu ds. zmian ustawy o komornikach sądowych i egzekucji przy ministrze sprawiedliwości. Pani Lidia Staroń od lat skutecznie walczy z korupcją i z przejawami patologii w życiu społecznym. Jest założycielką i prezesem Stowarzyszenia Obrony Spółdzielców. W maju tego roku pani senator złożyła w Senacie projekt nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych poparty przez wszystkie siły polityczne, którego zapisy znacząco polepszą sytuację spółdzielców. W Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej pani Lidia Staroń przez trzy kadencje była członkiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. W VII kadencji pracowała też w Komisji Ustawodawczej oraz pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego. Trybunał potwierdził wtedy niekonstytucyjność przepisów obowiązującej wówczas ustawy. Pani Lidia Staroń zainicjowała zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego m.in. w zakresie egzekucji. Jest autorką zmian ustawy o komornikach sądowych i egzekucji dotyczących m.in. obniżenia opłat komorniczych oraz nagrywania czynności komornika. Doprowadziła do zwiększenia dostępu do pomocy prawnej i wzmocnienia pozycji ofiar przestępstw, w tym zwiększyła uprawnienia osób pokrzywdzonych przestępstwem. Od lat walczy o nowe przepisy zapewniające realną ochronę przed lichwą. Przygotowała pakiet zmian, w tym zmianę ustawy o kredycie konsumenckim, w której radykalnie zmniejszono główną granicę kosztów pozaodsetkowych, a także nowelizację prawa o notariacie zakładającą m.in. wymóg nagrywania czynności notarialnych. Oprócz przepisów pani Lidia Staroń interweniowała w Prokuraturze Krajowej w sprawie lichwy, a efektem interwencji było polecenie wszystkim prokuratorom, aby pomagali ofiarom lichwy także na drodze cywilnej. Pani Lidia Staroń walczy o niezakłamywanie historii, wskazując na potrzebę prowadzenia polityki historycznej i wyeliminowania nieprawdziwych, krzywdzących określeń: polskie obozy śmierci, polskie obozy koncentracyjne czy polskie obozy zagłady.

Jest autorką podjętej przez aklamację w 2015 r. uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zmieniającej nazwę Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych. i Obozów Zagłady na Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady. Pani Lidia Staroń ustawicznie podejmuje interwencje w obronie pokrzywdzonych zarówno w sprawach indywidualnych, jak i w sprawach całych grup społecznych. Zawsze po stronie ludzi. Pomaga osobom pokrzywdzonym przez urzędy, instytucje, sędziów, prokuratorów, syndyków i komorników. Odzyskuje pieniądze, ruchomości, domy (Dzwonek) odebrane w wyniku przestępstwa. Zarówno wysoki poziom wiedzy merytorycznej, jak i bogate doświadczenie zawodowe, a także działalność społeczna wskazują, iż pani Lidia Staroń jest dobrym kandydatem na stanowisko rzecznika praw obywatelskich. W imieniu grupy posłów z Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni, grupy posłów Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska - PSL, UED, Konserwatyści, grupy posłów Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewicy (Nowa Lewica, PPS, Razem, Wiosna Roberta Biedronia), grupy posłów Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. grupy posłów Koła Parlamentarnego Polska 2050, grupy posłów Koła Poselskiego Polskie Sprawy oraz grupy posłów niezrzeszonych kandydaturę pana Marcina Wiącka przedstawi pan poseł Krzysztof Paszyk. Bardzo proszę.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu grupy posłanek i posłów, których przynależność polityczna wykracza ponad utarte podziały sali sejmowej, chciałbym zaprezentować i zarekomendować Wysokiej Izbie osobę pana prof. Marcina Wiącka jako kandydata na rzecznika praw obywatelskich. Pan prof. Marcin Wiącek jest prawnikiem. Od 2009 r. jest nauczycielem akademickim na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie jako profesor uniwersytecki od 2017 r. kieruje Zakładem Praw Człowieka. W 2009 r. prof. Wiącek obronił rozprawę doktorską, zaś w 2013 r. został doktorem habilitowanym. Jest uczniem znakomitego nauczyciela, prof. Janusza Trzcińskiego, który pełnił funkcję wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego oraz prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego. Pomimo młodego wieku prof. Wiącek w zasadzie od początku swojej kariery prawniczej sprawnie łączył naukę w zakresie prawa i praktykę prawniczą.

W tym samym okresie był również kierownikiem aplikacji legislacyjnej prowadzonej przez Rządowe Centrum Legislacji. Doświadczenie praktyczne prof. Wiącka jest więc rozległe i bardzo bogate. Jest autorem przeszło 100 publikacji naukowych o tematyce prawniczej, w szczególności w zakresie prawa konstytucyjnego, ochrony praw człowieka oraz sądownictwa konstytucyjnego i sądownictwa administracyjnego. Był uczestnikiem licznych krajowych oraz międzynarodowych konferencji naukowych. Pisał również opinie prawne, rozwiązujące problemy natury prawnej. W 2018 r. na prośbę Fundacji Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego prof. Wiącek przygotował projekt ustawy o zapewnieniu godnej pamięci i należytej ochrony miejscom spoczynku bohaterów powstania warszawskiego oraz innych osób zasłużonych w walkach o niepodległość i suwerenność państwa polskiego. Naukowo prof. Wiącek przez wiele lat zajmował się prawem konstytucyjnym oraz prawem administracyjnym, w tym kwestiami procedury administracyjnej. Obecnie w spektrum jego zainteresowań jest problematyka szeroko pojętych praw człowieka. Podkreślenia wymaga, że zagadnienia naukowe, które rozstrzyga prof. Wiącek, nie mają tylko i wyłącznie wymiaru naukowego.

Należy uznać bez wątpliwości, że przygotowanie naukowe, znakomity warsztat prawniczy oraz doświadczenie naukowe i praktyczne prof. Wiącka zdobywane podczas piastowania wielu wysokich funkcji, zarówno w organach polskiej władzy sądowniczej, jak i w instytucjach służących pomocą prawną, wymagających profesjonalnej, specjalistycznej wiedzy prawniczej, w szczególności w ramach działań Rady Legislacyjnej przy prezesie Rady Ministrów, w pełni predysponują jego kandydaturę do wyboru na nowego rzecznika praw obywatelskich. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proponuję, aby Sejm wysłuchał w dyskusji 2-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół. Przepraszam bardzo. Proszę pana posła Krzysztofa Lipca o przedstawienie opinii komisji. Bardzo dziękuję.

Proszę bardzo.

Naprawdę każdy, kto jest patriotą, powinien chcieć dzisiaj zakończyć ten spór. Zagłosujcie na prof. Wiącka, który ma gwarancję, że Senat go poprze, wyrazi zgodę. Naprawdę warto, żebyśmy pokazali, że jesteśmy Polakami, że zależy nam na tym, żeby Polska miała rzecznika praw obywatelskich, a nie rzecznika politycznego. Poprzyjcie profesora, który jest niezależny i który spełnia wszystkie gwarancje, a nie jest politycznym człowiekiem wyciągniętym z kapelusza. Naprawdę proszę was: pokażcie, że jesteście patriotami.

Proszę teraz pana posła Krzysztofa Lipca o przedstawienie opinii komisji. Bardzo proszę, panie pośle. Bardzo dziękuję. Wysoka Izbo! W imieniu Komisji Sprawiedliwości i Praw człowieka przedstawiam Wysokiemu Sejmowi opinię w sprawie wniosków dotyczących wyboru rzecznika praw obywatelskich. Komisja rozpatrywała dwa wnioski.

Dziękuję. Proponuję, aby Sejm wysłuchał w dyskusji 2-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął.

Proszę państwa. Dobrze, 3 minuty. Odstępujemy od głosowania, tak? Dobrze. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę.

Wysoka Izbo! Od 9 miesięcy trwa wybór rzecznika praw obywatelskich. To już piąte podejście do wyboru tego konstytucyjnego organu. Każde z ugrupowań reprezentowanych na tej sali mogło wskazać swoją kandydatkę lub swojego kandydata marzeń. Ani nasi kandydaci, ani posłowie PiS nie uzyskali wsparcia w Senacie. Jeśli jest się posłem lub senatorem, to każde głosowanie, każdy wybór to czysta polityka. To, że ktoś bardzo chce, nie może być wystarczającym atutem. Potrzebne są wyróżniająca wiedza prawnicza, niezależność, logika i precyzja w prezentowaniu wizji sprawowania urzędu, prawdomówność, ale także brak wątpliwości. Ostatnie zawiadomienia do prokuratury nie budzą respektu wobec jednej z kandydatur. PiS konsekwentnie poszukuje kandydatów na kluczowe urzędy, na których można mieć prokuratorskie trzymanie. Nie przesądzając zasadności zarzutów, badanie w trakcie kadencji rzecznika sprawy w prokuraturze mogłoby mieć wpływ na jego funkcjonowanie, być swoistym efektem mrożącym. Dostajemy dzisiaj również propozycję kompromisowego kandydata, zaproponowanego przez środowisko akademickie, a dokładnie przez Radę Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Prof. Marcin Wiącek to na pewno kandydat świetnie przygotowany, naukowiec. Wyróżnia się on wiedzą prawniczą, a w szczególności znajomością obszaru praw człowieka. Ponieważ konsekwentnie unika demonstracji swoich poglądów politycznych, swojego światopoglądu, może stworzyć model sprawowania urzędu otwartego dla wszystkich, do którego bez żadnego trybu każdy i każda mogą się zgłosić ze swoim problemem.

Nie bał się on merytorycznej rozmowy, debaty i nie uciekał od niej. Odpowiadał na zaproszenia. Nikt na tej sali nie ma żadnego powodu, by odmówić poparcia prof. Wiąckowi, ani merytorycznego, ani politycznego. Koalicja Obywatelska jest na tak. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Przez tyle czasu nie jesteśmy w stanie jako parlament wybrać rzecznika praw obywatelskich. Tyle czasu trwa klincz, którego ofiarą padają obywatele. którzy mają konstytucyjnie zagwarantowane prawo do złożenia skargi, do poszukiwania ochrony u niezależnego organu konstytucyjnego, jakim jest rzecznik praw obywatelskich. Tyle trwa klincz, którego autorem jest Prawo i Sprawiedliwość, które ciągle podejmuje próby upchania na tym stanowisku partyjnego albo upolitycznionego kandydata. Dzisiaj podejmujemy piątą próbę. Dzisiaj mamy szansę wybrać kandydata kompromisu, kandydata ponadpartyjnej zgody. To prof. Marcin Wiącek. Każdy musiał się posunąć. Każdy uznał, że dobro Polaków jest ważniejsze niż partyjny interes czy partyjny nominat. Dziś jest sprawdzian z odpowiedzialności i troski o państwo, o prawa obywateli. Możemy wybrać prawnika, profesjonalistę albo kandydatkę, której jedną z niewielu zalet jest to, że po prostu bardzo chce. Klub Lewicy będzie głosował za kandydaturą prof. Marcina Wiącka. Kontynuuje pani poseł Katarzyna Ueberhan, Lewica. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Czternastolatkę gwałci 26-letni kuzyn, a sąd II instancji obniża wyrok, bo ofiara nie krzyczała. 18-letni obywatel Ukrainy zbiera pieniądze na cel społeczny i zostaje pobity przez funkcjonariuszy Policji. Czternastolatek udostępnia post o Strajku Kobiet, w domu nachodzi go policja. Kolorowe flagi obrażają pomniki, gminne uchwały odczłowieczają, a 48 osób zostaje aresztowanych i wywiezionych na różne posterunki Policji za okazaną solidarność. Tysiące dzieci znika z systemu edukacji w czasie pandemii, bo nie wiadomo, kto i jak ma to kontrolować. To tylko kilka z 72 tys. ludzkich spraw z ostatniego roku, w których interweniował rzecznik praw obywatelskich i jego biuro. 72 tys. powodów, dla których potrzebujemy rzecznika praw obywatelskich dziś. Nadmierne upartyjnienie struktur państwowych, mało wydajny system opieki zdrowotnej, niewłaściwie reformowany system sprawiedliwości, kryzys praworządności, kryzys pandemiczny, a pośrodku tego człowiek. Osoby najsłabsze, których prawa i wolności wymagają dzisiaj szczególnej ochrony. Tylko wtedy, gdy człowiek i jego godność staną w centrum widzenia naszego świata, gdy w drugim, w tym innym, zobaczymy też człowieka, tylko wtedy i tylko tam, w człowieku i w obronie jego godności, odnajdziemy nasze wspólne wartości - nasz naród, nasze państwo i rzecznika naszych praw.

Pani Marszałek! Dzisiaj w tej Izbie, w tym momencie, trzeba zadać sobie pytanie, czy rzecznikiem praw obywatelskich powinna zostać osoba, o której szef klubu rekomendującego mówi: dlatego ją zgłaszamy, bo chce. Czy rzecznikiem praw obywatelskich ma zostać osoba, która kiedyś była w zarządzie krajowym jednej z liczących się partii politycznych w tym kraju. a dzisiaj, choć wybrana niezależnie, z własnego komitetu, opuszcza salę senacką w ramach obstrukcji działań Senatu Rzeczypospolitej? Czy osobą dzisiaj rekomendowaną przez Sejm na rzecznika praw obywatelskich powinna być osoba, co do której media ujawniają wiele wątpliwości dotyczących działalności, którą prowadziła przez ostatnie lata? Czy jednak powinniśmy wznieść się ponad tą polityczną zajadłość, ponad te polityczne spory i postawić na kandydata, który chce być rzecznikiem Polek i Polaków? Nie chce być rzecznikiem poglądów politycznych, idei politycznych, rzecznikiem jakiejkolwiek partii politycznej. Naszym zdaniem, zdaniem klubu Koalicji Polskiej - Polskiego Stronnictwa Ludowego, który mam przyjemność reprezentować, taką właśnie osobą jest pan prof. Marcin Wiącek. To osoba, która nigdy nie należała ani nie należy do żadnej partii politycznej, która w ostatnich latach absolutnie nie wikłała się, nie angażowała się po którejkolwiek stronie politycznych sporów, które wybuchały. To osoba, która naukowo, ale i praktycznie zajmuje się ochroną praw człowieka, rzeczą niezwykle dzisiaj ważną z punktu widzenia interesów Polek i Polaków.

Naprawdę chcielibyśmy bardzo prosić Wysoką Izbę, by raz wznieść się ponad te podziały, które są tu naprawdę w wielu momentach niezwykle destrukcyjne, i poprzeć osobę pana prof. Marcina Wiącka, o co chciałbym bardzo serdecznie prosić. Pan poseł Dobromir Sośnierz, Konfederacja.

Konfederacja nie interesuje się tym, kto kogo zgłosił, nie interesują nas te układy, układziki, przepychanki. Każdego kandydata zawsze ocenialiśmy i oceniamy indywidualnie. W tym przypadku również byliśmy otwarci, zaprosiliśmy oboje kandydatów na dyskusję. Niestety oboje tę dyskusję przegrali: pani Lidia Staroń walkowerem, ponieważ nie przyszła, a pan Wiącek oprócz tego, że mówił parę rzeczy rozsądnych, to niestety mówił też parę takich, których nie dało się słuchać, jak o walce z luką płacową, wydumaną przez feministki. W związku z tym posłowie Konfederacji ocenią indywidualnie każdego kandydata i zobaczymy, gdzie nas to doprowadzi. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan poseł Tomasz Zimoch, Polska 2050. Wysoki Sejmie! Koło Parlamentarne Polska 2050 udziela poparcia prof. Marcinowi Wiąckowi. To prawnik, naukowiec, specjalista z zakresu prawa konstytucyjnego i praw człowieka. Senator Lidia Staroń nie przekonała, że wyróżnia się wiedzą prawniczą, czego wymaga ustawa o RPO. W czasie posiedzenia komisji sprawiedliwości nie odpowiedziała właściwie na żadne pytanie posłów. Prof. Wiącek wie, jak skutecznie dochodzić praw obywatelskich. Daje rękojmię, że w swoich działaniach będzie niezależny, niezawisły i apolityczny. Przekonywająco brzmi jego zapowiedź, że będzie - niech pan posłucha, panie pośle Suski - niezależnym adwokatem całego społeczeństwa. Jego wystąpienie i odpowiedzi w czasie posiedzenia komisji były wykładem prawa. Szkoda, że pan, panie Suski, tam nie był i tej lekcji prawa dla każdego nie odbył. Podkreśla na każdym kroku, jak ważna jest ochrona godności człowieka, która zgodnie z art. 30 konstytucji stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Dlatego jesteśmy przekonani, że każda osoba szukająca wsparcia, niezależnie od poglądów politycznych i tożsamości religijnej, kulturowej, narodowej czy seksualnej, będzie mogła widzieć w tym kandydacie rzecznika swoich praw. W szczególności Koło Parlamentarne Polska 2050 docenia krytyczną ocenę funkcjonowania Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie, konieczną kontynuację w zakresie realizacji zadań z zakresu Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur, wyrażaną troską o prawa osób zatrzymanych i tymczasowo aresztowanych oraz osób w kryzysie bezdomności, jak również konieczność przestrzegania łamanej ostatnio przez rządzących wolności zgromadzeń. Cieszą deklaracje kandydata dotyczące konieczności pełniejszej realizacji przez Polskę międzynarodowych zobowiązań w zakresie ochrony środowiska, czyli np. wynikającej z podpisanej 23 lata temu, a ratyfikowanej przez Polskę w 2003 r. konwencji z Aarhus możliwości zaskarżenia planów urządzenia lasu czy planów łowieckich, które to prawa nie są realizowane w naszym ustawodawstwie, a także prawa do czystego powietrza. Pani Marszałek! Panie Posłanki i Panowie Posłowie! Zwracam się z kolejnym apelem, który tu już był słyszany z ust innych posłów: bądźmy dzisiaj naprawdę ponad podziałami. Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Rzecznik praw obywatelskich powinien być niezależnym adwokatem społeczeństwa. Tak mogłaby brzmieć skrócona definicja tej funkcji. Absolutnie zgadzam się z tym stwierdzeniem, a są to słowa pana prof. Wiącka. Wspólnie z pozostałymi posłami koła Polskie Sprawy podpisaliśmy się pod jego kandydaturą. Nie jest politykiem ani nie jest związany z żadną partią polityczną. Bardzo dobrze. Pracował w Radzie Legislacyjnej przy premierze za rządów PO-PSL, a także za rządów PiS. To również cieszy, bo pokazuje, że jego kompetencje były cenione i wykorzystywane bez względu na zmieniającą się władzę. Kieruje Zakładem Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Nie wiem jak dla państwa, ale dla mnie to również jest całkiem istotna zaleta. Uczestniczył w debacie, którą zorganizowała Konfederacja. To pokazuje, że nie obawia się konfrontacji. Niestety podczas debaty zabrakło kontrkandydatki. Szkoda, ale to również wiele mówi. Rzecznik praw obywatelskich musi być niezależny. Pożądane jest, żeby nie był powiązany z partią rządzącą, ponieważ w czasie jego pracy najprawdopodobniej będą występowały sytuacje, w których będzie stawał po stronie obywatela w kontrze do decydentów politycznych. Musi stać po stronie obywatela. Wysoka Izbo! Koleżanki i Koledzy Posłowie! Stańmy dziś na wysokości zadania. Parlament od kilku miesięcy nie może wybrać rzecznika praw obywatelskich. To wstyd. To kolejny argument za tym, aby obywatele sami wybierali swojego rzecznika. Na chwilę obecną nie jest to możliwe, dlatego liczę na to, że tym razem wszyscy schowamy interes partyjny do kieszeni i podejdziemy do tego głosowania odpowiedzialnie. Koło Poselskie Polskie Sprawy będzie głosować za kandydaturą pana prof. Wiącka. Lista posłów zapisanych do głosu została wyczerpana. Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka zaopiniowała pozytywnie kandydaturę pani Lidii Staroń na stanowisko rzecznika praw obywatelskich oraz negatywnie kandydaturę pana Marcina Wiącka na stanowisko rzecznika praw obywatelskich.

Wobec tego Sejm przeprowadzi w tej sprawie głosowanie za pomocą urządzenia do liczenia głosów, wykorzystując funkcję tego urządzenia umożliwiającą dokonanie wyboru z listy. Przedstawiam zasady głosowania z wykorzystaniem funkcji umożliwiającej dokonanie wyboru z listy. Po zarządzeniu głosowania na wyświetlaczu pojawią się nazwiska i imiona kandydatów. Aby oddać głos na kandydata, należy zaznaczyć jego nazwisko i imię. Potwierdzenie zaznaczenia pojawi się w polu wyboru. Aby zmienić decyzję, należy usunąć zaznaczenie kandydata, a znak potwierdzenia obok nazwiska i imienia zniknie. Po dokonaniu wyboru należy zatwierdzić swoją decyzję przez naciśnięcie przycisku „Zatwierdź i wyślij” Jest to równoznaczne z ostatecznym oddaniem głosu, a zatem brakiem możliwości zmiany decyzji. Niezaznaczenie żadnego kandydata i naciśnięcie przycisku „Zatwierdź i wyślij” jest równoznaczne z oddaniem głosu przeciwko wszystkim kandydaturom. Przechodzimy do głosowania.

Przypominam, że na stanowisko rzecznika praw obywatelskich zgłoszone zostały kandydatury pani Lidii Staroń oraz pana Marcina Wiącka. Po rozpoczęciu głosowania lista w kolejności alfabetycznej zostanie umieszczona w urządzeniu do liczenia głosów. Przypominam, że poprzeć można tylko jedną kandydaturę. Ponownie przypominam, że naciśniecie przycisku „Zatwierdź i wyślij” jest równoznaczne z ostatecznym podjęciem decyzji, a zatem bardzo proszę, aby tego przycisku użyć jako ostatniego. Przystępujemy do głosowania. Proszę obecnie panie i panów posłów o podejmowanie decyzji w sprawie powołania rzecznika praw obywatelskich.

Panie pośle, to państwo posłowie zgłaszają, że jest problem, i dlatego czekam, żeby uzyskać połączenie.

Zamykam głosowanie i proszę o wyniki.

Sejm bezwzględną większością głosów powołał panią Lidię Staroń na stanowisko rzecznika praw obywatelskich. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 7. porządku dziennego: Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr 1265) Prezydium Sejmu na podstawie art. 20 ust. 1 regulaminu Sejmu, po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów, przedłożyło wniosek w sprawie zmian w składach osobowych komisji sejmowych. Czy ktoś z pań i panów posłów pragnie zabrać głos w sprawie przedstawionych propozycji? Nikt się nie zgłasza. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku w brzmieniu z druku nr 1265, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

państwo już za długo siedzicie. Proszę bardzo. Dziękuję. Jakich wyników?

za, 1 - przeciw, wstrzymało się 19. Sejm podjął uchwałę w sprawie zmian w składach osobowych komisji sejmowych.

Jak to, nie było wyświetlonych wyników na tablicy?

Wznawiam obrady. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 8. porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1222) Proszę sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości pana Sebastiana Kaletę o przedstawienie uzasadnienia projektu ustawy. Proszę bardzo. Wysoka Izbo!

TSUE dostrzegł, że obecnie funkcjonujące w polskim systemie rozwiązania regulujące postępowania sądowe w sytuacjach, w których przedsiębiorca pozywa konsumenta o zapłatę, przedkładając sądowi wraz z pozwem wyłącznie wystawiony przez konsumenta weksel, mogą zniechęcać konsumenta do podjęcia obrony. Taka sytuacja wymaga zmian, które rozszerzą ochronę konsumentów, jednocześnie zniechęcając przedsiębiorców do sporządzania w obrocie konsumenckim umów, w których będą zawarte nieuczciwe postanowienia krzywdzące konsumentów. TSUE zakwestionował również regulację funkcjonującą w polskim postępowaniu cywilnym, która utrzymuje monopol operatora wyznaczonego na świadczenie usług pocztowych związanych z nadawaniem przez strony czy uczestników postępowania pism procesowych do sądu, kiedy to nadanie wiąże się z zachowaniem terminu do dokonania określonej czynności procesowej. Chciałbym podkreślić, że istotą tego projektu są zmiany, które będą służyć obywatelom, w szczególności konsumentom w postępowaniach sądowych. Po pierwsze, projekt ma spowodować, że sąd z urzędu będzie badał umowę, w której roszczenia przedsiębiorcy zabezpieczą wystawiony przez konsumenta weksel pod kątem istnienia w takiej umowie klauzul niedozwolonych. Kontrola sądu ma dotyczyć nie tylko samej umowy, ale również deklaracji wekslowej oraz załączników do umowy.

Korzyść dla konsumentów m.in. polega na tym, że termin do wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty będzie wydłużony do 1 miesiąca, a opłata od zarzutów nie będzie mogła wynosić więcej niż 750 zł. Konsekwencją wprowadzonych zmian do prawa procesowego jest rozszerzenie w dalszych przepisach projektu ochrony konsumenta na gruncie prawa materialnego, tj. prawa wekslowego, ustawy o kredycie konsumenckim oraz Kodeksu wykroczeń, których charakter jest w zasadzie służebny, jako skutek zmiany podstawowej regulacji, tj. prawa wekslowego. Zmiany w ustawie - Prawo wekslowe dotyczą w szczególności wyłączenia przenoszalności weksla, który wystawił konsument. Zmiana ta ma zapewnić, aby powód, który wystąpi na drogę sądową przeciwko konsumentowi, miał realną możliwość dysponowania umową, której postanowienia zostały zabezpieczone wekslem wystawionym przez konsumenta. Brak takiej zmiany mógłby prowadzić do sytuacji, w której kolejny nabywca weksla nie mógłby wykonać zobowiązania sądu do przedłożenia umowy, uniemożliwiając tym samym sądowi kontrolę nieuczciwych warunków. Kolejna istotna zmiana w tym projekcie dotyczy Kodeksu postępowania cywilnego. Projekt dostosowuje do wymogów prawa Unii Europejskiej przepis art. 165 § 2 k.p.c. w taki sposób, żeby oddanie pisma procesowego w formie przesyłki pocztowej w polskiej placówce każdego operatora pocztowego lub w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej było równoznaczne z wniesieniem go do sądu. Zagwarantuje to dostarczanie do sądu nadanych przesyłek w odpowiednim i przewidywalnym czasie oraz zachowanie terminu do dokonania czynności procesowej. Ostatnia kategoria proponowanych zmian dotyczy implementacji wyroku w sprawie C-670/15, który spowodował, że zachodzi konieczność nowelizacji ustawy o prawie pomocy w postępowaniach w sprawach cywilnych prowadzonych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz o prawie pomocy w celu ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem takiego postępowania. W tym zakresie projekt przewiduje zmianę, zgodnie z którą osoba ubiegająca się o pomoc prawną będzie mogła uzyskać zwrot poniesionych kosztów tłumaczeń dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku o przyznanie prawa pomocy. Bez tej zmiany brzmienie obowiązującego przepisu budziło wątpliwości i niepożądaną niepewność sytuacji osoby ubiegającej się o pomoc prawną, co oczywiście należy doprecyzować i co też przedłożony projekt czyni. Panie Marszałku! Pozostaję w przekonaniu, że dzięki zaproponowanym rozwiązaniom zostanie zapewniony wysoki poziom ochrony słabszych stron postępowania sądowego, w szczególności konsumentów. Proszę Wysoką Izbę o poparcie przedstawionego projektu. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu ministrowi. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół. Proszę o zabranie głosu pana posła Marka Asta, który przedstawi stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Panie Ministrze! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam zaszczyt przedstawić stanowisko wobec rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, druk nr 1222.

Nadto w konsekwencji projekt wyłączył też przenoszalność ze skutkiem indosu praw z weksla wystawionego przez konsumenta na osobę trzecią. Taka praktyka będzie niedozwolona. Zmianą w dobrym kierunku jest też zniesienie monopolu operatora pocztowego, jeżeli chodzi o kwestię doręczeń. Jednym słowem są to zmiany, które wzmacniają pozycję konsumenta względem przedsiębiorców, którzy do tej pory mieli procedury związane z egzekwowaniem należności z umowy w oparciu o weksel zdecydowanie bardziej korzystne, w szczególności jeżeli zawierali w umowach klauzule niedozwolone, a nie podlegało to kontroli. Należy więc stwierdzić, że z jednej strony jest to oczywiście implementacja, czyli obowiązek państwa polskiego, ale jednocześnie są to zmiany, które idą w dobrym kierunku. W tej sytuacji oczywiście w imieniu klubu wnoszę o skierowanie projektu ustawy do dalszych prac legislacyjnych we właściwej komisji. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Proszę teraz panią poseł Barbarę Dolniak o to, aby przedstawiła stanowisko Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Pojawia się tutaj kilka zmian, które dla stron postępowania sądowego będą miały znaczenie, m.in. możliwość nadania przesyłki do sądu nie tylko u jednego operatora pocztowego, ale w każdym przedsiębiorstwie, które jest wpisane do rejestru operatorów pocztowych zarówno w Polsce, jak i na terenie Unii Europejskiej. Ale to akurat dobre rozwiązanie, ponieważ strona będzie mogła zawsze wykazać, że złożyła pismo procesowe do sądu. Istotna jest również kwestia zmian dotyczących konsumenta. Składający pozew do sądu będzie musiał wskazać w pozwie, czy przeciwnik, czyli pozwany, jest konsumentem. Jeżeli tego nie zrobi, sąd będzie mógł wezwać stronę do uzupełnienia braku pod rygorem zwrotu pozwu.

Nadto przyznane jest uprawnienie do wydania z urzędu postanowienia zmieniającego treść nakazu, jeżeli chodzi o czas na zaskarżenie tego nakazu. Ważna jest również kwestia dotycząca weksla, a mianowicie projekt przewiduje zakaz przenoszenia praw z weksla wystawionego przez konsumenta na inne osoby, np. firmę windykacyjną, i obejmuje nie tylko, jak teraz, kredyt konsumencki, ale także wszelkie umowy konsumenta z przedsiębiorcą. Ochrona ta ma przy tym obejmować nie tylko dłużnika, ale także poręczycieli. Występujący z wekslem będzie musiał przedstawić sądowi umowę. Jeżeli tego nie zrobi i sąd stwierdzi jakiekolwiek wątpliwości, będzie mógł on przekazać sprawę do rozpoznania w postępowaniu zwykłym. Przypomnę, że nakazy zapłaty z weksla wydawane są w trybie nakazowym - to po pierwsze. Ponadto oprócz tych rozwiązań przewidziana jest również możliwość uzyskania zwrotu kosztów tłumaczenia. W ustawie o kosztach sądowych jest określenie rozwiązania dotyczącego górnej granicy opłaty od zarzutów dotyczących nakazu zapłaty. Będzie również możliwość uzyskania zwrotu kosztów dotyczących tłumaczenia.

Ustawa ta w zakresie swojej treści, jak i z uwagi na potrzebę zmian zgodnie z orzeczeniami, z wyrokami Trybunału Sprawiedliwości - co do niektórych kwestii sądy już stosują bezpośrednio orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej - wejdzie w życie. Uchwalimy projekt ustawy, który pozwoli stronom na szybsze i sprawniejsze dochodzenie swoich racji, a jednocześnie da on możliwość przedstawienia argumentów w postaci np. umowy, jeżeli mówimy o wekslu. To rozwiązanie daje szansę na ocenę (Dzwonek) przez sąd zasadności roszczenia przed wydaniem nakazu zapłaty w trybie nakazowym. Bardzo dziękuję. Proszę teraz panią poseł Katarzynę Ueberhan, która przedstawi stanowisko klubu parlamentarnego Lewica. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam przyjemność przedstawić stanowisko klubu Lewicy w sprawie rządowego projektu ustawy z druku nr 1222 o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, projekt, który ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej. Obowiązkowa kontrola umowy, a nie tylko weksla, dłuższy termin na odwołanie i niższe opłaty sądowe, mające wzmocnić obywateli w sporach z przedsiębiorcami i zwiększyć ochronę konsumentów przed działaniami dużych firm, w tym banków - takie zmiany przewiduje niniejsze przedłożenie, rządowy projekt noweli Kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Podstawowy cel zmiany ustawy wynika z wdrożenia wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie tzw. postępowania nakazowego z weksla w sporach przeciw konsumentom. Zgodnie ze wskazaniem Trybunału Sprawiedliwości krajowym sądom cywilnym, w tym orzekającym w nich referendarzom zmienione przepisy stwarzają możliwości kontroli umowy i jej załączników, którą przedstawiony sądowy weksel zabezpieczał, i to jeszcze przed wydaniem nakazu zapłaty. Wszystko po to, aby wychwycić niedozwolone abuzywne postanowienia umowne. Należy przy tym pamiętać, że wydany na posiedzeniu niejawnym bez udziału pozwanego, a nawet jego pisemnego stanowiska, nieprawomocny nakaz zapłaty z chwilą wydania stanowi tytuł zabezpieczenia wykonalny bez nadania mu klauzuli, który jest dla osoby pozwanej prawie tak samo dolegliwy jak zajęcie komornicze. Projekt poszerza też zakaz przenoszenia praw z weksla, tzw. indosu, wystawionego przez konsumenta na inne osoby, np. firmy windykacyjne, i obejmuje nie tylko, jak do tej pory, kredyty konsumenckie, ale wszelkie umowy konsumenta z przedsiębiorcą. Ochroną taką ma obejmować nie tylko samego dłużnika, to jest strony umowy zawartej z przedsiębiorcą, ale też i poręczycieli. Bez tego sąd nie wyda wyroku i skieruje sprawę do zwykłego procesu, więc pozwany konsument uzyska możliwość prezentacji swych racji przed wydaniem orzeczenia. Co równie ważne, przedłużony zostaje też termin na odwołanie od nakazu zapłaty na tzw. zarzuty - do miesiąca, jeśli dłużnik przebywa na terenie Polski, i 3 miesięcy, gdy doręczenie ma nastąpić poza Unią Europejską. Dla uniknięcia komplikacji terminy te mają dotyczyć zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. Nowe rozwiązania umożliwiają również oddanie pisma procesowego, z zachowaniem powyższego terminu, w placówce dowolnego operatora pocztowego świadczącego usługi powszechne - w formie przesyłki poleconej. To znacznie mniej niż obecnie w zwykłym postępowaniu. Ponieważ projekt dostosowuje polskie przepisy do orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zapadłych na kanwach spraw wniesionych z Polski oraz Niemiec i dzięki nowym rozwiązaniom zwiększy ochronę prawną obywateli, a konsumenci i inne strony postępowania cywilnego będą mogli korzystać z porównywalnego w całej Unii Europejskiej poziomu ochrony swoich praw, klub Lewicy popiera niniejsze przedłożenie w obecnie przedłożonym kształcie. Bardzo dziękuję. Proszę teraz pana posła Krzysztofa Paszyka, który przedstawi stanowisko Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska. Bardzo dziękuję. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska - PSL, Unia Europejskich Demokratów, Konserwatyści chciałbym przedstawić nasze stanowisko do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, zawartego w druku nr 1222. Jeśli chodzi o omówienie przedmiotowego projektu, to właściwie wszystkie jego główne założenia zostały przybliżone przez przedmówców. Chciałbym w swoim wystąpieniu zwrócić projektodawcom uwagę, która jest również wyrażana przez Naczelną Radę Adwokacką, a dotyczy tego, że przy okazji projektowanych zmian nie pomyślano o odmiejscowieniu, jeśli chodzi o nadawanie korespondencji, tylko pozostał wymóg nadania pisma w placówce operatora pocztowego, a jak wiemy, nasza rzeczywistość jest dzisiaj taka, że świat idzie do przodu. Mamy różnego rodzaju listomaty, formy coraz bardziej mobilne i ułatwiające nadawanie przesyłek.

Może uda się w toku prac pomyśleć o tym, aby to spostrzeżenie, które nie jest spostrzeżeniem o charakterze politycznym, tylko pochodzi od fachowców, od profesjonalistów, w projekcie ująć.

Bardzo dziękuję panu posłowi.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W prawie najważniejszą rzeczą jest to, żeby nie było często zmieniane.

Otóż ja nie jestem zwolennikiem niewolniczego naśladowania tego, co jest w Unii - wręcz przeciwnie. Jeżeli mają być jakieś zmiany, to powinny być dobre, nie złe, a nie - unijne albo nieunijne. Takie jest stanowisko Konfederacji. Chciałem tutaj rozczarować Lewicę, bo zmiany. Ustawodawcom się wydaje, że coś zmieniają, natomiast ludzie się do tego świetnie dopasowują. Mogę się założyć, że jeżeli chcemy tutaj po lewacku promować biednego, drobnego konsumenta przeciwko wielkim firmom, to wielkie firmy po prostu wynajmą sobie zwykłego szarego obywatela, który będzie za nich prowadził sprawy i trzeba będzie pozywać zwykłych szarych obywateli, a nie wielką firmę.

W tym celu musi być swobodna trasata weksla, tak samo jak jest swobodne przenoszenie stuzłotówki z obywatela na obywatela.

Oddając już głos mojemu szanownemu koledze, chciałbym poprosić również, żeby rząd zastanowił się nad zmniejszeniem opłat patentowych, bo liczba patentów w Polsce drastycznie spada, bo ludzi nie stać na nieprawdopodobnie wysokie opłaty za patent. Dziękuję za uwagę. Bardzo proszę.

Nie popieram przede wszystkim ingerencji prawa wykroczeniowego w stosunki umowne, a tym bardziej jej dalszego rozszerzania. Rozumiem, że od biedy można uznać, że jakieś postanowienia umowne są po prostu nieważne, jeśli bardzo się upieramy, żeby tę wolność umów ograniczyć, ale traktowanie jakiejś dobrowolnie zawartej umowy jako wykroczenia to jest zła droga. Nie idźcie w tym kierunku. Mam też mieszane uczucia wobec zmiany dotyczącej doręczeń. Zgoda na oddawanie przesyłek sądowych z innych krajów może sprzyjać niestety - jako efekt uboczny - dalszemu wydłużaniu tych postępowań.

Myślę, że problem zagranicznych przesyłek lepiej rozwiązać za pomocą doręczeń elektronicznych, nad czym też już pracujemy.

Dziękuję bardzo. Teraz pan poseł Tomasz Zimoch przedstawi stanowisko koła poselskiego Polska 2050.

Panie Ministrze! Zatem w trybie mini-maks: minimum słów, maksimum dobrego prawa. Koło Parlamentarne Polska 2050 popiera ten projekt, bo legislatorzy mówią w takich sytuacjach: nie ma wyjścia, trzeba wdrożyć wyroki Trybunału Sprawiedliwości do polskiego prawa. I panie ministrze, oby to nigdy nie budziło żadnych wątpliwości, jeśli chodzi o rozstrzygnięcia Trybunału. Projekt ustawy zmieniającej Kodeks postępowania cywilnego i inne ustawy powstał właśnie w wyniku kilku rozstrzygnięć Trybunału. Słusznie podkreśla się w uzasadnieniu, że konsekwencją zmian wprowadzonych do prawa procesowego jest rozszerzenie w dalszych przepisach projektu ochrony konsumenta na gruncie prawa materialnego.

Mam pytania dotyczące paru kwestii. Teraz będzie można kierować przesyłki z pismami do sądu za pośrednictwem operatora pocztowego wpisanego do rejestru. W związku z tym mam pytanie: Czy ministerstwo planuje na swojej stronie wskazywać, jakie są to podmioty, którzy operatorzy pocztowi prowadzący działalność wpisani do rejestru przyjmują przesyłki i do których można je składać?

Jest też możliwość uzyskania... [[Dzwonek]] 750 zł to górny pułap opłaty od zarzutów w nakazie zapłaty.

Dziękuję bardzo. Pytanie zada teraz pan poseł Michał Gramatyka. Panowie Ministrowie! Wysoka Izbo! W przedłożeniu zmieniają państwo m.in. art. 165 Kodeksu postępowania cywilnego. Tam używacie takiego sformułowania: oddanie pisma procesowego w formie przesyłki poleconej w placówce pocztowej w Polsce lub w Unii Europejskiej. W obecnym stanie prawnym funkcjonuje również art. 165 § 4 zawierający normę: wprowadzenie pisma do systemu teleinformatycznego sądu. Moje pytanie: Jak nowelizacja k.p.c., nad którą pracujemy, ma się do art. 63 ustawy o doręczeniach elektronicznych, która przygotowuje nas na cyfrową komunikację m.in. z sądami? Tam ten obowiązek przyjmowania pism cyfrowych jest wprawdzie wyrażony, ale jest osłabiony takim enigmatycznym sformułowaniem: jeżeli warunki techniczne i organizacyjne sądu to umożliwiają.

Bardzo dziękuję. Dziękuję. Pytanie zada pan poseł Jan Szopiński. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Czy Polska faktycznie musi być upokarzana przez TSUE wyrokami przywołanymi w tym druku sejmowym?

Czy tak trudno było dopilnować współbrzmienia Kodeksu karnego z Kodeksem postepowania cywilnego w kwestiach tak banalnych jak wskazanie operatora pocztowego lub zauważenie, że niemożliwa jest prawna egzekucja weksla sporządzonego do bezprawnej umowy określającej jego stosowanie? Szanowny Panie Ministrze! Dlaczego pańscy urzędnicy nie zajmują się sprawami, do których zostali powołani? Pytanie zada pani poseł Krystyna Skowrońska. Panie i Panowie Posłowie!

Państwo wskazujecie, że wprowadzamy zakaz przenoszenia indosu z weksla w zakresie przepisów prawa wekslowego i czekowego. W tym zakresie interesuje mnie również. Skoro do umowy czy do weksla dołączona jest deklaracja wekslowa, to jak w tym przypadku podchodzić do możliwości robienia czy rolowania, czy sekurytyzacji kredytów, w tym kredytów konsumenckich, i sprzedawania pakietów innym podmiotom? Jeżeli one nie wpływają (Dzwonek), jeżeli to zabezpieczenie nie działa, to wtedy otrzymujemy, sprzedajemy poniżej tej wartości. W tym zakresie, jeżeli zamykamy stosowanie m.in. przenoszenia indosu w sytuacjach z konsumentami, chciałabym zapytać, jak miałoby się to odbywać w życiu gospodarczym. Czy transakcje gospodarcze pomiędzy podmiotami, które prowadzą działalność gospodarczą, będą możliwe? Dziękuję bardzo. Jako ostatni pytanie zada pan poseł Przemysław Koperski, Lewica. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Zmiany są jak najbardziej potrzebne i w imieniu klubu parlamentarnego Lewicy koleżanka już powiedziała, że będziemy głosowali za. Ale mam pytanie, panie ministrze, zwracam się do pana jako członka polskiego rządu: Czy panu nie wstyd? Po wprowadzeniu tych zmian będzie można oddać pismo procesowe w formie przesyłki poleconej w dowolnym miejscu na terenie Unii Europejskiej, gdzie działa placówka pocztowa. Kiedyś standardem było to, że w miastach wojewódzkich, byłych miastach wojewódzkich placówki pocztowe Poczty Polskiej były czynne 24 godziny na dobę. Teraz mieszkańcy np. Bielska-Białej, żeby nadać przesyłkę w dniu wolnym od pracy, muszą dojeżdżać do Katowic. Czy teraz, panie ministrze, nie będzie panu wstyd, że polscy obywatele będą jeździć np. do Republiki Czeskiej i tam nadawać przesyłki, ponieważ tam te placówki pocztowe dłużej działają (Dzwonek) niż w Polsce? Bardzo dziękuję. Na tym lista osób zapisanych do pytań została wyczerpana. Odpowiedzi na zadane pytania udzieli pan minister Sebastian Kaleta. Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Odpowiadając na pytania, które się pojawiły podczas tej debaty, w pierwszej kolejności chciałbym odnieść się do kwestii kompetencyjnej, dlaczego jest ta ustawa.

W zakresie ochrony konsumentów te kompetencje Unia po prostu na mocy art. 169 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej wprost posiada. Zacytuję: „Dążąc do popierania interesów konsumentów i zapewnienia wysokiego poziomu ochrony konsumentów, Unia przyczynia się do ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i interesów gospodarczych konsumentów, jak również wspierania ich prawa do informacji, edukacji i organizowania się w celu zachowania ich interesów” To jest przepis kompetencyjny. Natomiast w tym obszarze, w którym rzeczywiście prowadzone są spory, jeśli ktoś z panów bądź pań posłów będzie w stanie wskazać przepis kompetencyjny, który mówi, że Unia może wpływać na organizację wymiaru sprawiedliwości w państwie członkowskim i decydować o kształcie i organizacji tego wymiaru sprawiedliwości, to wtedy rzeczywiście być może jest jakieś pole do dyskusji. Takiego przepisu w traktatach w zakresie sądów nie ma, stąd ten spór. Pani poseł pytała o kwestię opłaty, jak została ona ustalona. Dzisiaj opłata od zarzutów od nakazu zapłaty nie różnicuje konsumenta od innych podmiotów i właśnie celem tej ustawy jest wprowadzenie limitu dla konsumenta.

Takie jest źródło ustalenia kwoty w tym przedłożeniu. Jeśli chodzi o kwestię dotyczącą placówek pocztowych i generalnie doręczeń, przyjmowania pism, to lista podmiotów, które mogą świadczyć te usługi, znajduje się w BIP-ie Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Natomiast jeśli chodzi o drugą kwestię, przepis pozwala, z pewnością może wpłynąć na to, że usługi dotyczące jeszcze łatwiejszego nadawania pism mogą stać się bardziej konkurencyjne, ponieważ mogą być firmy, które będą zainteresowane tym, by w sposób bardziej dogodny dla osób, stron postępowań takie usługi świadczyć. A więc w tym zakresie jest tylko udogodnienie, prezentowanie kolejnego udogodnienia. Pozostałe kwestie z pewnością będzie można wyjaśnić na posiedzeniu komisji, niemniej w kilku tych kwestiach warto zaznaczyć od razu, jak się sprawy mają. Dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję. Marszałek Sejmu, po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu, proponuje, aby Sejm skierował projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, zawarty w druku nr 1222, do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w celu rozpatrzenia. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycję przyjął.

Na tym wyczerpaliśmy porządek dzienny 31. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Informuję, że zgłosili się posłowie w celu wygłoszenia oświadczeń poselskich. Czy ktoś z pań i panów posłów pragnie jeszcze wygłosić oświadczenie, dopisać się do listy? Listę posłów zgłoszonych do oświadczeń uważam zatem zamkniętą. Głos ma pan poseł Rafał Adamczyk, Lewica. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowana została zapowiedź projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz niektórych ustaw. Przepisy projektowanej ustawy mają na celu, jak wynika ze wstępu do opracowania, wzmocnienie roli organu nadzoru pedagogicznego, w tym w szczególności kuratora oświaty, tak aby jak najlepiej mógł wykonywać powierzone mu ustawowo zadania. Niestety zasadnicze zmiany dotyczą wyboru dyrektora i jego pozycji w szkole lub placówce. Dyrektor szkoły jest obecnie wyłaniany w drodze konkursu. Ten organizowany jest raz na 5 lat. Komisję konkursową w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora publicznej szkoły, przedszkola lub placówki powołuje samorząd, tj. organ prowadzący. Zasiada w niej trzech przedstawicieli samorządu, trzech przedstawicieli kuratorium oświaty, po dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej, po dwóch przedstawicieli rady rodziców i po jednym przedstawicielu zakładowych organizacji związkowych. MEN proponuje zwiększenie liczby przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny w komisjach konkursowych z trzech do pięciu, z zastrzeżeniem że kuratorium może zgłosić mniejszą liczbę swoich przedstawicieli w pracach komisji, ale zawsze przysługiwać im będzie łącznie 5 głosów. Propozycja ta ośmiesza państwo polskie, wypacza ideę konkursu, nie służy odpowiedzialnej ocenie kandydatów na stanowisko dyrektora, świadczy jedynie o zamiarze centralizacji oświaty. O intencjach Ministerstwa Edukacji i Nauki świadczy propozycja zawieszania niewygodnych dyrektorów na polecenie kuratora. Planuje się m. in. wprowadzenie możliwości złożenia przez kuratora oświaty wiążącego wniosku do organu prowadzącego szkołę o zawieszenie dyrektora szkoły w pełnieniu obowiązków, chodzi o złożenie wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego. Jest też zapis dotyczący odwoływania dyrektorów. Obecnie to organ prowadzący decyduje ostatecznie o takim kroku. Po wprowadzeniu projektowanych zmian samorząd będzie głównie wykonywał wolę kuratorium oświaty w tej kwestii i cały czas płacił. Jeżeli dyrektor szkoły nie będzie realizował zaleceń organu sprawującego nadzór pedagogiczny, kurator będzie mógł wystąpić do samorządu z wnioskiem o odwołanie dyrektora w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia. Po nowelizacji ustawy - Prawo oświatowe kurator oświaty będzie miał też decydujący wpływ na zajęcia prowadzone w szkołach przez organizacje pozarządowe. Dyrektor szkoły lub placówki będzie miał obowiązek uzyskać pozytywną opinię kuratora oświaty o prowadzeniu takich zajęć. Co więcej, dyrektor będzie musiał przedstawić rodzicom lub pełnoletniemu uczniowi pełną informację o celach i treściach realizowanego programu zajęć. Udział ucznia w tych zajęciach będzie wymagał pisemnej zgody rodziców lub pełnoletniego ucznia. W efekcie dyrektorzy i nauczyciele zrezygnują z poszukiwania dodatkowych wartościowych programów wychowawczych i edukacyjnych. Aby organizacja społeczna została wpuszczona do szkoły, będzie musiała najpierw przejść trudną procedurę administracyjną. Większość dyrektorów, chcąc uniknąć kolejnych obowiązków (Dzwonek), zrezygnuje z tych zajęć z niewątpliwą szkodą dla uczniów. Proponowane zmiany to niewątpliwie prosta droga do zniszczenia lokalnej polityki oświatowej i jej obywatelskiego wymiaru. Autorzy opracowania podkreślają, że powodem wprowadzenia zmian są nieprawidłowości w funkcjonowaniu szkół. W rzeczywistości trudno spotkać sytuację, by dyrektor nie wykonywał zaleceń kontroli kuratorium, nie wpuścił przedstawicieli kuratora oświaty czy nie udostępnił dokumentacji. Jest to z całą pewnością pretekst do wywrócenia do góry nogami dotychczasowego ustroju oświatowego. Propozycja zmian w oświacie, Prawo oświatowe, jest niewątpliwie zapowiedzią przejęcia nadzoru państwa nad szkołami. Po przyjęciu projektowanych przepisów samorządowe władze lokalne będą miały niewiele do powiedzenia jako organ prowadzący publiczne szkoły. Zostanie im tylko wykonywanie zadań administracyjnych i płacenie za większość rzeczy. Szkoła samorządowa przestanie nią być, zastąpi ją szkoła scentralizowana i upaństwowiona, przychylna władzy i poddana politycznej kontroli. Zgodnie z aktualnym prawem prowadzenie szkół jest zadaniem własnym gminy. Rola samorządu sprowadza się jedynie do roli płatnika. W ostatnich latach nie pojawiła się żadna rządowa inicjatywa w polityce oświatowej budująca klimat współpracy, zaufania między organem sprawującym nadzór pedagogiczny i organem prowadzącym.

Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę teraz o zabranie głosu panią poseł Wandę Nowicką. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chciałabym wyrazić ogromny żal i oburzenie, że Prawo i Sprawiedliwość po raz kolejny zlekceważyło środowisko pielęgniarek i położnych i odrzuciło jakże słuszne postulaty płacowe tego środowiska. PiS miał okazję zachować się przyzwoicie, a zachował się jak zwykle. Rząd napluł pielęgniarkom i położnym w twarz. A jeszcze niedawno rządzący na wyścigi licytowali się, kto głośniej i dłużej będzie klaskał białemu personelowi za jego heroizm i poświęcenie w walce z pandemią. Pielęgniarki i położne zamiast oklasków wolałyby godne pensje. Dziś sejmowa większość odrzuciła opozycyjne poprawki Senatu dotyczące podwyżek dla pielęgniarek i położonych. Wstyd. Tymczasem słyszymy o kolejnych premiach i nagrodach w ministerstwach, m.in. w Ministerstwie Zdrowia, za trudną pracę w pandemii, o milionach złotych dla dyrektorów i innych nominatów partyjnych.

To jest nie tylko szczyt hipokryzji, to jest po prostu bezwstydne i haniebne. Podwyżki i wzrost finansowania powinny być pierwszym krokiem do uzdrowienia polskiego systemu ochrony zdrowia, który od lat jest na skraju załamania. Dzisiejsze głosowanie pokazuje, że rządzący, którzy przyczynili się do tego, że umieralność w Polsce ostatnio poszybowała do góry, nic sobie z tego nie robią. Nic dziwnego, oni sami nie muszą czekać na karetkę czy miejsce w szpitalu. Średnia wieku polskiej pielęgniarki to 53 lata, położonej - 50 lat. Za kilka lat to będzie 60 lat. Corocznie szkoli się 5600 pielęgniarek, pracę w zawodzie podejmuje tylko 3600 osób. Z każdym rokiem sytuacja będzie coraz bardziej dramatyczna. Polska jest w Unii Europejskiej na trzecim miejscu od końca pod względem liczby pielęgniarek na 1 tys. mieszkańców. W Polsce jest ok. 1400 karetek pogotowia.

Rząd, lekceważąc słuszne postulaty środowiska pielęgniarek i położnych, działa na szkodę całego społeczeństwa. Przepracowane pielęgniarki i luka generacyjna uderzają w jakość świadczeń medycznych, a przez to w jakość naszego zdrowia. Jak rząd może być tak ślepy, by nie dostrzegać związku pomiędzy warunkami pracy pracowników ochrony zdrowia (Dzwonek), jakością świadczeń medycznych a naszym zdrowiem i życiem? Lewica nie zostawi pielęgniarek i położnych samym sobie. Nadal będziemy walczyć o godne pensje i warunki pracy dla całego białego personelu oraz o zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia. Proszę teraz o zabranie głosu pana posła Jana Szopińskiego, Lewica. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! 5 lat temu Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało, że Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 w Bydgoszczy będą produkować wojskowe drony w opcjach rozpoznawczych i w opcjach bojowych zdolnych do zwalczania całych zgrupowań wojsk nieprzyjaciela. Jak oświadczył wiceminister obrony narodowej, dronami z Bydgoszczy zainteresowane były także inne armie świata, bo były one rewelacyjne i rewolucyjne. Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne „Belma” rozpoczęły już nawet produkcję głowic bojowych.

Tymczasem kiedy spoglądamy w niebo, to dronów pana Antoniego niestety nie widzimy. Nie widzimy ich, bo ich nie ma. Niedawno dowiedzieliśmy się, że trzeba było kupić nowe drony w Turcji, bo w Turcji były. Nie znamy też odpowiedzi na pytanie, dlaczego Ministerstwo Obrony Narodowej i polski rząd robią prezenty tureckiemu rządowi, kupując broń wartą miliardy złotych bez umowy offsetowej. Tłumaczenia o nagłych i nieznanych wcześniej zagrożeniach są dla ekspertów mało wiarygodne. Przykro mi to mówić, ale rozmawiający ze mną wojskowi uważają, że takie postępowanie polskiego Ministerstwa Obrony Narodowej wobec polskiego przemysłu zbrojeniowego to nie tylko przejaw niekompetencji, lecz także swoisty sabotaż gospodarczy, bo potencjalne miejsce Polski na światowych rynkach zapełnią producenci dronów z innych krajów świata, a polski przemysł zbrojeniowy nie będzie miał z tego tytułu żadnych korzyści technologicznych ani ekonomicznych. Bydgoscy wojskowi pytają, dlaczego ministerstwo storpedowało własny program budowy polskich dronów.

To dobre rozwiązanie dla polskiej armii, dlatego uprzejmie polecam je panu ministrowi. Apeluję także do ministra obrony narodowej, by w modernizacji polskiej armii maksymalnie wykorzystywać potencjał polskich firm, bo nie są one gorsze (Dzwonek) od firm zagranicznych.

W tej sprawie skierowałem do pana ministra obrony narodowej interpelację i oczekuję na odpowiedź. Proszę o wygłoszenie oświadczenia panią poseł Monikę Falej, Lewica. Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Dotarcie do 22 tys. uczniów i uczennic oraz gruntowne zbadanie aspektu ich bezpieczeństwa, możliwości swobodnego wyrażania siebie jest nie do przecenienia. Szkoła z założenia powinna być instytucją przyjazną uczniom, miejscem, w którym mogą zdobywać wiedzę, odkrywać swoje pasje, ale również, co ważne, być sobą. Dlatego tak ważne jest, by wskazać na te szkoły, dla których jest to priorytetem. Okazuje się, że tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi młodych ludzi jest działaniem często heroicznym. Homofobiczne wypowiedzi i działania ministra edukacji, nagonka czołowych przedstawicieli władz państwowych są niedopuszczalnym aktem łamania praw człowieka. Rzecznik praw dziecka, który dopuszcza przemoc fizyczną wobec dzieci, który odmawia młodzieży dostępu do rzetelnej wiedzy i edukacji seksualnej, to smutna rzeczywistość, w której dorastają ludzie kształtujący swoją tożsamość i określający siebie wobec świata tak wrogiego na wielu płaszczyznach. Można się spierać o miarodajność czy zasadność rozmaitych rankingów poziomu kształcenia, efektywności nauczania oraz innych mierników przekazywanej wiedzy, jednak każde badanie, które analizuje otwartość szkoły i bezpieczeństwo uczniów i uczennic w jej murach, jest pożądane i z zainteresowaniem powinno być analizowane przez wszystkich, przede wszystkim ministerstwo edukacji, kierownictwa szkół, uczniów i uczennice, ich rodziców oraz opiekunów.

Dziękuję pomysłodawcom i organizatorom projektu badającego poziom bezpieczeństwa osób LGBTQ+ w polskich szkołach, otwartości placówek i rzetelności edukacji antydyskryminacyjnej, antyprzemocowej w nich realizowanych. Takie analizy powinny prowadzić główne instytucje w kraju, np. ministerstwo czy kuratorium oświaty. Mam nadzieję, że zaczniemy budować nowe standardy edukacji w Polsce, że szkoły będą z dumą chwaliły się czołowymi miejscami w takich rankingach, a te placówki, które znalazły się na dalekich pozycjach, już dziś zaczną analizować, co można zrobić, by uczniowie (Dzwonek) i uczennice czuli się bezpiecznie, by byli akceptowani i przyjaźnie traktowani w szkole, której są częścią.

Dziękuję bardzo, pani poseł. Proszę teraz o wygłoszenie oświadczenia panią poseł Klaudię Jachirę. Panie Przewodniczący Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Kaczyński! Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Jak to jest, że z partnera USA, z którym konsultuje się najważniejsze decyzje dotyczące Europy Środkowo-Wschodniej, staliśmy się pomijanym członkiem wspólnoty? Co trzeba zrobić, żeby wielki i szanowany na arenie międzynarodowej 38-milionowy kraj stał się wstydliwym krewnym, którego strach zaprosić do stołu, bo poobraża gości? Co stało się z pozycją Polski, że prezydent Duda przyjmowany jest z honorami przez Erdogana, dyktatora łamiącego prawa człowieka, za to prezydent USA, nasz strategiczny sojusznik, co najwyżej pozwoli sobie zrobić zdjęcie w holu, spiesząc się, już nawet nie chcę myśleć dokąd. Nie oczekuję od tego rządu odpowiedzi, bo to wasza konsekwentna polityka doprowadziła do upadku prestiżu Polski i nie ma w tym przypadku. To wy narażacie na niebezpieczeństwo życie Polek i Polaków. Osłabiliście naszą armię i sojusze, podczas gdy sytuacja międzynarodowa wymaga od Polski współpracy, jedności i zaufania. Jesteście w konflikcie ze wszystkimi naszymi sąsiadami. A co będzie, gdy przyjdzie godzina próby? Spójrzcie w lustro i odpowiedzcie sobie: Kto w Europie i na świecie będzie chciał umierać za ksenofobiczną i egoistyczną Warszawę? Warszawę, która nie szanuje nawet własnych obywatelek i obywateli. Bardzo dziękuję. Nie widzę. Zatem pan poseł Tomasz Olichwer. Proszę bardzo. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! 10 czerwca tego roku grupa zrzeszająca 2300 ratowników medycznych opublikowała list otwarty, w którym zwróciła uwagę na ciężkie warunki pracy. Autorzy listu poprosili mnie o publiczne odczytanie go na obecnym posiedzeniu Sejmu, dlatego to czynię w tym punkcie z wielką przyjemnością, tym bardziej że nie tylko oni, jak pokazuje dzisiejsza demonstracja przed Sejmem pielęgniarek i położnych, są traktowani przez rząd, mówiąc kolokwialnie, po macoszemu. Przechodzę do odczytania listu: Zwracamy się do państwa z prośbą o wsparcie i przyłączenie się do niezależnej akcji zrzeszającej ponad 2300 ratowników medycznych, która promuje prozdrowotne zachowanie wśród przedstawicieli tego zawodu. Założenie tego wydarzenia opiera się na wprowadzeniu zasady: chory personel nie podejmuje dyżuru. Dla społeczeństwa takie postępowanie wydaje się oczywiste, jednak dla ludzi pracujących w państwowym ratownictwie medycznym jest to nowa jakość. Do tej pory, mając świadomość, że jest nas zbyt mało, aby w razie niedyspozycji chory personel został zastąpiony, wykonywaliśmy swoje obowiązki niezależnie od stanu zdrowia. Nasze zadania realizowaliśmy zawsze z zaangażowaniem, poświęceniem i wysoką skutecznością, choć na skutek niedogodności związanych z chorobami, skrajnym zmęczeniem bez uśmiechu na twarzy. Przez ostatni rok nasze zdrowie zostało wystawione na ciężką próbę, a praca ratownika medycznego jeszcze nigdy nie była tak ciężka. Wpłynęło to również negatywnie na psychikę personelu dodatkowo obciążoną przez działania Ministerstwa Zdrowia, które nie buduje zaufania w kwestii stabilności zatrudnienia i możliwości przeżycia z ratowniczej pensji. Cała ta sytuacja bardzo osłabia morale ratowników medycznych. W związku z powyższym ratownicy medyczni podjęli decyzję, że w pierwszym tygodniu sierpnia konsultować się będą z psychiatrami, aby dokonać redukcji szkód w swoich osobowościach i ratować zgliszcza, które pozostały z ich rodzinnych egzystencji. Powstaje obawa, że konsultacje z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarzami psychiatrii wpłyną na dyżurową frekwencję oraz ograniczą dostępne zespoły ratownictwa medycznego, zespoły transportu medycznego, obsady szpitalnych oddziałów ratunkowych oraz innych miejsc, gdzie pracują ratownicy medyczni. Istnieje taka możliwość, ale z uwagi na brak szacunku do naszego zdrowia jako osób stanowiących filar ratownictwa medycznego w Polsce ze strony Ministerstwa Zdrowia musimy sami zacząć o nie dbać. Nie do pominięcia jest fakt, że akcja nie ma na celu (Dzwonek) wywołania konfliktu naszego środowiska z Ministerstwem Zdrowia, a jedynie jest to akcja profilaktyki zdrowotnej wśród ratowników medycznych. Więcej informacji na naszym facebookowym profilu „Ratownicy Medyczni. Proszę teraz pana posła Dariusza Olszewskiego o wygłoszenie oświadczenia. Szanowny Panie Marszałku! Stojąc w siedzibie polskiego parlamentu, pragnę przypomnieć o bardzo istotnych wydarzeniach zapisanych na kartach polskiej historii. 28 czerwca 1919 r. w Sali Lustrzanej Pałacu Wersalskiego podpisano traktat pokojowy z Niemcami będący fundamentem nowego porządku w Europie po zakończeniu I wojny światowej. W imieniu Polski traktat podpisali Ignacy Paderewski, ówczesny polski premier, oraz Roman Dmowski, najbardziej znany na Zachodzie polski polityk. 31 lipca 1919 r. Sejm Ustawodawczy Rzeczypospolitej po burzliwej debacie ratyfikował traktat pokojowy z Niemcami. Ostateczny bilans traktatu wersalskiego był wielkim zwycięstwem Polski, efektem zabiegów dyplomatycznych Józefa Piłsudskiego, Jana Paderewskiego i Romana Dmowskiego. Polska formalnie powróciła na mapę Europy, otrzymała swobodny dostęp do morza oraz znalazła się w gronie zwycięzców I wojny światowej. Marzenia wielu stały się faktem. Dążenia ojców niepodległości przyniosły pożądany skutek.

Fakt ten najlepiej dowodzi, iż Polska jest i będzie najsilniejsza, kiedy najistotniejsze sprawy Polacy będą realizować wspólnie, razem, bez oglądania się na podziały czy wizje. Kłótnie i swary nigdy nie przynosiły i nie przyniosą nikomu nic dobrego. Nie służą one budowaniu silnego, bezpiecznego i bogatego państwa. One tylko mogą w tym przeszkodzić i zniszczyć to, co zostało już osiągnięte. Marszałek Józef Piłsudski mówił: „Idźcie swoją drogą, służąc jedynie Polsce, miłując tylko Polskę i nienawidząc tych, co służą obcym” Dziękuję bardzo. Oświadczenie teraz wygłosi pan poseł Janusz Korwin-Mikke, Konfederacja. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Niestety posłanka Jachira miała dużo racji. Polityka zagraniczna naszego państwa postawiła nas w sytuacji dramatycznej.

Udało się nam zadrzeć z Czechami. I udało się nam zadrzeć w tej chwili ze Stanami Zjednoczonymi, które dziwnym trafem nie chcą iść na pasku polskiej polityki. Ewentualnie możemy mówić także o Szwecji, ale to też i potop, i będziemy z nią grali za parę dni i też może być bardzo niedobrze. Tak że, proszę państwa, zadarliśmy ze wszystkimi. Z Francją również mamy stosunki nie najlepsze, z Wielką Brytanią także. Powstaje pytanie, czy Wyszehrad, który też się z nami nie zgadza w sprawie polityki rosyjskiej. Tak że powtarzam: zostaliśmy sami. Zostaliśmy sami i trzeba dokonać zasadniczej reorientacji polskiej polityki zagranicznej, bo nie chciałbym znaleźć się w sytuacji, kiedy zostanie dokonany kolejny rozbiór Polski, tym bardziej, że - jak by to powiedzieć - armia polska opiera się na dwóch brygadach głównie kawalerii amerykańskiej.

Tak że, proszę państwa, wzywam rząd, żeby tę sprawę przemyślał.

Dziękuję bardzo, panie pośle.

Szanowny Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Na wstępie chciałam podzielić swoje oświadczenie na dwie części. Po pierwsze to, o czym mówiła pani poseł Wanda Nowicka w zakresie podwyżek dla pracowników ochrony zdrowia. Głosowaliśmy nad tym w Sejmie, jak również akceptowaliśmy poprawki Senatu w zakresie podwyższenia wynagrodzeń pracownikom ochrony zdrowia. Za swoją ciężką pracę powinni otrzymywać godne wynagrodzenie. A teraz drugie moje oświadczenie.

Mieczysława Karłowicza w Mielcu ma bogatą historię.

To podziękowania za pracę, za to, że nauczyli młodych ludzi kochać muzykę, za to, że stworzyli tak wspaniałe miejsce, które promieniuje na życie kulturalne miasta Mielca, jako że uczniowie tej szkoły i nauczyciele biorą udział w ok. 100 wydarzeniach kulturalnych miasta, tj. koncertach, recitalach, audycjach muzycznych i wielu innych wydarzeniach artystycznych. To właśnie tam uczniowie mogą realizować swoją pasję. Za tę atmosferę, za to szczególne miejsce, w którym słychać muzykę.

Raz jeszcze moje gratulacje i słowa mojego najwyższego uznania dla wszystkich, którzy przyczynili się do wieloletniego funkcjonowania tej placówki.

Myślę, Wysoka Izbo, że wszyscy dołączymy się do gratulacji dla zacnej Alma Mater. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! To niezwykła okazja do wszelkiego rodzaju podsumowań, analiz, ocen i podziękowań. Społeczna praca ludzka ma wymiar o wiele większy niż tylko kronikarski zapis. W okresie tych 40 lat byli żołnierze wykonywali kapitalną pracę patriotyczną w swoich rejonach oddziaływania. Przekazywali licznym pokoleniom młodzieży prawdę historyczną, której dziś tak bardzo im brakuje. Bliskie kontakty z samorządowcami pokazały, jak ważną rolę odgrywają w lokalnej społeczności. Byli żołnierze spełniają także ważną funkcję dla swojego wewnętrznego środowiska, niosąc pomoc potrzebującym, podtrzymując kontakty koleżeńskie i rodzinne, by wreszcie oddawać hołd ostatniego pożegnania odchodzącym na wieczną wartę. Ona jest darem serca dla Polski. Przez te lata różny był stosunek władz do działalności byłych żołnierzy. Nigdy nie był łatwy. Mimo wszystko związek skupiał dziesiątki tysięcy członków. Bliskie kontakty z miejscem dawnej służby obfitowały licznymi przyjacielskimi kontaktami, które materializowały się dla funkcjonowania związku w jednostkach oraz instytucjach wojskowych. Byli żołnierze czuli się zawsze związani ze swoimi macierzystymi jednostkami. Niestety okres transformacji ustrojowej położył się cieniem na tych doskonałych relacjach. Każda władza po 1990 r. dołożyła swoją cegiełkę do upadku znaczenia więzi międzypokoleniowej. Nowe wolnościowe władze zaprowadziły swój porządek prawny, którego efekty odczuwa naród po dzień dzisiejszy. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że ludzie wierzą w swój zbawienny dla narodu kierunek działania. Dopiero dziś, w dobie narodowego kryzysu, dostrzegają pilną potrzebę wzmacniania armii, którą tak bezmyślnie roztrwoniono wraz z jej majątkiem. Tego naród nie powinien nikomu wybaczyć. Dziś wystarczy być politycznie poprawnym w kategoriach wytyczanych przez władze.

Kto obniżył emerytom emeryturę o 25%? Kto pozbawił ich wojskowych asyst honorowych przy obchodach różnych świąt, rocznic czy pogrzebów?

Szanowni Państwo! Dzisiaj dziękujemy. Dziękujemy za to, co zrobiliście, i pamiętamy o waszej dewizie: zawsze wierni. Dziękuję bardzo panu posłowi. Jako ostatni oświadczenie wygłosi pan poseł Artur Dziambor. Chociaż audytorium nie za tęgie, to obiecujemy, że będziemy uważnie słuchali pana posła i jego oświadczenia. Wysoka Izbo! Jak zapewne wszyscy wiecie, Konfederacja sprzeciwia się wszelkiej maści rozdawnictwu publicznych pieniędzy, jednak w sytuacji, w której kolejne rządy są w stanie wydawać miliardy złotych na różne programy pomocowe, wsparcie socjalne itp., nie jesteśmy w stanie zrozumieć, że nie chcą zająć się stosunkowo niewielkim wsparciem dla osób najbardziej potrzebujących, jakimi są np. opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych. Ta niezbyt liczna grupa domaga się sprawiedliwego traktowania i swoją nierówną walkę z bezdusznym aparatem państwa prowadzi już siódmy rok, a więc drugą z rzędu kadencję tzw. Zjednoczonej tzw. Prawicy, która z ustami pełnymi frazesów o polityce prorodzinnej nadal nie pochyliła się nad najbardziej potrzebującymi: starszymi osobami, emerytami, którzy już niejednokrotnie sami wymagają opieki i leczenia, a mimo to nadal sprawują opiekę nad swoimi ciężko chorymi, niepełnosprawnymi dziećmi. Ci ludzie są traktowani skrajnie niesprawiedliwie i są jawnie dyskryminowani. Oni musieli przepracować zawodowo co najmniej 20 lat, aby nabyć prawa do wcześniejszej emerytury, która jest teraz na poziomie ok. 1200 zł, a osoby nabywające aktualnie prawo do świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości ok. 2000 zł nie muszą wykazać się żadnym stażem pracy i mają jeszcze opłacane składki emerytalne. Projekt nowelizacji ustawy dotyczący świadczenia wyrównującego do wysokości świadczenia pielęgnacyjnego, druk nr 745, leży w Sejmie od października zeszłego roku i jest to niebywały skandal, że nie został jeszcze wniesiony pod obrady i przegłosowany, zwłaszcza że dotyczy stosunkowo niewielkiej liczby osób, ok. 25 tys. ludzi. Ci państwo byli ze mną, z nami na konferencji prasowej w ubiegłym tygodniu tutaj, w Sejmie, dać swoje świadectwo. W ich sprawie złożyłem też stosowną interpelację i mam nadzieję, że sprawa ta zostanie wskrzeszona w tej Izbie jak najszybciej. Wnoszę o jak najszybsze zajęcie się tą bulwersującą sprawą, ponieważ, szanowni państwo z Prawa i Sprawiedliwości głównie i pani minister rodziny i polityki społecznej, skoro potraficie wolną ręką wydać 2 mld zł na Telewizję Polską, wydawać miliony na wybory, które się nie odbyły, na trefne maseczki, na loterię szczepionkową, na premie dla urzędników, na wszelkiej maści propagandowe programy z plusem, które w rzeczywistości, jak wiemy, bardzo często są minusami, to nie jest absolutnie do pojęcia to, że nie potraficie albo nie chcecie zająć się sprawiedliwym traktowaniem najbardziej potrzebujących ludzi, którzy nie mają do kogo się zgłosić, a jedyne, co im pozostało, to żebrać. Musicie się tym zająć. Jako państwo macie obowiązek zajmować się właśnie takimi ludźmi. To nie są masowi wyborcy, ale to są ludzie, którymi powinno się zajmować państwo prorodzinne, opiekuńcze, a nie zajmuje się niestety. Czas to zmienić. Bardzo dziękuję panu posłowi.